po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu, a w przypadku sprawozdania z druku nr 3591 zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusjach nad tymi punktami porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22. porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Przypominam, że postawienie pytania nie może trwać dłużej niż 2 minuty, zaś udzielenie odpowiedzi nie może trwać dłużej niż 6 minut. Prawo do postawienia pytania dodatkowego przysługuje wyłącznie posłowi zadającemu pytanie. Dodatkowe pytanie nie może trwać dłużej niż 1 minutę, a uzupełniająca odpowiedź nie może trwać dłużej niż 3 minuty. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Jako pierwsi pytanie zadają posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Zbigniew Chmielowiec i Mariusz Trepka z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę o zadanie pytania. Panie Ministrze! 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” Na realizację programu została przeznaczona kwota ponad 9 mld zł, z czego ponad 500 mln zł zagwarantowano na unowocześnienie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Nowy sposób podziału środków wzbudzał niezadowolenie przedstawicieli Zarządu Głównego OSP, a w przestrzeni medialnej pojawiały się nieprawdziwe informacje, jakoby nowa formuła dofinansowania miała prowadzić wręcz do likwidacji jednostek ochotniczych straży pożarnych. Te informacje początkowo wzbudzały niepokój druhów OSP w terenie. Szybko się okazało, że zgodnie z założeniami nowy system miał na celu optymalizację i zapewnienie transparentności podziału środków finansowych dla ochotniczych straży pożarnych. Pieniądze zaczęły trafiać do tych jednostek, które wcześniej nie mogły liczyć na dofinansowanie. Panie Ministrze! Trzeci rok funkcjonowania programu i nowej formuły przyznawania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych to dobry moment na podsumowanie. Dlatego uprzejmie proszę pana ministra o odpowiedź na pytania, w jakiej wysokości środki finansowe zostały dotychczas przekazane ochotniczym strażom pożarnym, na jakiego rodzaju zadania, w jaki sprzęt doposażono jednostki OSP, w tym ile samochodów ratowniczo-gaśniczych przekazano. Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego. Proszę, panie ministrze. Wysoki Sejmie!

W Polsce w ciągu roku występuje ponad 500 tys. zdarzeń, do których spieszą strażacy zawodowi bądź ochotnicy albo razem. Łatwo przeliczyć, że co minutę ktoś w Polsce potrzebuje ich pomocy.

A więc dbamy o te oba płuca jednakowo, bo one są jednakowo potrzebne i działając razem, zapewniają bezpieczeństwo Polakom w najróżniejszych sytuacjach, w sytuacjach różnych opresji. Bo przecież dzisiaj są to nie tylko pożary, ale także najróżniejsze inne tzw. miejscowe zagrożenia, wypadki komunikacyjne, działania sił przyrody, zagrożenia cywilizacyjne, techniczne - chodzi o różne sytuacje. I dzisiaj straż pożarna na wszystkie reaguje. Jest to najbardziej wielofunkcyjna spośród wszystkich służb. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wszystkich szczebli - razem dbamy o to, żeby wesprzeć strażaków ochotników i wzmocnić ich potencjał, tak by mogli skutecznie reagować na wszystkie zagrożenia.

Są także przeznaczane na zakup sprzętu informatyki i łączności: radiotelefonów nasobnych, systemów selektywnego alarmowania, syren alarmowych, zestawów podhełmowych do radiotelefonów, ładowarek do telefonów itd., a także na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego, a również wspieraniu inwestycji i remontów obiektów służących druhom ochotnikom. Chciałbym w tym miejscu, korzystając z okazji, jak najserdeczniej podziękować wszystkim strażakom ochotnikom, a jest ich w Polsce bardzo dużo. To jest w ogóle nasza polska, piękna specyfika. Ponad 100 tys. strażaków ochotników z jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i kilkaset tysięcy innych strażaków działających w pozostałych jednostkach OSP w tych ponad 16 tys. jednostek w Polsce. Wyrażam naprawdę wielką wdzięczność za ich ofiarność, za ich profesjonalizm, bo przecież jednostki i strażacy coraz bardziej się profesjonalizują, bo tego wymagają dzisiejsza sytuacja, charakter dzisiejszych zagrożeń i konieczność współdziałania specjalistycznego ze strażą zawodową. Chcę też podkreślić, że strażacy ochotnicy oprócz podstawowej działalności spełniają także bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o działania integracyjne, jeżeli chodzi o społeczność lokalną, działania z dziedziny kultury.

Zasługują na wielki szacunek i wielkie uznanie, dlatego wspieramy ich i będziemy wspierać, zwiększając nakłady. Między 2015 r. a 2018 r. zwiększyliśmy dofinansowanie z budżetu państwa o ponad 30% dla druhów ochotników.

Do tego doszło jeszcze wsparcie z innych resortów. Minister sprawiedliwości w ubiegłym roku wsparł druhów ochotników - przeprowadziliśmy ten proces wspólnie, ale to były pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości - kwotą ponad 100 mln zł. Dziękuję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze za wsparcie strażaków, za współdziałanie w tym zakresie.

Będzie to 480 samochodów w tym roku właśnie dzięki też życzliwości, dobrej współpracy z Ministerstwem Środowiska i podległymi mu instytucjami. Dziękuję także - już ostatnie zdanie w tej części, panie marszałku - chcę podziękować samorządom, bo ich wkład w zakup każdego samochodu także jest bardzo istotny. Panie Marszałku! Panie Komendancie! Bardzo serdecznie dziękujemy za tę pomoc. My, posłowie, jesteśmy również bardzo wdzięczni druhom i druhnom z ochotniczych straży pożarnych, bo właściwie na co dzień przyglądamy się ich pracy, jesteśmy blisko ich działań i widzimy, jak to się odbywa, jak to się dzieje, jak wielkie mają ambicje, jak są bardzo zdeterminowani, aby nieść pomoc innym, i jak świetnie potrafią integrować społeczeństwo, w którym działają. Chciałam zadać takie pytanie: Czy znowelizowany system dystrybucji środków finansowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych przyczynił się do zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i lepszych warunków pełnienia służby?

Dziękuję bardzo. W 2016 r. wprowadziliśmy te nowe zasady dofinansowywania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jakoś nie zniszczyliśmy, tylko wręcz przeciwnie - te jednostki są wzmacniane, ich potencjał jest coraz większy, a co najważniejsze, proszę państwa, budujemy poprzez ten jednolity system dofinansowywania spójny system ratowniczo-gaśniczy. Obecny na sali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i zarazem szef Obrony Cywilnej Kraju dysponuje tymi środkami i on widzi w całości te potrzeby w skali kraju, poszczególnych województw, poszczególnych powiatów, bo wnioskują o to oczywiście komendanci powiatowi w konsultacjach z jednostkami OSP poszczególnych szczebli, z ich organizacjami, bo to przecież są stowarzyszenia szczebla powiatowego, wojewódzkiego, wnioskują poprzez komendantów wojewódzkich i pan komendant główny oczywiście uwzględnia hierarchizację tych potrzeb, które są zgłaszane i są formułowane w powiatach i województwach. Tak że to się dzieje w konsultacji i ze strażakami zrzeszonymi na różnych szczeblach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, i z komendantami państwowymi, powiatowymi, miejskimi, wojewódzkimi, bo oni widzą te potrzeby bliżej. To wszystko naprawdę dobrze wygląda. Przy wzmocnieniu środków finansowych, przy takim coraz większym finansowaniu jednostek OSP z różnych źródeł, jak słyszymy, i przy właśnie tej jednolitości traktowania, nie kto bliżej, kto szybciej, tylko kto bardziej potrzebuje, kto jest bardziej potrzebny do akcji ratowniczo-gaśniczych, do działań, do których jest przeznaczona straż pożarna, ten otrzymuje wsparcie. Właśnie takim prawem, że one spełniają niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa i komendant musi wiedzieć, które czego potrzebują, które mają jaki potencjał i jakiego rodzaju działań potrzebują dla wzmocnienia.

Zresztą słyszę, otrzymuję też korespondencję z różnych stron, z różnych miejsc w kraju, że jest naprawdę akceptacja dla tych rozwiązań. Będziemy też przekazywać samochody.

To też jest zastrzyk, też jest zasilenie oprócz zakupu tych nowych samochodów. Naprawdę, szanowni państwo, nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie ma czasu, ale na te pytania, które pojawiły się odnośnie do poszczególnych województw, przekażę odpowiedź na piśmie. Jestem na to przygotowany, ale nie ma czasu. Chcę jeszcze zaznaczyć, że wszystkie województwa, wszystkie powiaty, wszystkie gminy i wszystkie jednostki OSP otrzymują na koniec roku czy na początku następnego roku po podsumowaniu dokładną informację o finansowaniu jednostek OSP w skali kraju, w skali województwa, w skali powiatu, gminy i dla poszczególnych jednostek, więc to jest transparentne. Tego nigdy nie było, bo wcześniej Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nawet nie dawał sprawozdań komendantowi głównemu, więc on nie wiedział, gdzie te pieniądze idą. Kolejne pytanie zadają posłanki Izabela Leszczyna i Halina Rozpondek, klub Platformy Obywatelskiej.

Wysoki Sejmie! Panie Premierze! Od 2016 r. premier Morawiecki i rząd PiS-u nacjonalizują banki, zapewniając, że to jest działanie pozytywne, bo państwowe banki są bezpieczne i przyjazne dla obywateli. To kłamstwo. Usługi bankowe są coraz droższe, zyski banków coraz wyższe, a banki państwowe rzeczywiście chętnie udzielają kredytów, ale prezesowi Kaczyńskiemu na budowanie dwóch wież w Warszawie, a nie na ratowanie miejsc pracy w Częstochowie. Dramatyczna sytuacja w częstochowskiej hucie trwa od maja. Od maja huta nie pracuje, pracownicy są na urlopach albo na tzw. postojowym, tzn. dostają niższe pensje. Dlaczego? Bo te państwowe, podobno przyjazne dla obywateli banki nie chciały udzielić kredytu funduszowi, który chce przejąć hutę za długi od obecnych właścicieli. Od 2 miesięcy hutnicy proszą o pomoc premiera, rząd i nic - cisza. Musiało 200 hutników zdesperowanych wizją utraty miejsc pracy przyjechać do Warszawy, pikietować pod bankiem, żeby prezes banku wyszedł i powiedział, że wróci do negocjacji. Gdyby huta upadła, to koszty społeczne będą następujące: oprócz ponad 1200 pracowników to jest 5 tys. miejsc pracy wokół huty. Panie Premierze! Oczekuję odpowiedzi tu, z mównicy sejmowej - że rząd będzie gwarantem tego, że negocjacje będą szybkie i skuteczne, że zakończą się do 10 lipca, że prezes banku wystraszony przez hutników nie wycofa się z tych negocjacji i że nie będzie tak, iż obietnica, jaką złożyliście wczoraj hutnikom, będzie taką obietnicą jak ta, którą daliście częstochowianom, że powstanie województwo częstochowskie, na które od 4 lat czekają bezskutecznie. Dziękuję bardzo. Odpowiedzi z upoważnienia prezesa Rady Ministrów udzieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pan Marek Niedużak. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Ja, prawdę mówiąc, jestem teraz troszeczkę w kropce, ponieważ te pytania, które zostały przedstawione na piśmie, całkowicie nie korespondują z tymi, które teraz zostały zadane. Zacznijmy.

Był to kapitał ukraiński z Donbasu, wydaje się, że obecnie jest to także kapitał rosyjski. W związku z tym szczegółowe informacje na temat sytuacji huty siłą rzeczy nie są nam znane - nie są, ponieważ nie jesteśmy jej właścicielami. Mamy tylko takie informacje, które są w domenie publicznej, które są w sferze publicznej, w mediach, również od związkowców.

Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie z tych przedłożonych na piśmie: „Dlaczego duże polskie banki nie współpracują ze sobą w celu ratowania huty?”, powiem w ten sposób: znowuż proszę pamiętać, że to są banki - pomimo że rzeczywiście w obu tych bankach ma udziały Skarb Państwa, są to jednak spółki akcyjne, publiczne, notowane na giełdzie, instytucje zaufania publicznego, które muszą działać w oparciu o przepisy Prawa bankowego, w oparciu o przepisy k.s.h.

Ten kapitał jest od ludzi, którzy trzymają swoje pieniądze na depozytach w tych bankach. W związku z tym nie możemy oczekiwać od nich, że oni będą, powiedzmy, podejmowali decyzje jakby w całkowitym oderwaniu od ryzyk związanych z daną sytuacją.

Znowuż - ja tutaj też się mogę odwołać tylko do informacji, które są w przestrzeni publicznej. Chciałbym więc zwrócić uwagę, że ten fundusz brytyjski, jeśli popatrzeć na dostępną w sferze medialnej, publicznej historię jego działania, to jest to też fundusz, który głównie inwestuje np. w aktywa w Wielkiej Brytanii, właśnie hutnicze, ale też raczej po to, by je likwidować, a niekoniecznie po to, aby je restrukturyzować.

Natomiast, tak jak powiedziałem, z tego, co mi wiadomo, jest komunikacja pomiędzy związkowcami, pracownikami a bankami.

Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Naszym dzisiejszym obradom przysłuchuje się delegacja Komitetu Rozwoju Społecznego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych z przewodniczącym komitetu panem He Yiting na czele, która przebywa w Polsce na zaproszenie przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Serdecznie witamy naszych gości. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pan Marek Niedużak. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Poseł! Powiem tak: ja jestem prawnikiem. Żadna moja wypowiedź nie ma w tym momencie jakiegokolwiek wpływu na zobowiązania prawne banku i vice versa.

Banki są wierzycielami. Z tego, co mi wiadomo, nie są jedynymi wierzycielami, bo jest jeszcze jakiś wierzyciel zagraniczny. To jest niezwykle skomplikowana.

Jest to niezwykle skomplikowana transakcja obciążona bardzo dużym ryzykiem.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Kolejne pytanie zadają posłowie Waldemar Andzel, Urszula Rusecka, Andrzej Gawron i Anna Kwiecień z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Jest to pytanie w sprawie kryteriów, jakie będą obowiązywały przy wypłacie świadczenia na pierwsze dziecko. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Program 500+ jest przełomowym programem wsparcia dla rodzin.

Jest możliwość składania wniosków, żeby ta wyplata była też na pierwsze dziecko. Prosiłbym pana ministra o taką informację bieżącą, ile tych wniosków już spłynęło. W tej chwili wiemy, że jest możliwość składania wniosków przez Internet. Jest to duży program, który obejmuje kilka milionów dzieci.

Czy pan minister ma takie informacje, czy pieniążki już zostały przelane na konta samorządów? Kiedy praktycznie pieniądze zostaną wypłacone?

Dziękuję bardzo. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie, bo ono jest jak najbardziej na czasie.

Wskaźniki ubóstwa.

No i inwestycja w kapitał ludzki.

I teraz to, o co pan zapytał, jeśli chodzi o realizację.

Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo!

Jest to na pewno przełomowy, historyczny program, którego dotąd w naszym kraju nie było. Na pewno macie państwo już dane w ministerstwie.

Ile jest takich rodzin, jak samorządy to monitorują i czy te przewidywania opozycji się sprawdziły? Dziękuję. Ponownie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Wysoka Izbo!

Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, że pierwsze wypłaty z programu 500+ już nastąpiły w nocy.

I sukcesywnie te środki są przekazywane. Środki są na kontach w poszczególnych gminach, wojewodowie przekazują je w transzach, tak że nie ma żadnego zagrożenia.

Jeśli chodzi o pytanie pani poseł, to oczywiście te prognozy absolutnie się nie potwierdziły.

Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pan poseł Paweł Skutecki z klubu Kukiz’15 zadaje pytanie w sprawie orzeczenia śmierci 11-miesięcznego Szymona w szpitalu przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Przebywał w tym szpitalu od blisko pół roku.

Natomiast ta sytuacja wzburzyła opinię publiczną na tyle, że pojawiły się bardzo poważne pytania, na które rząd dotychczas nie odpowiedział. Ja bym chciał usłyszeć te odpowiedzi od pana ministra dzisiaj.

Czy pan minister nie uważa, że należałoby ten aspekt w jakiś sposób unormować, żeby do takich sytuacji w przyszłości już nie dochodziło? Panie Ministrze! Czy rząd planuje debatę nad temat tzw. śmierci mózgowej, którą wielu lekarzy i specjalistów, m.in. bardzo znany prof. Talar, uznaje za jeden z największych medycznych mitów nowożytnych czasów? Wreszcie, panie ministrze, w ogóle w polskim prawie nie jest unormowane coś, co się nazywa uporczywą terapią, a semantycznie jest to sprawa bardzo bliska kwestii eutanazji, odbierania życia. Czy ministerstwo planuje jakiekolwiek prawne unormowania w sprawie tzw. terapii uporczywej? Dziękuję.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za te pytania. Art. 43 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jednoznacznie stwierdza, w jaki sposób lekarz orzeka o stwierdzeniu zgonu, a w kwestii stwierdzania tzw. śmierci mózgu są ramowe wytyczne dotyczące postępowania, które jednoznacznie wskazują, w jaki sposób należy to zrobić. Warto, nie wchodząc w szczegóły, wskazać, że postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe. Pierwszym etapem jest wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu, a drugim wykonanie badań potwierdzających tę śmierć. I tutaj nie ma mowy o tym, żeby te sprawy w jakikolwiek sposób pozostawić przypadkowi.

Szanowni państwo, ono zmarło po prawie 6-miesięcznej batalii, którą stoczyli lekarze, pielęgniarki, personel medyczny szpitala przy ul. Niekłańskiej.

Szanowni Państwo! Warto porozmawiać o faktach. Następnego dnia była ona już w szpitalu.

Jak wszyscy państwo wiecie, absolutnie nie ma możliwości, żeby z mównicy sejmowej omawiać szczegóły tej kontroli i omawiać szczegóły dotyczące stanu pacjenta.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Panie ministrze, proszę o jednoznaczną, krótką odpowiedź na pytanie, czy w związku ze sprawą tego chłopca został zgłoszony niepożądany odczyn poszczepienny.

A teraz ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Janusz Cieszyński. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Tak jak wspominałem w mojej poprzedniej wypowiedzi - wydaje mi się, że to powinno być oczywiste dla każdego z nas, bo wielu z nas jest pacjentami, członkowie naszych rodzin są pacjentami - panie pośle, nie będziemy udzielali jakichkolwiek informacji na temat spraw związanych ze stanem zdrowia i życia tego konkretnego pacjenta. Nie będziemy udzielali informacji o procedurach, które zostały wykonane. To są bardzo intymne sprawy, które pozostają do wyłącznej wiadomości lekarzy oraz rodziny pacjenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Posłowie Mirosław Maliszewski, Mieczysław Kasprzak, Jan Łopata i Krzysztof Paszyk zadają pytanie w sprawie niedoboru wody. Pytanie zadaje pan poseł Jan Łopata. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Długotrwałe susze, które tu występują, uwidoczniły jak w soczewce systemowe braki i problemy z brakiem wody.

Sytuacja jest tragiczna, coraz częściej brakuje wody również w kranach u Polaków, a także w każdej sferze produkcji. Problemy dotyczą przede wszystkim rolnictwa, ale także energetyki czy przemysłu. Rolnictwo szczególnie odczuwa brak aktywności rządu w zakresie systemu melioracji czy retencji. Jeśli w najbliższej przyszłości nie spadną długotrwałe deszcze, susza zabije polskie rolnictwo. Kiedy ruszy budowa małych zbiorników retencyjnych? Wiele stawów w obrębie gospodarstw zostało wykopanych przed laty, gdy nie było wymaganych zezwoleń wodnoprawnych. Co teraz należy zrobić, by legalnie z nich korzystać? Jak wygląda procedura legalizacji? W jaki sposób będą naliczane opłaty za korzystanie z wody wydobytej z takiego stawu [[Dzwonek]] i na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy dotknięci skutkami suszy? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Na pytanie odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście dotyczy ono kwestii poważnej: jak gospodarować wodą, której jest coraz mniej. Mówi pan o systemowych brakach w systemach melioracji i retencji, więc rozumiem, że tu jest uderzenie się w piersi również za lata, kiedy odpowiadaliście w Polsce i centralnej, i regionalnej za gospodarkę wodną. Jeżeli tak pan to traktuje i jest to rzeczywiście przyznanie się do zaniedbań wieloletnich, to dziękuję, bo faktycznie próbujemy naprawić to, co przez lata zostało zaniedbane.

Dane o dostępności wody, na które pan się powołuje, są generalnie poprawne, chociaż wydaje mi się, że jeśli chodzi o powoływanie się np. na dane instytucji, która została wymieniona w tekście, która m.in. była jedną z organizacji bardzo utrudniających zwalczanie afrykańskiego pomoru świń w Polsce, na którym poległ jeden z pana kolegów ministrów rolnictwa, to wolałbym się na te dane nie powoływać.

więc ten problem występuje od dawna i nic w tej materii przez lata nie uczyniono. Próbujemy ten problem rozwiązać i szybko przedstawię, jakie działania podjęliśmy. Od sierpnia - mam nadzieję, że opóźnienia nie będzie, a jeżeli wystąpi, to może w bardzo krótkim czasie - uruchamiamy program dofinansowania inwestycji związanych z nawadnianiem w gospodarstwach rolnych. Będzie to dotyczyło wykonania nowego nawadniania, łącznie z wykonaniem ujęcia wody z wód podziemnych lub powierzchniowych, modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej, ewentualnie z modernizacją ujęcia wody i modernizacji instalacji nawadniającej z powiększeniem obszaru. Chodzi o to, żeby rolnikom, którzy w szczególności uprawiają rośliny bardzo intensywne, dać możliwość nawodnień, chociaż zdaję sobie sprawę, że bardzo ważne jest nie tylko dostarczenie wody, ale i zwiększenie chłonności i pojemności wodnej gleb w Polsce.

Jeżeli ktoś chce rozszerzyć ten zbiornik wodny, to musi sprawdzić, czy nie pozostaje to w kolizji z obowiązującym prawem.

Opóźnienie we wprowadzeniu tej ustawy wynikające ze strachu przed wprowadzeniem nawet symbolicznych opłat za wodę powodowało, że Polska była zagrożona ogromnymi karami i utratą kilkunastu miliardów złotych z pieniędzy unijnych.

Ale chcę przypomnieć, że pobór wody powierzchniowej do nawodnień rolniczych jest zwolniony z jakichkolwiek opłat, również nie ma opłat stałych. Stawki, które w tej chwili obowiązują, są niższe niż w latach minionych, więc to są absolutnie symboliczne stawki dla rolników, którzy będą się decydowali na korzystanie z wód podziemnych. Sprawa suszy.

Zbliżają się żniwa i chodzi o to, by to oszacować. Sprawa naprawy istniejących systemów melioracyjnych. Pan zadał pytanie o to, kiedy zostanie wprowadzony rządowy program rozwoju melioracji wodnych. Najpierw trzeba naprawić to, co istnieje, co zostało zdewastowane, również przez lata zaniedbań. Zwiększyliśmy dofinansowanie pojedynczej spółki wodnej lub związku spółek z 500 tys. do 1 mln.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wbrew pozorom nie rozczarował mnie pan.

Przecież to nie o to chodzi. Problem jest? Myślę, że jest to jeden z wielu tematów, nad którymi wszyscy powinniśmy się pochylić, bo problem deficytu wody w Polsce, i nie tylko w Polsce, narasta. I dobrze by było, gdybyśmy rozmawiali i nie licytowali się, tylko mówili o problemach i programach i wspierali się wzajemnie. Tak myślę. Dziękuję za odpowiedź. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Panie Pośle! Pan mówi o systemowych brakach, pan mówi o tym, że rząd się chwali, że trzeba działać natychmiast, już, a nie czekać 2 lata.

Rzeczywiście, ma pan rację, liczę na pomoc również ze strony pana i pana formacji. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania.

Bardzo proszę, pierwsze pytanie zadaje pan poseł Lech Kołakowski. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia, z którego mają korzystać mieszkańcy polskiej wsi. Pomoc finansowa ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwoju gospodarstw rolnych, modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych, przeznaczanie premii dla młodych rolników, płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Z informacji przekazanych przez mieszkańców wsi wynika, że środki kierowane na pomoc finansową dla rolników trafiają przede wszystkim do dużych gospodarstw rolnych. Wiele z nich z pomocy takiej skorzystało wielokrotnie, co umożliwiło ich dynamiczny rozwój. Inaczej przedstawia się sytuacja małych i średnich gospodarstw rolnych, które dominują w Polsce, w tym w województwie podlaskim, którego jestem reprezentantem. Od lat nasz region boryka się z problemami emigracji, który dotyczy zwłaszcza młodych ludzi, i starzenia się społeczeństwa. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, aby zapobiec depopulacji regionu. Polska należy do najsilniejszych państw w Europie pod względem rolnictwa. Województwo podlaskie ze swym nieskażonym środowiskiem winno stać się najsilniejszym w kraju i Europie regionem rolnictwa rodzinnego i ekologicznego. Pytania: Jakie działanie podejmie ministerstwo na rzecz wsparcia małych i średnich gospodarstw w Polsce w najbliższych latach w zakresie pomocy rozwojowej oraz zwiększenia możliwości rozwoju produkcji w tych gospodarstwach? Z jakich środków mogą skorzystać małe i średnie gospodarstwa rolne i jakie zmiany w tym zakresie proponuje ministerstwo w kolejnej perspektywie finansowej? Pragnę też podziękować panu ministrowi i rządowi za wsparcie polskiej wsi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie. Ono zresztą mieści się w pewnym szerszym kontekście dotyczącym wspierania w Polsce również mniejszych i średnich gospodarstw rolnych, ważnych nie tylko z powodów ekonomicznych, produkcji żywności czy nieżywnościowych surowców, ale również dla utrzymywania żywotności społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich. Rola tych gospodarstw jest nie do przecenienia, bo od tego, czy takie gospodarstwa, uzyskując część swoich dochodów z produkcji rolniczej, część zapewne z innych źródeł, będą istniały, zależy również utrzymywanie żywotności, utrzymanie usług publicznych, w ogóle istnienie tych miejscowości. Błędy, jakie były związane z likwidacją rozdrobnionego rolnictwa np. w Hiszpanii, spowodowały przemieszczenie się milionów ludzi do wielkich miast, do metropolii i wyludnienie, pustynnienie prowincji hiszpańskiej. My tego błędu popełnić nie chcemy. Odejście od programu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego prowadzonego przez naszych poprzedników na rzecz rozwoju zrównoważonego jest właśnie tym racjonalnym działaniem na rzecz wzmocnienia terenów poza wielkimi miastami. Można zastosować kryterium wielkości ekonomicznej: do 13 tys. euro. Ono jest trochę mechanicznym ustaleniem pewnej granicy dostępności środków dla jednej czy dla drugiej grupy gospodarstw. Korzystają one ze wszystkich form wsparcia. To przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trwają kolejne nabory, będą także realizowane kolejne nabory. Z tego korzystają różne gospodarstwa.

Uprościliśmy warunki, które tego programu dotyczą.

To się wiąże z poprzednim pytaniem. Również umożliwienie wsparcia zakupu maszyn rolniczych w związku z realizacją inwestycji budowlanych z zakresu rozwoju produkcji zwierzęcej, dodatkowa forma pomocy w formie gwarancji bankowych. Zniesienie obowiązku ubezpieczenia w KRUS przed dniem złożenia wniosku o wsparcie. To był pewien zabieg może bezpiecznościowy, ale dość nielogiczny. Małe gospodarstwa z reguły to są gospodarstwa dwuzawodowców. Ktoś w rodzinie, często również prowadzący gospodarstwo rolnik, musi dorabiać w innych miejscach pracy, bo to gospodarstwo nie daje wystarczających środków na godziwe utrzymanie rodziny, a w związku z podjęciem pracy w innych podmiotach z konieczności wypadał z ubezpieczenia KRUS-owskiego na rzecz ubezpieczenia ZUS-owskiego. A więc rozdzieliliśmy możliwość udzielania pomocy - niezależnie od tego, z jakiej formy ubezpieczenia społecznego rolnik korzysta. To jest forma, z której korzystają wszystkie typy gospodarstw, również gospodarstwa mniejsze. Właściwie działaniem dedykowanym przede wszystkim mniejszym gospodarstwom, które ma umożliwić realizację sprzedaży, urynkowienie produktów wytwarzanych na stosunkowo niewielką skalę w gospodarstwach, jest gwałtowny rozwój i stworzenie odpowiednich przepisów prawa na rzecz rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej, również rozwoju małych przetwórni surowców pochodzenia zwierzęcego w ramach produkcji małej, lokalnej i ograniczonej. To się bardzo rozwija, głównie małe gospodarstwa się tym zajmują.

Podniesiona została kwota premii w przypadku zatrudnienia jednej osoby, w tym samozatrudnienia, do 150 tys., 200 tys. - w przypadku zatrudnienia dwóch osób, 250 tys. - w przypadku zatrudnienia trzech i więcej osób. To jest również zachęta do rozwoju przedsiębiorczości i pewnej zaradności. Nowa perspektywa. Tak, bardzo pilnujemy tego, żeby te mniejsze gospodarstwa w Polsce miały odpowiednią pozycję i w łańcuchu od pola do stołu, ale również żeby były im dedykowane wydzielone, szczególnie korzystne formy wsparcia, bo chcemy te gospodarstwa po prostu utrzymać. Ważne są nie tylko, jeszcze raz powtórzę, z powodów [[Dzwonek]] produkcyjnych, ale również w odniesieniu do rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów wiejskich.

Zachęcam panów posłów do szczegółowego zapoznania się z tym planem.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister przekrojowo praktycznie odniósł się do wszystkich tematów, które nawiązują do wsparcia małych i średnich gospodarstw w Polsce. Chciałbym dopytać, panie ministrze, ponieważ na jednym ze spotkań z rolnikami, bodajże w Kadzidle, ten temat się przewijał, był omawiany dość szczegółowo, właśnie temat sprzedaży bezpośredniej, o której pan minister mówił.

Czy może już jakaś strategia w tym zakresie jest wypracowana?

Bo wiemy, że duże już potrafią doskonale wykorzystywać środki unijne, europejskie. I jeszcze jedno pytanie, dotyczące. Bo już były dwa.

Ja nie wiem, co jeszcze w tym handlu poprawić. Wszystko, co w gospodarstwie urośnie, urodzi się, może być bezproblemowo przetworzone przez rolnika bez konieczności budowania oddzielnej fabryki czy jakichś pomieszczeń produkcyjnych - symbolicznie, że tak powiem, w kuchni, w której gospodyni przygotowuje pokarm dla tych, których najbardziej kocha, dla swojej rodziny. Rozwiązania są proste, nie wymagają zgody ani zezwoleń ze strony powiatowego lekarza weterynarii czy inspektora sanitarnego. Oczywiście kontrole będą i ja będę pierwszym, który nie dopuści do tego, żeby żywność bez kontroli trafiała na rynek.

Ale to jest duży obszar. Nie sądzę, żeby te produkty, produkowane przecież na stosunkowo niewielką skalę, musiały podlegać długim łańcuchom dystrybucji i krążyć gdzieś po świecie. Ten zapis jest absolutnie wystarczający, a jeszcze jest rozszerzony o to, że w ramach różnego rodzaju wydarzeń społeczno-kulturalnych, festynów, pokazów może to się odbywać na terenie całej Polski. Również wspieramy to finansowo. Pierwszy nabór, taki sondażowy, odbył się w lutym.

Te wnioski są w tej chwili w agencji obrabiane. Powtórzymy nabór, bo trochę środków jeszcze zostało, w sierpniu, we wrześniu. Trudno mi tu mówić o jakimś precyzyjnym terminie, ale nabory będą powtarzane. Na wsparcie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i MOL będziemy szukali pieniędzy również poza tą kwotą, którą w tej chwili dysponujemy. Ukierunkowanie na wsparcie mniejszych gospodarstw wynika z polityki rządu, polityki Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniałem przy poprzednim pytaniu o dużym programie [[Dzwonek]] wapnowania. Proszę być spokojnym, panie pośle. Przy tych wszystkich nowych strategiach, planach strategicznych związanych z nową perspektywą finansową właśnie małe gospodarstwa będą najbardziej preferowanymi beneficjentami. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie zadają posłowie Monika Wielichowska, Monika Rosa, Ewa Lieder i Mirosław Suchoń, klub Platformy Obywatelskiej, w sprawie nowej listy leków refundowanych. Pierwsza pytanie zadaje pani poseł Monika Wielichowska. Wysoka Izbo! Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz - księgowym, a szpital - przedsiębiorstwem. Każdy polski obywatel ma czuć się bezpiecznie wtedy, kiedy potrzebuje pomocy medycznej. Ma wiedzieć, że ta pomoc zostanie mu udzielona szybko, że będzie bezpieczny i że będzie to pomoc bezpłatna. Państwo ma dbać o zdrowie ludzi, a nie tworzyć nieludzkie procedury. Trzeba skończyć z bylejakością. To wypowiedzi pani premier Beaty Szydło. Mijają 4 lata. Ludzie umierają na SOR-ach, powiatowe szpitale są na skraju finansowego bankructwa. W historii nie było dłuższych niż dziś kolejek do lekarzy, a nowa lista leków refundowanych to lista waszej hańby, bo wielu chorych skazujecie na śmierć i cierpienie. W szczególności w trudnej sytuacji znajdują się chorzy na EB. Ta choroba w skali całej Polski dotyka kilkudziesięciu osób; kilkanaścioro z nich to dzieci. EB powoduje złuszczanie się naskórka i niesłychany ból od najmniejszego nawet dotknięcia. Są opatrunki, które działają na tyle delikatnie, że można je zmienić bez kolejnego zrywania naskórka. Te opatrunki w 2015 r. kosztowały miesięcznie 372 zł. Za waszych czasów, za czasów PiS-u, kosztowały 4 tys. zł, by od kilku dni kosztować 6 tys. zł miesięcznie. Tak wygląda opiekuńcze państwo? To skazywanie chorych na okrutne cierpienie. W dramatycznej sytuacji są także chorzy na rzadką chorobę Fabry’ego, 220 tys. pacjentów z cukrzycą, zaawansowanym rakiem jelita grubego i rakiem piersi. Bez dostępu do preparatu żywieniowego zostali chorzy na mukowiscydozę. Tak wygląda ta dobra zmiana? Wydajecie miliardy na kłamstwa i manipulacje telewizji, kiedyś publicznej. Wydajecie miliony na limuzyny z lodówką i [[Dzwonek]] z telewizorem.

Obydwa leki cały czas są na liście leków refundowanych.

Firmy, negocjując, bardzo często mówią, ponieważ jest wspólna grupa limitowa i to pacjent dopłaca, że pacjentowi nie zależy na tym, że może płacić więcej i więcej, że pacjent chce dopłacać do leków, pacjent chce dużo dopłacać. My się z tym nie zgadzamy i negocjujemy również w imieniu pacjenta - nie tak jak firmy chcą, tylko w imieniu NFZ, tylko również w imieniu pacjenta. W związku z tym zmniejszamy ceny dla pacjenta.

Jeśli chodzi o lek w zakresie poszerzenia wskazań do stosowania dla pacjentów opornych na kastrację raka gruczołu krokowego, to jest aktualnie stosowany jeden lek, który został objęty blisko 2 lata temu poszerzonym wskazaniem.

Nie możemy przy identycznych wskazaniach, przy identycznym zakresie przyjmować leku po znacząco wyższej cenie.

Nie możemy za tę samą terapię znacząco drożej płacić tylko i wyłącznie dlatego, że firma nam się podoba.

Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Ewa Lieder. Szanowni Państwo! Przedstawiciele ministerstwa często mówią, że zmiany na liście leków refundowanych nie stanowią żadnego problemu - o tym pan też mówił - bo pacjenci mogą korzystać z leków biopodobnych lub środków zastępczych. Tymczasem zmiana leków na inne o podobnym działaniu może negatywnie oddziaływać na organizm chorego. W związku z tym pojawia się pytanie, jakimi kryteriami kieruje się minister, decydując o tym, którzy pacjenci mają ryzykować pogorszenie swojego zdrowia przy zmianie leku.

Co 3 miesiące - dla starszych osób, proszę państwa, to jest naprawdę wielki niepokój. Obserwuję swoją mamę, która czyta te listy, i to jest naprawdę okrutne.

Widzimy ostatnio oszczędności na leku oryginalnym biopodobnych adalimumabów - ceny już są ponad ośmiokrotnie niższe niż były do tej pory.

W 2003 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy powstał pierwszy w Polsce ośrodek pozytonowej tomografii emisyjnej, w skrócie PET. Tomografia pozytonowa stanowi wyspecjalizowany system, który pozwala na wczesną ocenę zaburzeń biochemicznych w obrębie zmienionego chorobowo narządu z dokładną lokalizacją zmian chorobowych. W 2006 r. pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości opracował „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, który przewidywał powstanie w Polsce kilku ośrodków PET. W okresie ostatnich lat liczba tych ośrodków bardzo wzrosła. Z szacunków niezależnych ekspertów europejskich wynika, że zapotrzebowanie w Polsce na badania PET wynosi 70 330 badań rocznie i docelowo szacuje się, że powinno powstać 28 ośrodków diagnostycznych. Panie Ministrze! Ile funkcjonuje obecnie w Polsce takich ośrodków z wykorzystaniem urządzeń typu PET? Wiem, że te ośrodki pokrywają całą mapę Polski, są we wszystkich województwach. Ale w których województwach znajduje się najwięcej ośrodków PET? Jakie jest kryterium kontraktowania usług na urządzenia PET znajdujące się w jednostkach zdrowia? I takie pytanie związane już może z moim regionem, ze stolicą województwa podkarpackiego, w której nie ma ośrodka PET. Chciałem zapytać: W których miastach wojewódzkich w Polsce nie ma jeszcze ośrodków pozytonowej tomografii emisyjnej? Bardzo dziękuję. Odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Maciej Miłkowski.

Panie Ministrze! Samorząd województwa podkarpackiego wspierany przez wojewodę podkarpackiego czyni starania, aby w Rzeszowie, w stolicy województwa, zainstalowano w Szpitalu Klinicznym nr 1 urządzenie typu PET. Dyrekcja szpitala przygotowała na własny koszt specjalne pomieszczenia, żeby PET mógł być zainstalowany, Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył 2 mln zł na zakup tego urządzenia. I, panie ministrze, mam takie pytanie, dopytanie: Czy Ministerstwo Zdrowia może udzielić wsparcia finansowego na ten cel w Rzeszowie? Uniwersytet Rzeszowski - chcę nadmienić, że młody uniwersytet - kształci na kierunku lekarskim młodych lekarzy, a powstanie w Rzeszowie ośrodka pozytonowej tomografii emisyjnej w Szpitalu Klinicznym nr 1 wzbogaciłoby infrastrukturę dydaktyczną Uniwersytetu Rzeszowskiego [[Dzwonek]] i pomogłoby kształcić w tym celu studentów. Dziękuję bardzo. Ponownie odpowiada podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pan Maciej Miłkowski. Bardzo proszę.

Jako pierwsza pytanie zadaje pani poseł Gabriela Lenartowicz. Panie Ministrze! Chciałam zapytać o sytuację, która miała miejsce w ostatnich kilku dniach. Polaków zelektryzowała bulwersująca wiadomość o ryzyku utraty miliardów euro z przyszłej perspektywy finansowej na walkę ze smogiem. W związku z tym, że pojawiały się informacje zaprzeczające temu, chciałabym zapytać przede wszystkim o to, kto tak naprawdę w imieniu rządu polskiego negocjował i kto otrzymał list od Marka Lemaître’a, komisarza Komisji Europejskiej do spraw rozwoju regionalnego i miast i jakie jest stanowisko rządu polskiego wobec tego ultymatywnego w treści pisma. I tak naprawdę kto odpowiada za te negocjacje i ewentualne ryzyko utraty tych środków, bo w tej chwili mamy sytuację taką, jak w tym przysłowiu ludowym: kowal zawinił, cygana powiesili? Chcielibyśmy wiedzieć, kogo mamy rozliczać jako Polacy z tego, w jak skuteczny sposób zabiega o wsparcie europejskie w kwestii tak poważnego problemu, który mają Polacy, z powodu którego umierają ich dziesiątki tysięcy rocznie wcześniej. Dziękuję. Dziękuję. Drugą część pytania zadaje pan poseł Ryszard Wilczyński. Panie Ministrze!

Przechodzę na lokalne podwórko.

Bardzo proszę.

Bardzo dziękuję za możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania pana posła.

Jest to oczywiście naturalny proces związany z tym, że program cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów.

To również on jest osobą, która dyskutuje na temat przyszłości alokacji funduszy europejskich dla Polski na następną fazę finansowania.

Jeżeli chodzi o optymalizację programu, to oczywiście prowadzimy takie prace. W naturalny sposób jest to przedsięwzięcie mające bardzo fundamentalne, cywilizacyjne znaczenie dla naszego kraju. To jest potężny potencjał 3 mln domów.

Dotyczy to również kwestii sposobu dystrybucji środków.

To tyle z mojej strony, panie marszałku, bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Z całym szacunkiem, ale wielosłowie ani nie namnoży pieniędzy, ani nie odpowie ma pytania Polaków. Ja panu odpowiem, dlaczego ten program nie działa. Pan mówi - 103 mld.

Dlatego ten program nie działa - nie macie na to pieniędzy. Robicie wszystko, żeby stworzyć bariery, bo jest to wielka fikcja. To nie jest czyste powietrze, to jest czysta fikcja. Stąd się to bierze. Dostęp do tego programu jest żaden. Konstrukcje są takie, że biednych na to nie stać, a bogaci nie mają dostępu. Tak jest od wyborów do wyborów.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Michał Kurtyka. Bardzo dziękuję.

Po drugie, my w tym momencie robimy wszystko, żeby ten program uprościć, by przyspieszyć alokację funduszy i ułatwić Polakom korzystanie z tych środków. Jednym z elementów jest włączenie gmin. To jest ten partner, który ma bezpośredni kontakt z obywatelem. My w tym momencie chcemy wprowadzić zmianę w postaci uproszczenia wniosków oraz procedury weryfikacji. Jednym z najbardziej istotnych uproszczeń, jakie planujemy, będzie domniemanie podpisania umowy przez beneficjenta w momencie składania wniosku. Innymi słowy, chcemy, żeby maksymalnie łatwo było naszym obywatelom takie wnioski podpisywać. A zatem zlikwidujemy konieczność podwójnego przychodzenia, umowa stanie się wiążąca po decyzji zarządu odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Bardzo dziękuję.

Bardzo proszę, jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Andrzej Melak. Nasze pytanie dotyczy w ogóle polityki klimatyczno-energetycznej polskiego rządu. Komisja Krajowa z wielkim uznaniem odnosi się do tego, co polski rząd w tej sprawie robi. Cytuję: „Solidarność” z ogromną aprobatą przyjęła odrzucenie przez polską delegację wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej dotyczących kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Trzeba jasno i wyraźnie pokreślić, że akceptacja zapisów o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. oznaczałaby katastrofę dla polskiej gospodarki oraz trwałe zubożenie mieszkańców naszego kraju.

Wcześniej, zwłaszcza w trakcie rządów poprzedniej koalicji, ponosiliśmy na tym polu wyłącznie dotkliwe porażki. Trzeba pamiętać, że Polska w ostatnich dziesięcioleciach wykonała ogromny wysiłek dotyczący redukcji CO2 i z nawiązką wypełniła zobowiązania zawarte w protokole z Kioto. Tymczasem najwięksi emitenci tego gazu, USA, Indie, Chiny, także inne kraje, nie podejmują adekwatnych działań w tym zakresie. Duże firmy europejskie lokują produkcję, często uciążliwą dla środowiska, w krajach poza Europą. W tej sytuacji przyjmowanie kolejnych celów redukcyjnych przez Unię Europejską odbywa się kosztem obniżenia konkurencyjności europejskiej gospodarki, likwidacji przemysłu i radykalnego wzrostu cen energii. Jak na tle innych krajów europejskich wygląda bilans emisji CO2 w Polsce i czy w bilansie przodujących gospodarek europejskich [[Dzwonek]] liczą się także zakłady pracujące poza Europą? Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pan Michał Kurtyka. Bardzo proszę, panie ministrze.

Dotyczy ono absolutnie fundamentalnej kwestii, która jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej, ale również wykracza poza nasze europejskie podwórko, dlatego że mamy przed sobą szczyt sekretarza generalnego Antonio Guterresa, który będzie odbywał się 23 września w Nowym Jorku. Przedmiotem prac zarówno na poziomie unijnym, jak i na poziomie ogólnoświatowym jest kolejna perspektywa, w tym kolejny rozdział, jeżeli chodzi o składanie przez państwa strony porozumienia paryskiego krajowych kontrybucji, tzw. NDC. Jednym z elementów krajowych kontrybucji są oczywiście cele na 2030 r. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarkę unijną, takim przedmiotem debaty, również na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej, jest kwestia neutralności klimatycznej. To był jeden z tych elementów, na który również Polska na konferencji w Paryżu zwracała uwagę, a mianowicie że niezbędne jest uzyskanie równowagi pomiędzy emisjami i pochłanianiem dwutlenku węgla. Z tego powodu to sformułowanie „neutralność klimatyczna” nie sygnalizuje od razu, że we wszystkich państwach członkowskich czy też we wszystkich sektorach gospodarczych należałoby zlikwidować emisję. Natomiast należałoby zrównoważyć sumę tych emisji sumą pochłaniania. Niewątpliwie osiągnięcie neutralności klimatycznej to jest nie tylko ogromne wyzwanie dla sektora energetycznego, co zostało zawarte w pytaniu pana posła, ale również wyzwanie cywilizacyjne, ponieważ mówiąc o neutralności klimatycznej, mówimy również o takich sektorach jak transport, i to jest dyskusja, która przecież już zawitała na forum unijnym, jak również w Polsce, jeżeli chodzi o kwestię elektromobilności, ale to wykracza również poza ten sektor. Wchodzimy tutaj w kwestię przemysłu, produkcji towarów, wchodzimy również w kwestię rolnictwa. Jako Polska jesteśmy w środku stawki unijnej, jeżeli chodzi o wielkość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na głowę, na mieszkańca. To nieco kontrintuicyjne w stosunku do dyskusji, w której sugeruje się, że Polska byłaby ponadwymiarowym emitentem gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Największym emitentem pozostaje nasz zachodni sąsiad, Niemcy, to jest ok. 20% gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dla porównania Polska emituje nieco ponad 9%. Natomiast jako cała Unia Europejska jesteśmy odpowiedzialni za ok. 10% globalnych emisji i ten udział Unii Europejskiej w emisjach stopniowo maleje. Same Chiny to jest 20%, Stany Zjednoczone to kolejne 15% światowych emisji.

Jeżeli myślimy o neutralności klimatycznej, to dzisiaj ta dyskusja koncentruje się na tych źródłach emisji CO2, które są zawarte na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, natomiast nie odnosi się do konsumpcji towarów. Mamy do czynienia z tego typu sytuacjami, w których nawet zdawałoby się trudne do przewożenia, ciężkie towary są importowane z krajów, które emitują, i w tej sytuacji narasta rozbieżność pomiędzy produkcją śladu węglowego czy też emisji na poziomie Unii Europejskiej a konsumpcją towarów, w których zawarta jest emisja, które pochodzą z importu. Niewątpliwie jest to jedno z wyzwawań nie tylko dla europejskiej, ale również dla światowej polityki klimatycznej. Partykuły CO2 nie mają paszportów i niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, w dalszym ciągu trafiają do atmosfery. Dziękuję bardzo. Dziękuję, już nie mam dodatkowego pytania, odpowiedź była pełna, wyczerpująca. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. To pytanie kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego. Przypominam, że na obecnym posiedzeniu Sejmu zostanie rozpatrzona informacja w sprawie doniesień medialnych dotyczących apelu banków o wsparcie przez rząd Polski w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w procesie dotyczącym tzw. kredytów frankowych, o którą wnosił Klub Poselski Kukiz’15. Przypominam również, że przedstawienie uzasadnienia wniosku przez posła przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a udzielenie odpowiedzi przez przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Wystąpienia posłów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty. Na zakończenie dyskusji głos zabierają kolejno przedstawiciel wnioskodawców oraz przedstawiciel Rady Ministrów. Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawców nie może trwać dłużej niż 5 minut, a wystąpienie przedstawiciela Rady Ministrów - dłużej niż 10 minut. Marszałek Sejmu może wyrazić zgodę na wydłużenie wystąpienia przedstawiciela Rady Ministrów. Czas przeznaczony na rozpatrzenie punktu: Informacja bieżąca nie może być dłuższy niż 90 minut.

Chciałoby się powiedzieć: A nie mówiłem? Bo tak się składa, że klub Kukiz’15, że ja jako poseł wnioskodawca tym tematem zajmuję się od 4 lat.

Abuzywność, o której od 4 lat z tej mównicy mówię jak mantra, rzecznik finansowy mówi, UOKiK mówi, sąd pierwszej instancji, drugiej instancji, Sąd Najwyższy. Milczą. Są ślepe, głuche i nie reagują.

Jedni mówią, że cała umowa jest nieważna. Inni przeciwnie: klauzula jest nieważna, a co za tym idzie - również umowa. Trzeci pogląd jest taki, że klauzulę trzeba uważać za nieistniejącą, a umowę za obowiązującą, z tym że skoro nie ma w niej umowy o indeksacjach i zasadach wyliczenia rat w walutach obcych, kredyt walutowy zamienia się na złotowy oparty na LIBOR, a przypomnę, że dzisiaj LIBOR jest ujemny. Proszę państwa, bardzo długo z tej mównicy słyszałem: widziały gały, co brały. A dzisiaj możemy powiedzieć: widziały gały, co dawały. Bo każda umowa, proszę państwa, ma dwie strony: dającą i biorącą, podpisy są dwóch stron i jest akceptacja dwóch stron. Na dzisiaj, proszę państwa, przeraża mnie jedna rzecz, że oto dzisiaj ktoś, kto wszedł świadomie w proceder tzw. pseudokredytów frankowych, które na dzisiaj - wszyscy doskonale to wiedzą - są poważnym problemem, żeby nie powiedzieć: przestępstwem wobec polskiego konsumenta, Polaka, ten problem próbuje sprzedać polskiemu rządowi. Mówiły: niech ludzie idą do sądów. Panie premierze, ratunku, toniemy. Jak podaje „Puls Biznesu”, to będzie 60 mld. Nie mówimy o drobnych, proszę państwa. To są dobre 3 lata czy 2 lata 500+. Czy polski rząd na serio traktuje polskich obywateli? Czy polski rząd zamienia się w adwokata broniącego banków? Ja tylko powiem, że banków prywatnych mamy więcej niż 24, a 10 jest skażonych tymi kredytami. To oznacza, że nie mamy problemu 100% polskiego systemu bankowego, ale mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, które było wygodne przez lata, zarabiania przez tłuste kocury bankowe [[Dzwonek]] dużych pieniędzy, a dzisiaj one krzyczą, że nie mają pieniędzy. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o udzielenie odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana Piotra Wawrzyka. Bardzo proszę, panie ministrze.

Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o którym mowa w wystąpieniu pana posła, znajduje się obecnie na końcowym etapie. Wniosek prejudycjalny w tej sprawie został złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 16 kwietnia ub.r.

Etap pisemny postępowania został zakończony w listopadzie ub.r., a Trybunał zrezygnował w tej sprawie z przeprowadzenia rozprawy. Obecnie oczekujemy już tylko na ogłoszenie wyroku, które powinno nastąpić w ciągu najbliższych tygodni, natomiast konkretna data nie jest jeszcze określona. Obecnie więc, ze względu na etap postępowania, nie jest już możliwe przedkładanie dodatkowych, uzupełniających uwag pisemnych, jak to postuluje Związek Banków Polskich. Trzeba też wyraźnie przy tym podkreślić, że środowisko bankowe było reprezentowane w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości, ponieważ uczestnikiem tego postępowania jest jeden z prywatnych banków, który przedstawił w postępowaniu bardzo obszerne uwagi pisemne. Środowisko bankowe miało więc pełną możliwość, aby swoje racje i argumenty przedstawić Trybunałowi, i z tej możliwości skorzystało. Jeżeli chodzi o stanowisko rządu, to jego celem była przede wszystkim ochrona praw słabszej strony kredytów walutowych, tzn. konsumentów.

Przypomnę przy tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie, który zwrócił się z pytaniem do Trybunału, rozstrzyga sprawy konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich. W umowie kredytu bank zawarł niedozwolone postanowienie umowne dotyczące sposobu obliczania kursu franka. Bank zastrzegł mianowicie, że to on w swojej tabeli określa i jednoznacznie podaje kurs, według którego oblicza się sumę kapitału do spłaty i wysokość raty kredytu zaciągniętego we frankach, które konsument musi spłacić w złotówkach. Nie budzi wątpliwości również w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że takie postępowanie jest niedozwolone w rozumieniu dyrektywy, o której wspomniałem, a w konsekwencji nie wiąże konsumenta. Problem prawny dotyczy tego, jak po wyeliminowaniu takiego niedozwolonego postanowienia umownego dalej spłacać kredyt. W tej sytuacji konsumenci żądają alternatywnie albo uznania umowy za nieważną, co wiąże się z koniecznością natychmiastowego oddania bankowi takiej sumy, jaką bank pożyczył konsumentowi, albo też dalszego spłacania kredytu, ale w złotówkach, takiej sumy, jaką konsument rzeczywiście otrzymał od banku, przy zachowaniu niższego oprocentowania obejmującego marżę oraz stawkę LIBOR dla franka szwajcarskiego. Ponieważ obie opcje są niekorzystne dla banku, bank chciałby utrzymać ważność umowy przy zastąpieniu postanowienia niedozwolonego kursem franka ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski. W konsekwencji sąd okręgowy spytał, czy dyrektywa o nieuczciwych warunkach umownych pozwalałaby na zastąpienie postanowienia niedozwolonego w oparciu o kurs franka, ustalony na podstawie klauzul generalnych, wynikający z Kodeksu cywilnego, tj. w oparciu o zasady współżycia społecznego albo zwyczajów. To, zdaniem sądu, pozwoliłoby na zastąpienie postanowienia niedozwolonego kursem ustalanym według innego wskaźnika, np. ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Obecnie w Polsce toczy się kilka tysięcy podobnych spraw, które są zawieszone w oczekiwaniu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rząd wskazał, że uzupełnienie luk w umowie w oparciu o przepisy prawa krajowego, które zawierają klauzule generalne, w żadnym wypadku nie jest możliwe, jeżeli skutkiem uznania określonych postanowień umownych za nieuczciwe byłby korzystny dla konsumenta upadek całej umowy. Ocena skutków upadku całej umowy jest dokonywana przez konsumenta po uprzednim pouczeniu go przez sąd o wszystkich tych skutkach. Ocena wyrażona przez konsumenta powinna zostać uwzględniona przez sąd przy rozstrzyganiu o skutkach uznania postanowienia za niedozwolone. Jakie mogą być skutki wyroku Trybunału? Banki, które zawierały umowy kredytów we frankach szwajcarskich zgodnie z obowiązującym prawem, tzn. nie zamieszczały w tych umowach nieuczciwych klauzul, nie muszą się obawiać żadnych niekorzystnych skutków. Z kolei banki, które z naruszeniem prawa wykorzystywały swoją przewagę nad konsumentem i wprowadzały do umów kredytów nieuczciwe klauzule, muszą liczyć się konsekwencjami wynikającymi z prawa unijnego, tak jak każdy przedsiębiorca, który dopuszcza się podobnych praktyk. Prawo unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości bardzo wyraźnie i jednoznacznie chronią słabszą stronę umów kredytowych, jaką są kredytobiorcy. Stanowisko polskiego rządu przedstawione w postępowaniu przed Trybunałem w całości opiera się na wspomnianej dyrektywie oraz dotychczasowym orzecznictwie Trybunału. Do tej pory orzecznictwo polskich sądów w sprawach konsumenckich nie było jednak jednolite. Nie zawsze uwzględniało wymagania prawa unijnego i nie zawsze skutecznie chroniło słabszą stronę umów kredytowych. Mamy zatem nadzieję, że wyrok Trybunału w tej sprawie przyczyni się do tego, że wymagania wynikające z dyrektywy i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostaną spopularyzowane zarówno wśród polskich sądów, jak i w sektorze bankowym i będą w przyszłości zapobiegać stosowaniu przez banki niedozwolonych postanowień umownych. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z pan i panów posłów chce jeszcze zapisać się do głosu? Jako pierwszy głos ma pan poseł Jan Szewczak, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Szkoda, że pan minister uznał, że stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej akurat w tej sprawie jest konieczne, i że zapomniał pan o tym, że przecież wasz prezydent 4 lata temu obiecał wszystkim frankowiczom, że przewalutuje kredyty po kursie z dnia zaciągnięcia. Do innych rzeczy stanowisko TSUE nie jest wam potrzebne, a czasem wam wręcz przeszkadza. W tej sytuacji czekacie na to stanowisko nie wiadomo dlaczego. Sprawa jest oczywista. To, że premier Morawiecki jest niezwykle życzliwy dla banków i że rząd PiS-u podjął szereg decyzji, które wspierają bankowców, właścicieli banków, zarządy banków, a są niekorzystne dla obywateli - to wiemy wszyscy. Po co? Po to, żeby tworzył miejsca pracy w Polsce. Gdzie? Nie na wschodzie. Nie w małych miasteczkach. W Warszawie. Czy w Warszawie jest bezrobocie? Czy zachodni bogaty bank musi dostać 20 mln polskich podatników, żeby tworzyć miejsca pracy i zarabiać w Polsce? Takie rzeczy tylko premier Morawiecki potrafi wymyślić. Narzędzie uszczelniające.

Banki nimi obracają, zarabiając ogromne pieniądze, a polski rząd musi zaciągać zobowiązania, długi i te długi później spłacać - znowu z pieniędzy polskiego podatnika.

Bardzo proszę, pan poseł Andrzej Maciejewski, Klub Poselski Kukiz’15. Panie Ministrze! W toku naszych dyskusji, pytań na pewno padnie wiele sformułowań i zwrotów, ale one będą miały jedną puentę - afera frankowa.

Ale mam tu bardzo konkretne pytanie do pana premiera, do strony rządowej. Chciałbym, żeby opinia publiczna dowiedziała się - to jest bardzo ważne też w interesie pana premiera, chodzi o transparentność i jasność - że pan premier, jako były bankowiec, gra fair i nie ma żadnych ukrytych intencji. Mnie interesuje odpowiedź na bardzo ważne pytanie: Ile pieniędzy przez ostatnie lata, przed wprowadzeniem podatku bankowego, wypłynęło czy ile banki zagraniczne będące w Polsce przekazały swoim centralom za granicą? To były grube miliardy. Rzecz trzecia, bardzo istotna, panie ministrze. Pytanie: Czy polski rząd wreszcie podejmie działania prawne wobec osób, instytucji zaangażowanych w aferę frankową? Nazywam to aferą frankową, bo NIK potwierdził zaniechania urzędów i agend rządowych. Jak trzeba, idzie do więzienia.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoki Sejmie! Chcę przede wszystkim podziękować panu ministrowi za wyczerpujące, dokładne i gaszące niepotrzebne emocje w tej trudnej sprawie stanowisko rządu. Tak, najważniejsza jest norma sprawiedliwości społecznej. Nią się kierujemy i na tym polega zmiana sytuacji. A jeżeli chodzi o tzw. obronę banksterów i bankowców, to trzeba, proszę państwa, zajrzeć do Internetu i sprawdzić, kto w co grał, kogo bronił i za kim jest. To nie kto inny jak właśnie opozycja, może nie cała, ich broniła, i to jeszcze z wielkim patosem, strasząc polski parlament, że jeżeli skubniemy na 2 mld banki, mówię o podatku bankowym - to wszystko można sprawdzić - to banki odkują się kosztem zwykłych Nowaków, Malinowskich, Zielińskich, Zakrzewskich i innych. Jest pytanie w tym momencie, kto ma za co płacić. Prawo to jest jedna kwestia, a poczucie elementarnej sprawiedliwości - druga.

Wszyscy, nawet nieprawnicy, o tym wiedzieli. To nie jest tak, że.

Banki drżą. A to, że się zwracają? Zwracają się, były pisma - o to pyta teraz opozycja - ale polski rząd się nie ugiął, nawet nie brał tego pod uwagę. Przechodzę do pytania, bo czas już jest króciutki.

Pani poseł Małgorzata Pępek. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Historia pomysłów, które miały pomóc polskim frankowiczom, jest tak długa, że na tej podstawie można by napisać książkę. Przez ostatnie 4 lata mieliśmy do czynienia z prawdziwym festiwalem propozycji i projektów ze strony rządu. Jaki jest efekt, każdy z państwa widzi. Kredytobiorcy, którzy przed laty zadłużyli się w szwajcarskiej walucie, są w matni. Spłacają raty, a ich dług rośnie. Najwięksi pechowcy mają do spłacenia dwa razy więcej, niż dostali z banku. Według Biura Informacji Kredytowej pod koniec 2018 r. w Polsce spłaconych było 470 tys. kredytów we frankach o łącznej wartości aż 107 mld zł. Realnej pomocy, jak nie było, tak nie ma. Pan prezydent podczas kampanii wyborczej obiecywał wszem i wobec przewalutowanie kredytów. Co z tymi obietnicami, drodzy państwo? Sytuacja jest na tyle poważna, że bankowcy, bojąc się katastrofy, zwrócili się do premiera o pomoc. Panie premierze, co zamierzacie z tym zrobić? Czy dalej będziecie ludziom mydlić oczy i udawać, że coś robicie? Bo to jest zwyczajne mydlenie oczu. Po 4 latach waszych rządów społeczeństwo czuje się oszukane. Naobiecywaliście bardzo dużo i na tym się skończyło. Z roku na rok bagatelizujecie ten problem, a tutaj potrzeba realnej pomocy. Bardzo proszę, pan poseł Stefan Romecki. Panie Ministrze!

W związku z tym mam dwa pytania. Czy rząd stanie po stronie poszkodowanych polskich obywateli, czy będzie bronił prywatnych zagranicznych banków? I drugie pytanie: Jakie są zyski banków z tytułu sprzedaży toksycznych produktów bankowych, zwanych powszechnie kredytami bankowymi? Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć, panie pośle, tra ta ta ta, tra ta ta ta i mijają 4 lata, a rząd PiS-u nie rozwiązał problemu frankowiczów, [[Oklaski]] a jak wiemy, to była obietnica wyborcza pana prezydenta z waszego środowiska.

Jeśli decyzja TSUE zostanie potwierdzona i będzie tak, jak zapowiedział rzecznik generalny, to jak szacują eksperci kosztować to będzie banki od 60 do 80 mld zł i ta kwota będzie wyższa niż przewiduje jakikolwiek projekt prezydencki, panie pośle. Bankowcy już apelują o wsparcie do rządu, a ja pytam pana premiera Morawieckiego, dlaczego ma pomagać bankierom, a nie obywatelom. Dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpowiedzi na jedno z pytań już wcześniej stwierdził, że umowa nie może upaść wbrew interesowi konsumenta. I to konsument wskazuje, co leży w jego interesie. Polska od kilku lat wprowadza tę zasadę. Bardzo ważny dla mniej zamożnych kredytobiorców jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który procedowaną obecnie ustawą mamy zamiar uelastycznić.

Wskazane byłoby, moim zdaniem, przeprowadzić analizę, którym konsumentom, którzy wzięli kredyt w walucie obcej, opłacałoby się ewentualnie przewalutowanie czy zmiana ich umów, a którym nie. Którzy kredytobiorcy, zdaniem pana ministra, w zależności od roku udzielenia im kredytu, stracili na tym, że wzięli kredyt we frankach czy w innej obcej walucie, a którzy nie. Dziękuję bardzo. Naszej debacie przysłuchują się przedstawiciele stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, których serdecznie pozdrawiamy. Bardzo proszę, pan poseł Marek Wójcik. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dziś rozmawiamy o skutkach finansowych kredytów frankowych dla polskiego systemu bankowego, natomiast trzeba przypomnieć, że 4 lata temu prezydent Andrzej Duda obiecywał, ale też politycy PiS-u w kampanii wyborczej obiecywali rozwiązać problem kredytów we frankach. Obiecywali i część obywateli państwu uwierzyła, głosowała na państwa, wierzyła w to, że takie ustawy rzeczywiście zostaną przyjęte. Niestety czas pokazał, że to były tylko pozorowane działania. Do Sejmu wpłynęły dwie ustawy: jedna w sierpniu 2016 r., druga w sierpniu 2017 r., dwa prezydenckie projekty, które w zamyśle miały pomóc frankowiczom, a okazało się, że są to tylko i wyłącznie pozorowane działania w tej sprawie. Co więcej, ci frankowicze, którzy uwierzyli państwu i liczyli na ustawę, są w gorszej sytuacji, dlatego że z roku na rok, z miesiąca na miesiąc koszty ich kredytów rosną i tracą oni coraz więcej pieniędzy.

Wczoraj jakieś pozorowane działania, ale przecież do końca kadencji Sejmu zostały raptem dwa posiedzenia. Nieufność pana Ryszarda wzrosła, kiedy premierem polskiego rządu został pan Mateusz Morawiecki, były prezes banku udzielającego kredytów we frankach.

Pan poseł Jan Kilian, zapraszam. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak, to prawda, jest jedna sprawa, bardzo poważny problem, który nie doczekał się rozwiązania. 90% różnych bardzo trudnych spraw zostało rozwiązanych przez minione 4 lata. Cóż, rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze kieruje się zasadą pomocy wszystkim obywatelom. Obecnie procedowany projekt ustawy jest taką pomocą dla wielu. Czy to prawda, że to jest taki uniwersalny projekt, który ma pomagać różnym grupom zadłużonych obywateli?

Pani poseł Bożena Kamińska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Teraz, kiedy mamy kwestie dotyczącą naruszenia prawa Unii Europejskiej, rząd Polski stoi na stanowisku, że trzeba coś naprawić, ale gdzie państwo byliście przez 4 lata?

Dlaczego przez 4 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zadbał o to, żeby to prawo naprawić i pomóc obywatelom polskim? Dlaczego ani premier, ani również pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie pomagał tym obywatelom i tym kredytobiorcom w tych trudnych sytuacjach, nawet przez powołanie pełnomocnika, który profesjonalnie by udzielał im podpowiedzi i rad, co oni w tych kwestiach mają robić? Tak jak pan poseł powiedział, ci ludzie zaciągnęli kredyty. Oni chcą spłacić to, co zaciągnęli, z właściwymi należnymi odsetkami, ale nie trzy razy tyle, co wzięli.

Amber Gold, nieszczelne podatki, teraz dzięki Ministerstwu Finansów mamy na szczęście uszczelnianie finansów publicznych. Jest to problem bardzo poważny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę wyciągnął rękę do Polaków i Polek, a państwo nie widzieliście problemu. Państwo w ogóle nie dostrzegaliście, że finanse publiczne są, winny być pod pewnym rygorem, że Polacy i Polki powinni mieć ochronę ze strony państwa. W ogóle was to nie interesowało. Bardzo dziękuję tutaj rządowi, że podjął się trudnego zadania i że Polacy dochodzą swoich praw w sądach, wygrywają dzięki współpracy z ekspertami, bo przecież te umowy były niejasne, dochodzą swoich praw i uzyskują zadośćuczynienie finansowe. W związku z powyższym mam pytanie do pana ministra: Czy klauzula pozwalająca bankowi na dowolne ustalenie oprocentowania kredytu jest niejasna, niejednoznaczna i nieczytelna, więc nie powinna wiązać konsumentów?

Dziękuję, panie marszałku. Szanowni Posłanki i Posłowie PiS-u! Już w poprzednich wyborach państwa obóz polityczny deklarował rozwiązanie problemu kredytów frankowych. Mówią o tym przedstawiciele frankowiczów, ale mówi też o tym rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, największego sądu w Polsce, zalanego wręcz falą pozwów w sprawie unieważnienia umów kredytowych lub zamiany tych kredytów na kredyty złotówkowe po kursie z dnia wzięcia kredytu. Teraz dowiadujemy się, że koledzy premiera, banksterzy, chcą, by Mateusz Morawiecki stanął po stronie banków, a nie po stronie obywateli i prawa. Prawo bowiem stoi po stronie frankowiczów i tego się boją bankowcy. Proszę się nie dać zwieść bujdom o 60 mld strat sektora bankowego. Banki stracą, to prawda, ale tylko część swoich ogromnych zysków. Proszę pamiętać, banki nie posiadały franków szwajcarskich i nie wypłacały ich swoim klientom.

Czy Prawo i Sprawiedliwość w tej sprawie stanie po stronie obywateli, czy po stronie wielkiego kapitału? Panie premierze, niech pan odpowie Polakom: Dlaczego rząd PiS-u pomaga banksterom, a nie obywatelom? Pani poseł Krystyna Skowrońska.

Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam prostym zewsząd nędza” - a frankowiczom nędza. To cytat z „Krótkiej rozprawy między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem” Mikołaja Reja. To jest o czarowaniu w okresie kampanii, obiecywaniu, że rozwiążemy wszystkie problemy frankowiczów - 500 czy 700 tys. umów. Dzisiaj mogłabym zacytować, powiedzieć, że te obiecanki z kampanii to jest tak jak w przysłowiu: „Pojawia się i znika - taka rola magika” A leżą cztery projekty. Ale warto przedstawić krótki wstęp - dla tych państwa posłów, którzy mówią, że nic nie robiono. W 2006 r. zarówno minister finansów z Prawa i Sprawiedliwości, jak i państwo posłowie mówili, że Polacy mają prawo do ryzyka, i nic nie robiono w sprawie udzielania kredytów frankowych. Dopiero później wstrzymano udzielanie kredytów denominowanych. Wtedy państwo również mieli swojego szefa Komisji Nadzoru Bankowego, a później szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Państwo jeden poprawiacie. W 4 lata PiS nie zrobił nic. Moje pytanie: Jaką opinię ma Komitet Stabilności Finansowej? Jakie są ryzyka w związku z przygotowaniem do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ryzyka kredytowe, płynności, operacyjne, zgodności, utraty reputacji przez banki, kapitałowe?

Nie zrobiliście nic. Poprawiacie tylko ustawę Platformy Obywatelskiej, która niezwłocznie po uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego w stosunku do euro podjęła tę działalność. Zacytuję.

Wysoka Izbo! To, że ci ludzie, którzy są reprezentowani tam, na galerii, wygrywają w sądach, to jest fakt.

W związku z tym chciałbym spytać: Czy macie jakiś plan, plan prawdziwy, plan rzetelny, plan systemowy, jak temu zaradzić? A nie, tak jak w przypadku reprywatyzacji, po prostu będziecie czekać, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo od ustawy reprywatyzacyjnej też uciekacie i jak nie było nic uchwalone, tak nie jest. W związku z tym proszę o odpowiedź: Czy macie, szanowny panie ministrze, jakiś rządowy projekt systematyzujący ten bajzel, który wszyscy tutaj zaraz będziemy mieli zgotowany? Bardzo proszę, pani poseł Paulina Hennig-Kloska. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Tak naprawdę w zasadzie po 4 latach, u schyłku kadencji okazuje się, że żadnych problemów obywateli nie rozwiązaliście w zakresie, w którym składaliście bardzo konkretne obietnice, na bazie poparcia których budował swoją kampanię zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i Prawo i Sprawiedliwość. Frankowicze są ogromnie rozczarowani 4 latami pracy, a ostatnie prace, panie pośle, w podkomisji to była tak naprawdę kpina, bo najpierw przekonywaliście, że rozwiązania, które proponujecie, są doskonałe, są świetne i uratują życie wszystkim pokrzywdzonym przez system bankowy, a potem wycofaliście się z kluczowych dla obywateli rozwiązań, które fakt faktem nie były najlepsze. Bo kadencja się kończy, problem, jak wiele, z którymi szliście do wyborów, kompletnie nie został rozwiązany. Za chwilę może być tak, że faktycznie na poziomie europejskim jakieś decyzje zapadną, ale obywatele w Polsce wciąż muszą ze swoimi indywidualnymi sprawami walczyć w sądach, a nie każdego na to stać. I w ten sposób powodujecie dość spore wykluczenie, bo jak ktoś nie ma pieniędzy na dobrego prawnika, to tej sprawy w sądzie nie wygra.

Dziękuję. Naszej debacie przysłuchuje się z galerii grupa dzieci i młodzieży z gminy Kołaki Kościelne z ks. Piotrem Ćwikłą. Serdecznie witamy. I bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gadowski. Panie Ministrze! Można odnieść takie wrażenie, że propaganda to wasze siła wyborcza i dalej chcecie na fali tych wszystkich obietnic, które obiecywaliście 4 lata, i teraz procedowanych ustaw tę propagandę wyborczą nieść. Panie Ministrze! Ja mam konkretne pytanie do pana.

Czy ta kwota związana z kredytami gospodarczymi spowoduje wzrost wielkości tej kwoty i o ile? Jeśli pan ma takie informacje, to bardzo o nie proszę. Tak się jednak okazuje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo chętnie pomaga bankowcom, a państwo zapomnieliście o obywatelach. Przez lata mówicie o tym, że jesteście blisko obywateli, że chcecie, że rozmawiacie, macie konkretne propozycje, a taki prosty banał pomocy bezpośrednio konkretnemu, wymienionemu z imienia i nazwiska obywatelowi pozostaje dla was jakimś spektrum dalszych uwag i obietnic, a nie realizacji swoich wygłaszanych programów wyborczych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Właśnie niedawno obchodziliśmy czwartą rocznicę spotkania kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, tutaj w Sejmie, ze środowiskiem frankowiczów, podczas którego pan prezydent Duda obiecywał złote góry. Pan prezydent powiedział: Kredyty te mogłyby być przewalutowane według kursu, po jakim były brane. Prezydent ma olbrzymią legitymację, żeby załatwiać trudne sprawy na poziomie państwowym. Nawet padła konkretna data: 3 miesiące po wyborze pan prezydent miał przedstawić taką ustawę. Z dużej chmury mały deszcz, a tak naprawdę wielkie nic.

Szanowni Państwo! Ostatnio mieliśmy wyrok, można powiedzieć, prezydenta Dudy wobec marszałka Kuchcińskiego, który został zawarty w uzasadnieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Totalna krytyka prac legislacyjnych w tej Izbie. Trzeba również, panie pośle Cymański, skrytykować pana pracę w podkomisji, bo ten projekt nieustannie leżakował. Niestety jest to grupa osób, mówię o frankowiczach, bardzo duża grupa osób, która po prostu została ewidentnie przez was oszukana. Troszczą się o system bankowy, a nie o tych, dzięki którym uzyskano poparcie wyborcze w roku 2015. Pan poseł Jan Szewczak. Wysoka Izbo! To jest odpowiedzialność całej klasy politycznej, że ten wrzód nie został już dawno przecięty, jak to się stało w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Sektor bankowy przez lata nie chciał słuchać. Mało tego, wykazywał się wyjątkową arogancją wobec tych, którzy mówili: zróbcie coś, przewalutujcie te kredyty. Rozpiszecie to na lata, będzie po 1 mld rocznie.

Banki się zorientowały, że jednak nie zostanie zalegalizowane bezprawie w tej kwestii.

Pan poseł Błażej Parda. Ja w podobnym tonie, bo ostatnie lata to rekordowe zyski banków. Oni są na tyle bezczelni, że kilka miesięcy temu w mediach podali informację, w zasadzie zapowiedzieli podwyżki opłat nie z tego tytułu, że jest strasznie źle, że bankrutują, tylko dlatego, że Polacy zarabiają trochę więcej, że gospodarka rozwija się troszkę szybciej. Twierdzą, że w związku z tym muszą podnieść opłaty wszystkim Polakom.

Stąd też pytanie: Czy w tej materii rząd planuje jakieś zmiany? On został zablokowany z tego tytułu, że nie było opinii rządu w sprawie tego projektu. Pytanie, czy ta opinia rządu już się pojawiła. Dziękuję bardzo. Pan poseł Henryk Wnorowski. Wysoka Izbo!

Moim zdaniem tutaj nie zanosi się na żaden armagedon.

Ja jestem bardzo zadowolony ze stanowiska rządu. Natomiast wychodzi na to, że ta sprawa, wydawać by się mogło, bardzo trudna, będzie należała do tych, które w jakiejś części rozwiązują się same. Wyrok trybunału, taki, jakiego się spodziewamy, może nam bardzo w tym pomóc.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela wnioskodawców pana posła Andrzeja Maciejewskiego. Panie Marszałku!

Dzisiaj nawet Nowoczesna mówi jak Kukiz. Wielkie gratulacje, że po 4 latach potraficie się nawrócić. Wtedy odrzuciliście nasz projekt, chcieliście odrzucić, ale, jak widzę, edukacja działa. Pierwsza lekcja dla pana posła Gosiewskiego: to jest frank. To jest frank, to już raz pokazywałem, pięć dych polskich.

Jaki algorytm? Jaki kurs? Jak 5 dych przeliczyć na 5 dych? Politolog zakasował gości. Wybaczcie, ale tak to działa. Proszę państwa, druga sprawa, wtedy co do mojego projektu ustawy, który Kukiz składał, BAS wydał taką ciekawą analizę z wnioskiem: Nie wydaje się też celowe obciążenie budżetu państwa kosztami wynikającymi z podjętych błędnych decyzji przez niektórych kredytobiorców oraz banki. Nie jest bowiem rolą państwa ratować każdą grupę, która z powodu podjętych przez siebie decyzji wpadła w kłopoty finansowe.

Dlaczego? Otóż w magiczny sposób w projekcie rządowym w Ministerstwie Finansów pojawia się zmiana w art. 95, która powoduje, że klient staje się jak worek ziemniaków, który można sobie sprzedawać w relacjach między bankiem, funduszem na Cyprze i gdziekolwiek, i nawet o tym nie wie.

Co to znaczy? Ja chciałbym to rozwikłać i chciałbym, żeby w końcu zaczęto na serio mówić o Polakach jako partnerach i o obrońcach. Tak jak Kukiz’15 stał po stronie obywateli, zachęcamy, abyście państwo także stali po stronie obywateli. Będą tam musieli słupki zreflektować swoich zysków na lata. Ale, jeszcze raz powtarzam, we wcześniejszych dekadach zarabiali grube miliardy, nie miliony i wy jako rząd tego na oczy nie widzieliście, ani w Platformie, ani w PiS-ie. To dopiero podatek bankowy pokazał, że te 3 mld z hukiem, większym czy mniejszym, banki mogą oddać do budżetu państwa, mogą nimi wesprzeć budżet państwa. Pytanie, ile miliardów wypłynęło do central bankowych, ile miliardów poszło na boki. My to straciliśmy jako Polacy, a nam się jeszcze ciągle mówi: macie zapłacić 80 mld, 100 mld.

Dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pana

na ten szereg pytań może zacznę po kolei.

Te czasy się skończyły. Mówimy o sprawie Banif Bank, pani poseł. Jeżeli mówimy o historii, to zwracam uwagę, że te kredyty nie zaczęły być udzielane w roku 2015.

Mało tego. Przynajmniej tak mnie poinformowano, państwo posłowie na pewno o tym wiecie, że wczoraj było drugie czytanie tej ustawy na posiedzeniu Sejmu, ustawy mającej pomóc frankowiczom. Jak państwo doskonale wiecie, ci, zajmujący się finansami, to nie jest sprawa prosta, stąd - tak jak była o tym mowa przy pytaniach zresztą - były prace w podkomisji, później były prace w komisji.

Kolejna kwestia.

Kolejna sprawa.

I takie jest stanowisko rządu: jeżeli mamy unijną dyrektywę, jeżeli mamy wdrożenie unijnego prawa, a ta dyrektywa jest wdrożona, to prawo musi być stosowane. Na pytania pana posła Gosiewskiego z racji ich szczegółowości pozwolę sobie udzielić odpowiedzi pisemnej, bo wymagają one zebrania informacji z odpowiednich instytucji.

Czy istnieją rozwiązania. Jeżeli chodzi o projekt Kukiz’15, to z tego, co wiem, było stanowisko rządu przedstawione w formie ustnej.

Co do kwoty 60 mld, o której tutaj wielokrotnie była mowa, to zwracam uwagę, że kwestia musi być badana z innego punktu widzenia.

W związku z tym nie jest to proces prosty i w zależności od tego, jak poszczególne umowy były sformułowane, te zapisy były sformułowane, tak będzie można określić skalę zjawiska, to, czy to jest 60 mld czy mniej, czy więcej. Jeżeli chodzi o art. 95, o którym tutaj była mowa, to była to ustawa związana z implementacją jednej z dyrektyw unijnych. W związku z tym tutaj wchodzi w grę kwestia dostosowania polskiego prawa do dyrektywy unijnej.

Chciałabym zwrócić uwagę pana ministra na pismo generalnego inspektora nadzoru bankowego z 8 lutego 2006 r., który sprzeciwił się zakazowi ograniczania udzielania kredytów walutowych, w tym frankowych. Chciałabym również zadedykować panu ministrowi wypowiedzi m.in. ówczesnej minister finansów pani Zyty Gilowskiej albo pana przewodniczącego klubu Przemysława Gosiewskiego wskazujące w tej dyskusji na potrzebę ograniczenia.

Chciałem tylko powiedzieć, że pani poseł zwróciła uwagę na pismo, które dotyczyło kredytów frankowych, walutowych, a nie tzw. kredytów walutowych czy tzw. kredytów frankowych.

Już wtedy się orientowaliście, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem, i postanowiliście troszkę nagiąć, zmienić to Prawo bankowe, żeby te kredyty denominowane i indeksowane również traktować jako kredyty walutowe. Jeszcze raz powtarzam: nie ma najmniejszego sensu się wzajemnie oskarżać, pani poseł.

Dobrze. Dziękuję państwu bardzo. Ta wypowiedź kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 3551 i 3591) Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawienia w imieniu Komisji Finansów Publicznych sprawozdania tejże komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk nr 3551. Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 r., zgodnie z art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu, skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 r. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył powyższy projekt ustawy. Pragnę nadmienić, że w trakcie prac komisji nie została złożona żadna poprawka. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Głos ma pan poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Wczoraj do Sejmu wpłynął, a właściwie w pierwszym czytaniu był analizowany, przedmiotowy projekt z druku nr 3551, dotyczący propozycji rządowej wprowadzenia stawki zerowej PIT, podatku dochodowego od osób fizycznych, dla osób do 26. roku życia.

Po pierwsze, jeśli chodzi o konstytucyjność projektu, to w uzasadnieniu rządowym mamy powołanie na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z maja 1996 r., które wyraźnie mówi, że rząd, że ustawodawca, że Sejm mają pełną swobodę kształtowania tego typu relacji i wybierania beneficjentów polityki podatkowej. Wydaje się dość oczywiste, że zasada, którą przyjęto w tym programie, mieści się w ramach tak określonego pola manewru, jakim dysponuje ustawodawca.

Po pierwsze, faktem jest jedna zasadnicza sprawa.

Cieszę się bardzo z tego powodu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma zdecydowanie lepszą ofertę niż nasi poprzednicy.

My mamy rzetelne rozwiązania, które są oczekiwane przez młodych ludzi, i znam już wielu młodych ludzi, którzy bardzo cieszą się na myśl o wprowadzeniu tej regulacji. Bardzo proszę, pani poseł Marta Golbik, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Z przykrością muszę stwierdzić, że w trakcie prac w komisji żadna z wątpliwości zarówno naszych jako Platformy Obywatelskiej, jak i związków przedsiębiorców, związków samorządowych nie została rozwiana, a wręcz nie odpowiedziano na podstawowe pytania.

A tymczasem mamy sytuację, w której osoba do 26. roku życia, która jest zatrudniona na umowę o pracę, będzie miała zwolnienie z PIT, a osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, będzie miała podwyższony ZUS w przyszłym roku o 120 zł. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości nie promuje osób przedsiębiorczych.

Muszę odnieść się do słów przedmówcy z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o tym, że to jest świetny program, a opozycja programu nie ma. Szanowni państwo, 2 lata zostały zmarnowane od momentu, kiedy Platforma Obywatelska złożyła program „Wyższe płace”, który zakładał podwyżki wynagrodzeń na rękę tym wyższe, im mniej ktoś zarabia, program, który nie ucinał nagle zwolnień i podwyżek zarobków w momencie, kiedy osoba kończy 26 lat, w końcu program, który był skierowany do wszystkich, a nie jedynie do pewnej grupy osób, które w momencie ukończenia 26. roku życia nagle przestaną z tych zwolnień korzystać, i co najważniejsze, z państwowego punktu widzenia, program, który system podatkowy upraszcza, a nie komplikuje. Młode osoby znów będą musiały się zastanawiać - już się zastanawiają - jak skorzystać z największej ilości ulg, a nie o to powinno nam chodzić.

Musimy pamiętać, że wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko interesariuszy i osób, które te ulgi otrzymają, ale przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego.

To o 13,5 mld zł mniej wpływów do Skarbu Państwa, ale i o 11,8 mld zł mniej wpływów do samorządów, a to oznacza mniej środków na wydatki publiczne skierowane do mieszkańców, samorządów, na żłobki, przedszkola. To jest bardzo duży problem. Dlaczego wprowadzane są rozwiązania, które nie są dla wszystkich nawet w zakresie tej samej kategorii wiekowej? Szanowni Państwo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska składa poprawkę, która ma na celu uwzględnienie również osób zatrudnionych na umowę o dzieło oraz osób samozatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, tak aby wszyscy byli traktowani równo. Naszej debacie przysłuchuje się grupa gości z Hartowca, z powiatu Działdowo. Serdecznie państwa witamy.

Jeżeli ktoś z państwa chce się jeszcze zapisać, zapraszam. Pan poseł Michał Szczerba. Nie widzę. Pani poseł Zofia Czernow.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! To prawda, że rząd chce pomóc młodym ludziom wchodzącym w dorosłe życie i ułatwić im start, ale dlaczego tej pomocy odmawia się też młodym ludziom, w tym samym wieku, którzy nie chcą podejmować pracy na umowę zlecenie, tylko chcą pracować na własny rachunek? Mają inicjatywę, mają pomysły i ta przedsiębiorczość powinna być promowana. Powinniśmy się cieszyć z tego, że coraz więcej naszych obywateli chce działać na własny rachunek, podejmując różne inicjatywy, otwierając swoje własne firmy.

Przecież powinniśmy promować właśnie taką przedsiębiorczość.

Pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytanie: Czy ministerstwo próbowało oszacować, jak dużej grupy młodych ludzi pracujących w tzw. szarej strefie mogą dotyczyć wprowadzone rozwiązania? Dziękuję. Dziękuję. Wysoka Izbo!

Mam tutaj na myśli młodych lekarzy.

utraty wpływów do budżetu z tytułu podatku dochodowego dla osób zatrudnionych na umowę o dzieło, wypełniających umowę o dzieło, albo osób prowadzących działalność gospodarczą są wysokie, istotne? Jaką stanowią kwotę? Zdaję sobie sprawę z tego, że tamtędy mógłby pójść dodatkowy strumień obciążający dochody budżetu państwa i stąd wynikała pewna ostrożność w zawężeniu tych ram beneficjentów - dla mnie jest to absolutnie zrozumiałe.

I wydaje mi się, że powinniśmy rzetelnie pokazać to obywatelom, dlaczego nie mogliśmy iść taką drogą. Prawo i Sprawiedliwość rozwiązuje problemy systemowo, zwracając się do wielomilionowych grup zawodowych, branżowych i społecznych. Tak samo jest w tym przypadku - 2,2 mln osób staną się beneficjentami tej ustawy, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zapraszam podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana Piotra Nowaka. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Celem tej ustawy, tego projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im właśnie wejścia na rynek.

Ponadto ten wiek 26 lat pojawia się w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, zgodnie z którymi osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jeżeli są uczniami lub studentami, do ukończenia tego roku życia.

Pojawiła się również taka narracja, wydaje nam się, nie do końca sprawiedliwa, mówiąca, że rząd dyskryminuje samozatrudnionych, dyskryminuje przedsiębiorców.

W stosunku do tej pierwotnej propozycji po konsultacjach i rozmowach zostało to rozszerzone o umowy zlecenia, które są częstą formą zatrudnienia wśród młodych. Jednocześnie celem projektu nie jest wsparcie każdej formy aktywności zarobkowej młodej osoby, a wyłącznie wzrost aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach stabilnych i najbardziej popularnych form zatrudnienia, do których ma zastosowanie umowa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Stąd też projekt nie obejmuje ulgą dla młodych przychodów z umowy o dzieło oraz działalności gospodarczej. Umowa o dzieło nie stanowi bowiem podstawy prawnej zatrudnienia. Co się zaś tyczy działalności gospodarczej, w tym m.in. jednoosobowej, która tu była podkreślana, to przychody te mogą być już dziś opodatkowane podatkiem PIT na preferencyjnych zasadach, to jest według liniowej stawki podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyboru tych form opodatkowania nie mają natomiast pracownicy lub zleceniodawcy, zleceniobiorcy, przepraszam, nieprowadzący działalności gospodarczej. Stąd projektowane wsparcie kierowane jest właśnie do tej grupy podatników. Ponadto w ostatnim czasie rząd wprowadził dla przedsiębiorców wiele dodatkowych rozwiązań, które skutecznie obniżają ich obciążenia fiskalne. Postaram się wymienić pięć podstawowych. Jest to ulga na start. To jest wsparcie dla przedsiębiorców. Od 30 kwietnia 2018 r. przedsiębiorcy mogą nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przez 6 miesięcy, natomiast po 6 miesiącach przez kolejne 24 miesiące są składki dużo niższe. Wprowadzono również mały ZUS. Od 1 stycznia br. przedsiębiorcy mogą opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od faktycznych przychodów. Kolejne było to, że od 1 stycznia 2019 r. umożliwiono szybkie rozliczenie straty poprzez wprowadzenie prawa do obniżenia jednorazowego dochodu z danego źródła przychodów, do kwoty nieprzekraczającej aż 5 mln zł. Również od 1 stycznia br. wprowadzono możliwość zaliczania do kosztów wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, należnego z tytułu np. stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

To również wspiera innowacyjność naszej gospodarki. Dlatego nieprawdziwe są stwierdzenia, że rząd w tym przypadku dyskryminuje samozatrudnionych czy przedsiębiorców.

rozpatrzyła projekt ustawy wdrażający dwie dyrektywy unijne do krajowego porządku prawnego. Projekt po rozpatrzeniu przez komisję, z jedną poprawką legislacyjną zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne, dotyczącą art. 1 pkt 1, został przyjęty bez głosów sprzeciwu. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Z tego względu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim zawierający regulacje wdrażające do polskiego prawa przepisy obu wzmiankowanych dyrektyw. Kluczowe dla bezpieczeństwa statków pasażerskich rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim dotyczą m.in. zapewnienia morskim służbom ratowniczym natychmiastowego dostępu do danych osób podróżujących na statkach pasażerskich, co jest niezwykle istotne w przypadku prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych pojedynczych pasażerów lub członków załóg tych statków, jak również w przypadku prowadzenia tzw. masowych operacji ratowniczych dotyczących całego statku pasażerskiego oraz wszystkich osób znajdujących się na jego pokładzie. Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa statków pasażerskich mają również zawarte w projekcie ustawy regulacje dotyczące systemu inspekcji statków pasażerskich typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich uprawiających żeglugę na liniach regularnych. Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa osób podróżujących statkami pasażerskimi, nowelizowane przepisy będą miały również pozytywny wpływ na funkcjonowanie sektora morskiego transportu pasażerskiego, m.in. poprzez zniesienie dublujących się wymogów i ujednolicenie wymagań dla statków pasażerskich niezależnie od ich przynależności. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako poseł sprawozdawca rekomenduję przyjęcie przedmiotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Dziękuję. Ja również dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Głos ma pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałam przedstawić stanowisko w sprawie druku nr 3540, a mianowicie projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim wraz z poprawkami, które panu marszałkowi przekażę w imieniu mojego klubu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim zawiera szereg zmian prawnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich obszarach morskich. Przede wszystkim projektowana ustawa zawiera przepisy wdrażające do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa statków pasażerskich.

Kierunek zmian w prawie europejskim, wyznaczony m.in. przez potrzebę ciągłego usprawniania procedur działania morskich służb ratowniczych, został odzwierciedlony również w poprawkach, które chciałabym złożyć. Są to cztery poprawki, a proponowane zmiany dotyczą funkcjonowania jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, służby powołanej w celu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu oraz wykonywania innych zadań związanych z bezpieczeństwem morskim. Pierwsza zmiana jest wprowadzana na wniosek pracowników brzegowych stacji ratowniczych oraz Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego MSPiR. Zmiana umożliwi pełnienie w tych jednostkach 24-godzinnych dyżurów, obecnie dyżur trwa 12 godzin, podczas których ratownicy, inspektorzy pozostają w pogotowiu ratowniczym, prowadzą nasłuch radiowy i wykonują zadania związane z utrzymaniem w gotowości operacyjnej sił i środków, którymi dysponuje MSPiR. Analogiczny system pracy funkcjonuje od dawna m.in. w straży pożarnej czy w zakładowych służbach ratowniczych, a więc w formacjach o zbliżonej specyfice zadań. Rozwiązanie to sprawdza się w praktyce, wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników, a pracodawcom daje niezbędną elastyczność przy planowaniu pracy i odpoczynku personelu ratowniczego. Druga proponowana zmiana przepisów usprawni działania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i pozwoli uniknąć sytuacji absurdalnych, jak np. pozostawienie statku ma łasce żywiołu po ewakuacji jego załogi lub wielogodzinne pozostawianie statku ratowniczego w tzw. asyście przy uszkodzonej jednostce, na wypadek gdyby pojawiło się zagrożenie życia jej załogi na skutek zmiany pogody lub rozwoju awarii. 3. poprawka również stanowi o zmianach w ustawie, ale biorąc pod uwagę, że MSPiR została powołana w celu wykonywania nieodpłatnego ratownictwa życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska morskiego, natomiast ratownictwo morskie w rozumieniu ustawy Kodeks morski jest działalnością odpłatną, konieczne jest uregulowanie w ustawie o bezpieczeństwie morskim zasad zwrotu do budżetu państwa kosztów działalności służby wykraczającej poza jej pierwotne, statutowe zadania. 4. poprawka dotyczy zmiany brzmienia art. 8 projektu ustawy, określającego termin wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Zgodnie z proponowanym nowym brzmieniem art. 8 projektu zmiany dotyczące funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wejdą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Projektowane zmiany prawne mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich osób uprawiających żeglugę na polskich obszarach morskich, m.in. poprzez harmonizację wymogów dotyczących statków pasażerskich jak również przez usprawnienie funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Aziewicz, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim wdraża do polskiego prawa regulacje dwóch dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa na statkach pasażerskich. Biorąc pod uwagę przepisy unijne, zaproponowane rozwiązania zapewnią jednolite zasady przeprowadzania inspekcji na statkach pasażerskich typu ro-ro, chodzi o statek pasażerski przystosowany do wtaczania i wytaczania pojazdów drogowych lub szynowych, oraz na szybkich statkach pasażerskich przewożących powyżej 12 pasażerów w trakcie uprawiania żeglugi na linii regularnej. Chodzi m.in. o serię podróży statku wykonywanych w celu obsługi ruchu między tymi samymi dwoma portami lub większą liczbą tych samych portów. Celem nowych przepisów jest włączenie inspekcji przeprowadzanych na tego typu statkach w system inspekcji przeprowadzanych przez państwo bandery na statkach o polskiej przynależności, a przez państwo portu - na statkach pływających pod obcą banderą. Zaproponowano również przepisy, które umożliwią sprawniejsze przekazywanie informacji o liczbie i tożsamości osób znajdujących się na pokładzie statku, z uwagi na ich szczególne znaczenie dla skuteczności prowadzonych akcji poszukiwawczych i ratunkowych. Rozwiązania te pozytywnie wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 21 grudnia 2019 r., ponieważ do tego dnia państwa Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć przepisy dyrektyw pasażerskich. Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w dniu 3 lipca 2019 r. Jeżeli chodzi o poprawki zgłoszone przez panią poseł Arciszewską, to odniesiemy się do nich w trzecim czytaniu. Dziękuję za uwagę. Pana posła Kobylarza nie ma. Pan poseł Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów jest za kontynuowaniem prac legislacyjnych, bowiem - jak już stwierdził mój przedmówca - ten rządowy projekt przedłożony do pierwszego czytania na posiedzeniu komisji nie wzbudził czy nie wywołał, nie spowodował w czasie prac różnicy zdań. Nie było kontrowersji.

Stąd też te dwa głównie wskazywane obszary dotyczą i pasażerów, i zachowania stosownego, dobrego, na wysokim poziomie stanu technicznego statków, które służą do przewozu ludzi. To uważamy za właściwe i dobre.

Co do ewidencji pasażerów to sprawa jest oczywista i jasna.

Dochodzą do tego sytuacje awaryjne.

Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Mam pewną wątpliwość, którą chciałbym wyjaśnić, dotyczącą przesyłu danych. Czy wprowadzenie nowej, mówiąc w cudzysłowie, końcówki systemu po stronie obsługi jednostek pływających będzie monitorowane przez ministerstwo pod kątem właściwego zaprojektowania bezpieczeństwa przesyłu danych, tak aby cały system pozostał bezpieczny i odporny na ingerencję z zewnątrz? Pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Ministrze! W art. 103 opiniowanego projektu ustawy przewiduje się obowiązek rejestracji danych o osobach odbywających podróż morską na jachtach komercyjnych oraz ich przekazywania przy użyciu aplikacji mobilnej do pojedynczego punktu kontaktowego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie!

Wiąże się to z pytaniami, które zostały przed chwilą zadane.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projektu do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedłożyła sprawozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, druk nr 3501. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 26. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (druki nr 3519 i 3567) Proszę pana posła Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z posiedzenia w dniu 3 lipca tego roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, druk sejmowy nr 3567. Na wstępie chciałbym podkreślić, że po raz pierwszy od 1990 r. rządzący zajęli się sprawą modernizacji Służby Więziennej.

Dodatkowe środki finansowe będą rozdysponowane w 2019 r. na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wysoka Izbo! Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Klub Prawo i Sprawiedliwość popiera nowelizację ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” Zależy nam na tym, aby Służba Więzienna działa lepiej. Zależy nam także na tym, aby funkcjonariusze Służby Więziennej zarabiali lepiej. Przypomnę, że ustawa z 2016 r. przewidywała m.in. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych, czyli chodziło, z jednej strony, o sprawy funkcjonariuszy Służby Więziennej, z drugiej strony, o sprawy pracowników cywilnych pracujących w zakładach karnych. Środki, które były zaplanowane na realizację tego, nie uwzględniały tych zmian, o których mówił pan poseł Matusiewicz, i były skalkulowane stosownie do warunków, które panowały w roku 2017, ale w związku z tym, że doszło do zwiększenia liczby etatów w służbie - jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, to tu chodzi o 438 etatów, jeśli chodzi o pracowników cywilnych, to jest to 125 etatów - potrzebna jest korekta, potrzebna jest zmiana ustawy.

Ten wzrost wynagrodzeń w przypadku funkcjonariuszy wynosi 438 zł, w przypadku pracowników cywilnych - 300 zł. Reasumując, dobrze, że ta nowelizacja została przygotowana. Klub Prawo i Sprawiedliwość ją wspiera i na pewno w kolejnych latach będzie starał się o poprawę warunków pracy w Służbie Więziennej. Dziękuję. Pana posła Michała Szczerby nie widzę. Zapraszam pana posła Andrzeja Maciejewskiego, Klub Poselski Kukiz’15. Wysoka Izbo!

Cieszymy się, że pochylamy się nad ważnym zagadnieniem, zapewniając szacunek, godność i prestiż pracy w Służbie Więziennej.

Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów przedstawić nasze stanowisko w sprawie sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” Omawiany projekt ma w założeniu zapewnić podstawy prawne do zaangażowania dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację programu modernizacji Służby Więziennej w związku ze zwiększeniem limitu etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej w latach 2017–2018. Zakłada się zwiększenie liczby etatów o 438 w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 125 w odniesieniu do pracowników cywilnych. I tu trzeba się zgodzić z założeniami projektodawców, bo faktycznie ilość etatów, jeśli chodzi o więziennictwo, wymaga zdecydowanych działań.

Więcej środków ma trafić na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Sytuacja w tej materii zmieniła się w ubiegłym roku, kiedy to wraz ze zmianą przepisów dozór elektroniczny trafił w ręce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Po zmianie przepisów Służba Więzienna przyjęła obowiązki patroli obsługujących cały system wykonywane wcześniej przez firmę prywatną wyłonioną w drodze przetargu. Wobec przejęcia nadzoru elektronicznego przez Służbę Więzienną konieczne jest odpowiednie przystosowanie tej formacji do przejęcia nowych obowiązków zarówno pod względem kadrowym, jak i finansowym. Chodzi również o zabezpieczenie środków na poprawę konkurencyjności wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, co jest uzasadnione w sytuacji, kiedy stawki na rynku pracy szybko rosną.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś z państwa chce się jeszcze zapisać do głosu, zapraszam. Głos ma pan poseł Michał Szczerba. Nie ma. Bardzo proszę, pan poseł Piotr Pyzik. Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o system dozoru elektronicznego. Powierzenie Służbie Więziennej nadzoru nad tym systemem to krok oczywisty. Obywateli interesuje również strona finansowa tego przedsięwzięcia. Dodatkowe etaty funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej to dodatkowe koszty dla budżetu państwa. Jednocześnie następuje oszczędność w postaci braku ponoszenia kosztów dotychczasowego systemu, w którym zadania te wykonywała wynajęta firma. Bardzo proszę w imieniu wyborców o informację, jakie oszczędności udało się uzyskać z tego tytułu. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Gawron. Zapraszam. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonują trzy zakłady karne.

Z zapisów ustawy wynika również, że w większości te środki pójdą na zwiększenie wynagrodzeń. Mam takie pytanie, panie ministrze: Czy w 2019 r. była już podwyżka dla pracowników Służby Więziennej, dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych? Mówi się też w ustawie, w uzasadnieniu o motywacyjnym systemie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wysoka Izbo! Ustawa ta z pewnością wpisuje się w „Program modernizacji Służby Więziennej” Chciałbym dopytać, jak wyglądają plany budowy nowych więzień, nowych pawilonów. Czy planowane zwiększenie etatów Służby Więziennej jest wystarczające w kontekście rozbudowy więzień? Dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Zapraszam sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Michała Wójcika.

Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za wszystkie pytania, także za odniesienie się do projektu ustawy, ważnego projektu, który jest kolejnym krokiem wzmacniającym Służbę Więzienną.

Oczywiście ta ustawa, ten projekt przewiduje sfinansowanie określonych etatów w liczbie 313, które wynikają ze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego i możliwości kierowania osób skazanych poza granicami Polski do polskich więzień, do polskich jednostek penitencjarnych.

Jest kilkaset takich osób. Oczywiście działa to w dwie strony. I jest 250 etatów, zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych, jeżeli chodzi o system dozoru elektronicznego, o który pytał pan poseł Pyzik, któremu chciałbym odpowiedzieć, że istotnie, tak jak pan poseł raczył zauważyć, dobrze, że system dozoru elektronicznego jest w tej chwili całkowicie zależny od służby czy też nadzorowany przez Służbę Więzienną. Jeszcze do niedawna była taka sytuacja, w której podmioty prywatne decydowały o tym, jak w terenie realizowane są określone sprawy związane z systemem dozoru elektronicznego, a tylko centrala monitorująca była w Warszawie.

Pytał się pan poseł o kilka spraw, m.in. o sprawę dotyczącą kosztów. Otóż na początku chcę powiedzieć, że jest ok. 5 tys. osób w tym systemie dozoru elektronicznego.

W tej nowelizacji, która w tej chwili była procedowana, niedawno była procedowana w Sejmie, w Senacie, znajduje się taki przepis, który dotyczy również systemu dozoru elektronicznego. Przypomnę, że w obecnej sytuacji, jeszcze w obecnym stanie prawnym jest to taki system, w którym musiałoby nastąpić skazanie do 12 miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście osoba skazana miała prawo czy ma prawo ciągle wystąpić z wnioskiem o to, żeby zastosować system dozoru elektronicznego wobec niej. Jeżeli sąd penitencjarny wyrazi taką zgodę i tak rozstrzygnie, to ten system dozoru elektronicznego będzie zastosowany, czyli krótko mówiąc, jest to opaska elektroniczna, która pozwala odbywać karę pozbawienia wolności w warunkach wolnościowych. To też jest taki sygnał, bo w ostatnim czasie w mediach przetoczyła się bardzo gruntowna, bardzo szeroka, głęboka dyskusja na temat nowelizacji Kodeksu karnego. Jakoś nikt nie dostrzegł tego, że tam przecież również dotyka to kwestii systemu dozoru elektronicznego. Oczywiście w czasach naszych poprzedników w ogóle doszło do załamania tego systemu, bo przyjęto zupełnie inne regulacje. Dopiero kiedy nastąpił rząd dobrej zmiany, stwierdziliśmy, że trzeba przywrócić możliwość, żeby osoby skazane na karę pozbawienia wolności, a nie ograniczenia wolności mogły odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego. To jest według mojej wiedzy ok. 350 zł miesięcznie, przy czym rozmawiałem tu przed chwilą z panem dyrektorem z Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, który mówił, że te koszty mogą być nieznacznie wyższe. 10 razy mniej. Normalnie kara miesięczna, koszt wykonania takiej kary w jednostce penitencjarnej to jest ok. 3,5 tys. zł.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Ogłaszam 5 minut przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druki nr 3520 i 3578) Proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, druki nr 3520 i 3578. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym. Projektowana regulacja wprowadza zmianę polegającą na umożliwieniu osobom podjęcie kształcenia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, jak również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze do 6 dni rocznie np. celem uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach naukowych i kursach naukowych. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą nie jest możliwe prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo w formie niestacjonarnej, co z kolei jest możliwe na jednolitych studiach magisterskich na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Standardy kształcenia dla kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo określają m.in. czas trwania studiów, minimalną liczbę godzin zajęć i praktyk, a także szczegółowe efekty kształcenia, niezależnie od formy studiów. W związku z tym projektowana zmiana gwarantuje, że treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz liczba godzin na tych studiach będą takie same jak w przypadku studiów prowadzonych w formie stacjonarnej. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej będą mogły podejmować przede wszystkim osoby pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodzie pielęgniarki lub położnej. Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku: pielęgniarstwo również przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. przez ratowników medycznych czy opiekunów medycznych. Powyższa zmiana wpłynie na realizację jednego z priorytetów przyjętych w dokumencie o charakterze strategiczno-wdrożeniowym pn. „Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”, w tym celu operacyjnego, jakim jest wspieranie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych, oraz Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce z 2017 r.

Zgodnie ze strategią jednym z priorytetów jest podjęcie działań na rzecz zwiększenia liczby kandydatów przyjmowanych na kierunki: pielęgniarstwo i położnictwo przy uwzględnieniu jakości kształcenia.

Drugą istotną zmianą, jaką zawiera projekt ustawy, jest wprowadzenie możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę lub położną celem stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach innych niż dotychczas możliwe, tj. szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego, a także celem odbycia kształcenia podyplomowego bez skierowania, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy - w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Projekt ustawy jest jednym z elementów mających poprawić w przyszłości sytuację dotyczącą liczby pracujących pielęgniarek i położnych. Temu celowi służą działania rządu polegające na zwiększeniu liczby uczelni, na których kształci się na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, zwiększeniu liczby przyjmowanych studentów, zwiększeniu środków przeznaczonych na kształcenie, poprawie warunków wynagradzania, uczynieniu zawodu pielęgniarki i położnej atrakcyjnym. W trakcie procedowania projektu ustawy zgłoszono i przyjęto 3 poprawki. Cały projekt, wraz z poprawkami, został przyjęty przez komisję bez głosu sprzeciwu. Dlatego w imieniu komisji wnoszę o poparcie projektu ustawy przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Otwieram dyskusję. Głos ma pani poseł Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, druki nr 3520 i 3728. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Ustawa zakłada, że kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej będą mogły podejmować osoby również pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w ww. zawodzie. Podkreślić pragnę, że projektowana zmiana gwarantuje, iż treści programowe studiów I stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz liczba godzin na tych studiach będą takie same jak na studiach stacjonarnych na tych kierunkach. Druga zmiana w ustawie zakłada wprowadzenie dodatkowego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w innych formach niż te, które określone są w art. 66 ust. 1 ustawy - tj. szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy dokształcające - w wymiarze do 6 dni roboczych. Urlop ten jest płatny zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Należy podkreślić, że zmiana wprowadzająca płatny urlop szkoleniowy jest realizacją porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a ministrem zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany wprowadzone w ustawie są bardzo korzystne społecznie i zgodne ze „Strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” Zmiany te przyczynią się do zwiększenia liczby osób kształcących się w zawodach pielęgniarki i położnej, a to ma ogromny wpływ na podniesienie jakości ochrony zdrowia. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość rekomenduje omawiane zmiany w ww. ustawie i głosować będzie za ich przyjęciem.

Wysoka Izbo! Jaka sytuacja kadrowa jest w systemie ochrony zdrowia, chyba każdy z nas dobrze wie. Mamy niedobory nie tylko pielęgniarek i położnych, mamy niedobory całej kadry medycznej. A prawdą oczywistą jest to, że pacjentów nie będą leczyć mury szpitali, łóżka czy nie będą leczyć najnowocześniejsze urządzenia. Dlatego to jest krok w bardzo dobrym kierunku, że rząd reaguje, na razie w przypadku jednego zawodu medycznego, a właściwie dwóch, i otwiera możliwości kształcenia większej ilości chętnych do podjęcia tego zawodu. Bo faktycznie ta ustawa ma dwa główne kierunki, czyli zwiększenie ilości studiujących i, być może, trafiających do zawodu, a z drugiej strony - to jest też jeszcze rzecz nie do niezauważenia - dajemy szansę, aby pielęgniarki i położne miały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Nie ma co ukrywać, że fachowość tej kadry, która dość często jest lekceważona i niedoceniana, fachowość pielęgniarek i położnych siłą rzeczy odciąża lekarzy. To z punktu widzenia pacjenta, zwłaszcza pacjenta, który ma doświadczenie w chorowaniu, jeśli tak mogę powiedzieć.

Kwestia pielęgniarek jest rzeczą, którą, powiedzmy, w tej chwili można najłatwiej zrobić, bo dużo trudniejsza jest kwestia lekarzy.

Tego, co w tej chwili mówię, nie mówię bezpodstawnie, bo w moim rodzinnym mieście, czyli w Kaliszu, jest kierunek pielęgniarski w szkole wyższej i niestety nie jest to dobry wynik procentowy, jeśli chodzi o to, ile absolwentek, absolwentów trafia do zawodu, pomimo że jest świetna współpraca z kaliskim szpitalem i naprawdę jest dobry poziom kształcenia. Dlaczego tak się dzieje? Jest Polska A, czyli wielkie miasta, Warszawa, Poznań, gdzie pielęgniarki tak naprawdę nie mogą się opędzić od ofert pracy i mogą być roszczeniowe w tym przypadku, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Dlatego że jest pewien problem w przeznaczonych pieniądzach, na POZ chociażby. POZ, żeby utrzymać racjonalność współpracy z pacjentem, musi mieć te dwa, trzy etaty, a pieniądze, które otrzymuje, tak naprawdę starczają na jeden etat, jeśli chcemy tę pielęgniarkę dobrze wynagradzać. I nie dziwmy się, że pielęgniarki w tym przypadku szukają innych pomysłów na zarabianie pieniędzy, a czasami po prostu zasilają konkurencyjne - bo jest to konkurencja - inne systemy ochrony zdrowia, w innych krajach. I to jest paranoja, dlatego że my kształcimy za nasze pieniądze, z naszych podatków kadrę, która siłą rzeczy, przy braku motywacji w Polsce, wyjeżdża za granicę. Samo to, że zwiększymy łatwość kształcenia poprzez studia niestacjonarne i damy możliwość dokształcania się pielęgniarkom, to bardzo dobrze, ale to za mało.

Jest późno, ale jeszcze nie za późno. Dziękuję bardzo.

Zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych jest bezsprzecznie potrzebne i powinno stanowić jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Biorąc pod uwagę fakt, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce to prawie 51 lat, oraz że z końcem przyszłego roku aż 44% z nich uzyska prawa emerytalne, to trzeba mieć świadomość, że bez podjęcia realnych działań sytuacja w ochronie zdrowia będzie krytyczna. Procedowany dzisiaj rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ma właśnie przeciwdziałać temu kryzysowi. Ustawa ta wprowadza bowiem możliwość kształcenia niestacjonarnego na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo. Z pozoru wydaje się to dobre rozwiązanie, które pozwala na podjęcie studiów większej liczbie osób. Jednak, jak słusznie zauważa Biuro Analiz Sejmowych oraz, co ważniejsze, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, problemem może być zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia. Jak wynika obecnie z wymogów określonych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 9 maja 2012 r., studenci, którzy zdecydowali się na studia w trybie stacjonarnym, muszą wziąć udział w 1100 godzinach zajęć praktycznych oraz odbyć 1200 godzin praktyk zawodowych. Wymagania te mogą być bardzo ciężkie do spełnienia w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, którzy na co dzień pracują zawodowo. Kolejnym krokiem zatem może być zmiana wspomnianego rozporządzenia regulującego tę liczbę godzin, obniżając ją do bardziej urealnionego poziomu dla studentów zaocznych. To rozwiązanie doprowadzi jednak do obniżenia poziomu kształcenia naszych pielęgniarek, a przecież chcemy, żeby pacjenci mieli zapewnioną najlepszą z możliwych opiekę. Szanowni Państwo! Chcąc zwiększyć liczbę pielęgniarek i położnych w Polsce oraz przekonać młodych ludzi do podjęcia się tak odpowiedzialnej pracy, w pierwszej kolejności powinniśmy zagwarantować im godne warunki pracy i płacy. Prawodawca w tym projekcie podjął taką próbę, bo tak należy ocenić dodatkowe dni płatnego urlopu szkoleniowego, ale tradycyjnie wszystkimi kosztami, z którymi wiąże się ten płatny urlop, obarcza szpitale, czyli de facto podmioty, które nie są stroną porozumienia. To jak w soczewce obrazuje metody rządzenia w dzisiejszej Polsce: my obiecujemy, a zapłacą inni. Sytuacja ta jest o tyle niebezpieczna, że ekwiwalent za ten urlop nie jest uwzględniony w żadnych planach finansowych, a w przypadku dużych ośrodków te koszty mogą być znaczące. Pogłębi to kryzys finansowy wielu placówek. Podsumowując, projektodawca chce rozwiązać problem niedoboru pielęgniarek i położnych tylko pozornym zwiększeniem dostępu do kształcenia na tych kierunkach lub poprzez obniżenie poziomu edukacji na skutek zmniejszenia liczby godzin zajęć praktycznych. Koszty płatnych urlopów szkoleniowych, które mocą tych przepisów mają przysługiwać pielęgniarkom i położnym, przerzuca się na dyrektorów szpitali. Rozumiem że rekordowe zadłużenie polskich szpitali nie robi na ministrze zdrowia żadnego wrażenia i chce śrubować ten bardzo niechlubny rekord. Bo przecież płatne urlopy to będą dodatkowe koszty nieplanowane na początku roku i nieuwzględniane przy wyliczaniu ryczałtu. Co gorsze, przypuszczam, że w przyszłości ten fakt również będzie ignorowany przy wyliczeniach środków przyznawanych szpitalom przez NFZ. Takie gospodarowanie środkami finansowymi w ochronie zdrowia spowoduje w niedługim czasie bankructwo wielu szpitali, zamykanie kolejnych oddziałów, co znacząco ograniczy dostęp do ochrony zdrowia wszystkim pacjentom, także nam i naszym bliskim. Jeśli w środku roku rozliczeniowego wprowadzamy przepisy, które są kosztowne dla wielu placówek, to kwestią uczciwości jest finansowanie ich w całości, a dopiero potem rozpoczęcie negocjacji z placówkami w zakresie współfinansowania przez nie tych pomysłów. Pomimo mojego szczerego poparcia dla postulatów pielęgniarek, doceniając ich pracę i zaangażowanie, które sam obserwuję na moi oddziale, to nie mogę zgodzić się na przyjęcie projektu obciążającego kosztami stronę, która ani nie brała udziału w dyskusji o tych rozwiązaniach, ani nie jest stroną zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. porozumienia, w efekcie którego powstała ta ustawa. W związku z powyższym wstrzymam się od głosu.

Pani Minister! Mam następujące pytanie: Czy w związku z faktem, że na wspólnotowym rynku pracy istnieją wciąż bardzo duże dysproporcje pod względem wynagrodzeń w zawodach pielęgniarskich, proponowane rozwiązanie jest wystarczające do osiągnięcia zakładanego skutku w postaci wskaźnika liczby pielęgniarek na poziomie średniej OECD? W gruncie rzeczy mógłbym poprzestać tylko na tym pytaniu, natomiast doświadczenie z kadencji poprzedniej i z tej kadencji wskazuje na to, że warto zapytać jeszcze o następujące kwestie. Kwestia odbiurokratyzowania pracy pielęgniarek, żeby oprócz ciężkiej, bardzo ciężkiej pracy, którą wykonują, nie musiały wykonywać jakichś rzeczy biurowych, nazwijmy to tak subtelnie. Kwestia średniego wieku pielęgniarek wskazuje na jedną rzecz, a mianowicie - przepraszam, że tak brzydko to nazwę - wymieranie tej przestrzeni naszej służby zdrowia, na co wskazuje nie tylko średni wiek pielęgniarek, ale również to, co dzieje się ze szkołami pielęgniarskimi.

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Starostwo Powiatowe w Wieluniu jako organ prowadzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu podjął w tym roku inicjatywę wraz z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu zmierzającą do tego, ażeby właśnie w Wieluniu otworzyć wydział zamiejscowy pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych. W związku z powyższym mam pytanie do pani minister. Czy procedowane rozwiązania i zmiany wpłyną jakoś na rekrutację roczników studentów pielęgniarstwa, jak również czy wprowadzona zmiana wpłynie na jakość kształcenia pielęgniarek?

Wysoka Izbo! Pani Minister! Projekt ustawy ma na celu zwiększenie liczby osób kształcących się w zawodach pielęgniarki i położnej oraz dostosowanie w średnim okresie liczby osób pracujących w tych zawodach do rosnących potrzeb związanych z tymi usługami. Mam pytanie do pani minister: W jaki sposób ustawodawca chce zachować wymogi dotyczące jakości kształcenia, a w szczególności zagwarantowania nie mniejszej liczby godzin kształcenia zawodowego na studiach niestacjonarnych niż liczba godzin w ramach formy stacjonarnej? Drugim celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie dodatkowego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych. Czy ustawodawca nie dostrzega ryzyka związanego z tym, że prawo do tego dodatkowego urlopu szkoleniowego może pogłębić istniejące problemy kadrowe w podmiotach leczniczych?

Czy to prawda, pani minister, że pracodawcy nie byli stroną porozumienia, na które powołuje się rząd, wprowadzając przedłożoną nowelizację? Dziękuję. Pan poseł Andrzej Gawron. Panie Marszałku! Pani Minister!

Pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Marszałku! Pani Minister! Przeglądając strony uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, można zauważyć, że zainteresowanie tym zawodem jest poniżej oczekiwań.

Pan poseł Michał Szczerba. Panie Marszałku! Pani Minister! Stawiam pytanie kluczowe, pani minister: Czy czeka nas ostatni dyżur?

Niedawno minister Szumowski uczestniczył w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, gdzie wypowiedział takie słowa: Bez nowych pielęgniarek i pielęgniarzy grozi nam likwidacja systemu ochrony zdrowia w Polsce. Podpisujemy się, pani minister, pod tymi słowami. W przyszłym roku 103 tys. pracujących pielęgniarek osiągnie wiek emerytalny. To stanowi 44% obecnie zatrudnionych. Niewiele lepiej wygląda sytuacja kadr lekarskich, co czwarty lekarz jest w wieku emerytalnym. Bardzo niska płaca za katorżniczą pracę - tak wygląda praca polskiej pielęgniarki.

To także bardzo niskie wydatki państwa na ochronę zdrowia. Przypomnijmy, 4,7% PKB wydajemy na ochronę zdrowia, w sytuacji kiedy Czechy wdają 7,8%. To jest sytuacja, która powinna nas [[Dzwonek]] skłaniać do refleksji. Dziękuję. Pani poseł Anna Kwiecień. Dziękuję. Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Sejmie! Ja chciałam rozpocząć od podziękowań.

Ten niedobór to nie jest kwestia ostatnich 3 lat, tylko to jest kwestia długoletniej polityki, wielu lat zaniedbań w tym zakresie. Pojawiła się ogromna dziura pokoleniowa, która zaczęła się tworzyć już w latach 90., kiedy był ogromny odpływ zarówno personelu pielęgniarskiego, jak i lekarskiego do innych zawodów.

Ale ja mam pytanie odnoszące się do tych 6 dni urlopu.

Pewne wątpliwości przy tej ustawie w związku z wprowadzeniem studiów niestacjonarnych budziło to, czy standard kształcenia na tych studiach będzie zabezpieczony. Chodzi zarówno o poziom kadry wykładającej, jak i odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych, teoretycznych itd. Ale, jak sądzę, ustawa zobowiązuje do respektowania standardów ministra nauki i szkolnictwa wyższego i możemy być spokojni, że te kwestie będą pod kontrolą, czyli pod kontrolą będzie jakość kształcenia na takich studiach.

Czy pani minister mogłaby coś bliżej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że to jest bardzo istotna sprawa? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Pani Minister! To, że brak jest pielęgniarek i położnych, to jest fakt i dziękuję za to, że ministerstwo myśli o tym i wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Ale moje pytanie jest takie: Czy w ministerstwo wspólnie z ministerstwem edukacji nie myśli nad tym, aby np. wprowadzić też edukację w tym zakresie, na pewno nie pełną, ale na poziomie szkoły średniej? Jest młodzież, która np., zdarza się, nie zdaje matury. Czy mamy szkoły policealne roczne, dwuletnie, które by przygotowywały do tego zawodu?

Biuro poselskie to jak półkonfesjonał, można powiedzieć. Dowiadujemy się rzeczy, o których niekoniecznie chcielibyśmy wiedzieć, bo nie jest dobrze wszystko wiedzieć. Chcę powiedzieć, pani minister, następującą rzecz.

Czy lekarzy - 2,4% na 10 tys. mieszkańców, czyli o połowę mniej w stosunku do innych państw - w jakiś sposób przybędzie? Najwięcej skarg, 80%, jest właśnie na lekarzy, niewłaściwe odnoszenie się itd., itd. Oni są zmęczeni, ci lekarze, też.

To jest konieczne, jeśli chodzi o lekarzy.

Choroby Parkinsona, neurodegeneracyjne to jest koszmar, pani minister.

Szanowni Państwo Posłowie! Gdy czyta się projekt dotyczący zmian ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, najbardziej zdumiewa fakt, że ustawodawca jest przekonany, że wprowadzone zmiany w jakimkolwiek stopniu zmienią obraz tego zawodu.

Do końca 2020 r. 44% pielęgniarek nabędzie prawo do przejścia na emeryturę, a my serwujemy kosmetyczną ustawę, która dodatkowo obniży standardy kształcenia i prestiż zawodu. Nie ma możliwości, by zajęcia praktyczne, które według ustawy mają być jednakowe dla obu trybów nauczania, nie zróżnicowały umiejętności zawodowych. W jaki sposób studenci odbywający praktyki zawodowe w szpitalu wyłącznie w weekendy mają posiąść te same umiejętności, które nabędą studenci odbywający praktykę permanentną? To moje pytanie do twórców ustawy. Wszyscy dobrze wiemy, że potrzebne są rozwiązania systemowe zachęcające absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie i pozostania w Polsce. Trzeba przywrócić temu zawodowi godność. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zatrzymać pielęgniarek w Polsce wynagrodzeniem, to stwórzmy program stypendialny, grantowy, [[Dzwonek]] preferencji mieszkaniowej i wykreujmy okoliczności, które zmotywują do pracy w polskich szpitalach i ośrodkach. Zaangażujmy dodatkowo samorządy terytorialne do wsparcia tego programu. Nie siedźmy tutaj nad ustawą odwracającą kota ogonem i udającą, że coś zmieni. Na to pytanie i wcześniejsze pytania odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Bardzo chciałabym podziękować za te pytania, szczególnie opozycji.

Ta ustawa, którą dzisiaj prezentujemy, to jedno z wielu rozwiązań, które obecny rząd od 3 lat systematycznie przygotowuje i wprowadza w życie. Szkoda, że państwo w trakcie 8 lat rządów nie zrobiliście nic. Dowody na to państwu podam. Pan poseł Szczerba zarzuca obecnemu rządowi, że przeznacza za mało środków na ochronę zdrowia.

To nasz rząd po raz pierwszy przyjął ustawę, która gwarantuje systematyczny, coroczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia - do 6% produktu krajowego brutto w 2024 r. A za waszych czasów, w 2015 r., przeznaczono 72 mld zł. Szanowni Państwo! Kolejnym zarzutem, który państwo czynicie, jest to, że pielęgniarki wyjeżdżają za granicę. W ostatnim roku, szanowni państwo, do samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu zgłosiło się więcej pielęgniarek, niż ukończyło studia. To znaczy, że 100% pielęgniarek uzyskuje prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego że podjęliśmy konkretne, systemowe działania, które realizujemy od 4 lat.

To są zaplanowane, systematycznie realizowane działania. Wskazaliśmy, że pierwszym elementem, który należy zrealizować, jest zwiększenie wynagrodzenia pielęgniarek, bo rzeczywiście kilka lat temu pensje były żałosne. Jest to wynagrodzenie o ok. 30% wyższe niż ok. 3 lata temu. To my zrealizowaliśmy dodatek 4 razy 400 i wprowadziliśmy od września podwyższenie wynagrodzenia o 1100 zł. Dzięki temu mamy więcej pielęgniarek w systemie.

W ramach tego produktu, który będzie oddzielnie finansowany, pielęgniarki będą mogły wykorzystać m.in. takie kompetencje, jak przepisywanie leków, ordynowanie leków, wystawianie skierowań na badania, badanie fizykalne, czyli te kompetencje, które nabywają w toku kształcenia zawodowego.

Podjęliśmy takie działania; m.in. z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych realizujemy promocję tego zawodu. To jest konkretny projekt, który w tej chwili startuje i jest realizowany. Ale zachęcamy również poprzez uatrakcyjnienie procesu kształcenia.

Polega on na tym, że przekazujemy środki w ramach umowy do szkoły, która kształci pielęgniarki, na stypendia w wysokości 800 zł dla każdej studentki od II roku studiów. W ubiegłym roku ten program rozszerzyliśmy nawet o etap po zakończeniu studiów, czyli absolwentka, która ukończy studia i podejmie pracę w polskim systemie ochrony zdrowia finansowanym ze środków publicznych, może jeszcze przez 2 lata otrzymywać dodatkowo 1 tys. zł, oprócz wynagrodzenia, które zaproponuje jej pracodawca. Rozumiem, że jest to pytanie zadane po to, żeby państwa o tym poinformować. Uczelnie, które kształcą, są tym zainteresowane i takie programy realizują. W 2015 r. były w kraju 74 uczelnie, które kształciły na kierunku pielęgniarstwo, a teraz mamy ich 98. Jest różnica? O 30% zwiększyła się liczba uczelni, na których kształcone są pielęgniarki.

W tym roku nabór to 6600. Ten nabór będzie skutkował konkretnymi efektami za 3, 4 lata. To są też twarde dane z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

To są fakty, to są dane, które wynikają z rejestrów. Rzeczywiście mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

To nie jest tak, że zwiększamy liczbę miejsc, a nie przekazujemy środków. Teraz kwestia urlopów. Zresztą kryteria określone w warunkach udzielania świadczeń świadczą o tym, że pielęgniarki muszą ustawicznie podnosić swoje wykształcenie. Zdecydowaliśmy się, że wprowadzimy jako przepis ogólnie obowiązujący 6-dniowy urlop szkoleniowy, który pielęgniarka może wykorzystać właśnie na kształcenie podyplomowe.

Chcę państwu przypomnieć, że na wielu stanowiskach pracy wymagane są odpowiednie kwalifikacje podyplomowe, specjalizacja, kurs kwalifikacyjny czy specjalistyczny, i oczywiście pracodawca może przyjąć pielęgniarkę, która posiada takie kwalifikacje, jednak jest to problem, ale może też własną pielęgniarkę wykształcić, umożliwiając jej to m.in. poprzez udzielenie jej urlopu szkoleniowego. Pytali państwo również o to, czy zamierzamy zmienić zakres czynności pielęgniarek, które wykonują w szpitalu, gdyż są zbyt obciążone pracą, która nie wymaga kwalifikacji pielęgniarskich, administracją. Tak, rzeczywiście, to my wprowadziliśmy od 1 stycznia obowiązek zatrudniania przez pracodawców sekretarek medycznych i opiekunów medycznych, bo opiekunów medycznych mamy na rynku, są w kraju szkoły, które kształcą opiekunów medycznych, natomiast oni nie byli zatrudniani w szpitalach i pielęgniarki wykonywały czynności, które niekoniecznie muszą wykonywać, np. transport chorego czy transport materiału do badań. W związku z tym podjęliśmy te regulacje. Dyrektorzy, którzy nie widzieli takiej potrzeby, teraz są zobligowani przepisem prawa, bo istnieje w tym zakresie stosowne rozporządzenie. Reasumując, nie jest to kosmetyczna zmiana. Ta zmiana jest elementem realizowania konkretnej strategii, strategii opracowanej w 2016 r., która została przyjęta przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. Obecnie ta strategia będzie przyjęta przez rząd w formie uchwały, czyli będzie to dokument, który będzie realizowany przez kolejne rządy, w którym wskazujemy, jakie działania, w jakim okresie muszą być realizowane, żebyśmy nie doszli do sytuacji, do której tutaj jeden z panów posłów nawołuje, czyli ostatniego dyżuru. Mamy nadzieję, że te działania do takiej sytuacji nie doprowadzą.

Jeden z posłów sygnalizował kwestię uruchamiania w Wieluniu nowej szkoły. Współpracowaliśmy w tym zakresie i udało się ją uruchomić.

Ta strategia jest realizowana i przynosi konkretne efekty w postaci wzrostu liczby pielęgniarek na rynku. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.

Pani Minister!

Pani Minister!

Trzeba bić na alarm.

odniesie się ktoś do treści wystąpienia. Chwali się to i cieszą uszy słowa, które pani wypowiedziała. Ale opinia publiczna musi wiedzieć jedną rzecz.

Druga sprawa. Żeby zwiększyć ilość wykształconych pielęgniarek, trzeba przygotować określoną ilość miejsc edukacyjnych itd. Tu potrzebny jest czas. Nie zrobi się tego w 1 czy 2 miesiące. Pani Minister! Kryzys gospodarczy to inne pojęcie niż boom gospodarczy. To są zupełnie inne światy.

Dziękuję bardzo. Zamykam. Chyba że pani minister chce jeszcze się odnieść do tego.

Po pierwsze, chciałabym odpowiedzieć na komentarz pana posła. zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Jest to pierwsza regulacja sektorowa, która gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia systematyczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Mamy określone minimalne poziomy, które obowiązywały w 2017 r., i rzeczywiście z dniem wprowadzenia tej ustawy był taki poziom podstawowego wynagrodzenia zasadniczego minimalnego.

To obecny rząd, pan premier Morawiecki podjęli decyzję, że kwotą bazową, od której liczymy wskaźniki, które są trochę skomplikowane, więc nie będę o nich mówić. Kwotą bazową w chwili, kiedy przygotowywaliśmy tę uchwałę, była kwota 3900 zł.

Tak jak pan poseł mówił.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań.

Pan poseł Maciej Małecki przedstawi sprawozdanie komisji. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Komisja pracowała nad tym dokumentem na dwóch posiedzeniach. Pierwsze czytanie odbyliśmy 12 czerwca. Wtedy pojawiły się poprawki zgłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i były one omawiane do czasu dzisiejszego posiedzenia, kiedy to rozpatrzyliśmy cały projekt ustawy. Zostało zgłoszonych 7 poprawek. Komisja przyjęła te poprawki i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tego bardzo ważnego dla nas dokumentu regulującego, wzmacniającego polskie interesy na naszym odcinku gazociągu jamalskiego. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wystąpi pan poseł Maciej Małecki. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne.

Konkretnie doprecyzowaniu będą podlegały obowiązki operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu połączonego gazowego, a także kompetencje prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego.

Natomiast operatorem polskiej części Jamału jest spółka Gaz-System - tu nastąpiło wyznaczenie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do roku 2025. Obecnie obowiązująca umowa o powierzeniu obowiązków operatora gazociągu jamalskiego, którą zawarły Gaz-System i EuRoPol GAZ, regulująca jednocześnie zasady wzajemnych relacji pomiędzy spółkami, wygasa z końcem tego roku, czyli 31 grudnia. Należy także zaznaczyć, że treść obecnie obowiązującej umowy nie pozwala spółce Gaz-System na wykonywanie wszystkich funkcji operatorskich gazociągu jamalskiego, m.in. w zakresie obsługi tłoczni gazu czy obsługi systemu informatycznego, a tym samym jest niezgodna z polskim interesem i z prawem europejskim. Dlatego istnieje poważne ryzyko, że podpisanie nowej umowy powierzeniowej, ale takiej, która będzie zabezpieczała polskie interesy i będzie zgodna z prawem europejskim, zostanie zablokowane przez rosyjskiego akcjonariusza EuRoPol Gazu, czyli spółkę Gazprom, i tym samym od 1 stycznia 2020 r. nie byłoby żadnej umowy powierzeniowej, a Polska miałaby jeszcze mniejszy wpływ na kontrolę nad gazociągiem jamalskim na naszym terytorium.

Obliguje strony do zawarcia stosownej umowy i jednocześnie - to bardzo ważne - wyposaża prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w kompetencję do ustalenia warunków nowej umowy powierzeniowej w drodze decyzji w sytuacji, w której nie doszłoby do zawarcia umowy między Gaz-Systemem a EuRoPol Gazem na 30 dni przed wygaśnięciem obecnie obowiązującej umowy. Ponadto projekt zawiera przepisy umożliwiające egzekucję wykonania decyzji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Projekt, mimo że dotyka bardzo wąskiej materii, skutki będzie miał bardzo poważne, bowiem bardzo mocno podniesie bezpieczeństwo energetyczne Polski. I to jest priorytet Prawa i Sprawiedliwości, wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Im mniej rosyjskiego wpływu na system gazowy Polski, tym lepiej. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera ten projekt i zachęcam do tego całą Wysoką Izbę. Zapraszam pana posła Pawła Bańkowskiego z klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska do przedstawienia wystąpienia w imieniu tego klubu. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, druki nr 3497 i 3501.

Proponowane w projekcie ustawy zmiany mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne dotyczących obowiązków operatora systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego oraz operatora systemu połączonego gazowego, a także kompetencji krajowego organu regulacyjnego, czyli prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie kształtowania relacji pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesyłowego gazowego albo operatorem systemu połączonego gazowego.

Proponowana zmiana tego przepisu polega na dodaniu ust. 6b, który ma stanowić, że w przypadku powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora dystrybucyjnego gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego, operator ten w obszarze swojego działania jest odpowiedzialny za wydawanie warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do sieci. Art. 9h ustawy określa zasady powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego. Zmiana tego przepisu polega na wprowadzeniu do niego postanowień, które dotyczą sytuacji, gdy prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczy przedsiębiorstwo energetyczne na operatora systemu przesyłowego gazowego na określonej sieci przesyłowej na okres dłuższy niż okres obowiązywania umowy powierzającej pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego z wykorzystaniem tej sieci. W takiej sytuacji zgodnie z propozycją wnioskodawców właściciel sieci przesyłowej miałby obowiązek zawrzeć z operatorem koleją umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego. W art. 23 ust. 2 ustawy - określa on zakres działania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - wnioskodawcy proponują wprowadzenie do niego zmian, które są konsekwencją zmian w art. 9h ustawy. Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Prawo energetyczne decyzja prezesa URE o wyznaczeniu operatora sieci przesyłowej gazowej nie reguluje w sposób zupełny praw i obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego oraz właściciela sieci związanych z pełnieniem przez to przedsiębiorstwo funkcji operatora sieci przesyłowej. W związku z tym konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy właścicielem sieci a przedsiębiorstwem energetycznym. W projekcie ustawy wprowadzono również możliwość wydania przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postanowienia, którym do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego określone zostaną warunki powierzenia pełnienia obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego, co pozwala na zapewnienie ciągłości w wykonywaniu funkcji operatora. W przepisach przejściowych przesądzone zostało, że do umów powierzających wykonanie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego zawartych pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej wchodzącej w skład systemu przesyłowego, który w dniu 3 września 2009 r. należał do przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, a przedsiębiorstwem energetycznym posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania paliw gazowych, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu wygaśnięcia tych umów stosuje się przepisy Prawo energetyczne w brzmieniu dotychczasowym. Z uwagi na charakter przedmiotowej regulacji oraz konieczność pilnego uzupełniania przepisów Prawa energetycznego wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przemawia za tym potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego gazowego oraz możliwości korzystania z tego systemu. Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie przewiduje wydania aktów wykonawczych, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, nie wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz średnich przedsiębiorstw, nie został również poddany konsultacjom. W czasie rozpatrywania projektu ustawy zgłoszono siedem poprawek, które wynikają z uwag zgłoszonych przez Urząd Regulacji Energetyki oraz mają charakter redakcyjno-legislacyjny. Podsumowując moje wystąpienie, pragnę poinformować Wysoką Izbę, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim to uczyni, pozwolicie państwo, że pozdrowię gości, członków klubu seniora z Rymanowej, którzy przyjechali do Warszawy do Sejmu na zaproszenie pani poseł Joanny Frydrych.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Będziemy wspierać pracę nad tą ustawą.

Liczę, że dzięki temu będziemy jako państwo bezpieczni. Przechodzimy do pytań w tym punkcie posiedzenia. Czy ktoś z pań posłanek i panów posłów chce wpisać się na listę? Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Przy okazji procedowania nad tym przedłożeniem chciałbym zapytać pana ministra: Czy prowadzone są prace zmierzające w kierunku wsparcia budowy infrastruktury gazowej na obszarach, gdzie przyłączenie na warunkach komercyjnych jest nieopłacalne dla operatorów systemu dystrybucji w związku z kosztami inwestycji? Takie mechanizmy, jak się wydaje, mogłyby być skuteczne w ramach walki ze smogiem. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Mianowicie po pierwsze oczywiście wiemy, że bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z tych najważniejszych wyzwań, które stoją przed naszym krajem, natomiast przeczytałem ten projekt ustawy i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie: Dlaczego te umowy właścicieli sieci przesyłowej gazowej, które zawiera się z operatorem systemu przesyłowego gazowego, są zawierane na okres, jak to wynika z ustawy, nie dłuższy niż 3 lata, tzn. dlaczego jest taki okres zaproponowany, a nie przykładowo 4 czy 5 lat?

Dlaczego nowelizacja Prawa energetycznego, nawet tak specjalistyczna, jak ta, która tutaj jest, nie została poddana konsultacjom? Bardzo proszę. Pani Marszałek! Moje pytanie nie dotyczy dokładnie tej nowelizacji, ale zadam je w imieniu mieszkańców Chorzowa, zwłaszcza dzielnicy Chorzów Stary, ponieważ jest to bardzo duży problem dla mieszkańców tej dzielnicy. Mianowicie elektrownie, elektrociepłownie mają obowiązek spalania biomasy. Odór pochodzący z pryzm, w których magazynowana jest ta biomasa, jest nie do wytrzymania nawet w promieniu 1,5 km od danej elektrowni, a mówię tutaj konkretnie o elektrowni CEZ w Chorzowie. I dlatego mam takie pytanie, a jeżeli pan minister nie może zaraz odpowiedzieć, to prosiłabym o odpowiedź na piśmie: Jakie są normy dotyczące tej biomasy, jakie są normy gromadzenia biomasy? Myślę, że to, jeżeli. Ja wiem, że to pytanie nie dotyczy. Nie ten minister. To w takim razie będę z tym pytaniem zwracała się w imieniu mieszkańców do innego ministerstwa, bo jest to problem, który utrudnia życie wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy. Pani poseł Zofia Czernow, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Wysoki Sejmie! Projekt ustawy zmieniający ustawę Prawo energetyczne jest bardzo ważnym projektem, bo reguluje niezwykle ważny problem bezpieczeństwa energetycznego Polski. I ja absolutnie jestem za tym, żeby nad tym projektem procedować i czuwać nad bezpieczeństwem energetycznym, i wyprzedzać wszystkie działania, które są potrzebne, ale proszę państwa, tak ważny projekt, żeby był projektem poselskim, to się nigdy nie zdarzyło, nie zdarzało. Po pierwsze, jest projektem poselskim, po drugie, nie był poddany żadnym konsultacjom, co jest w ogóle przy tak ważnych sprawach, uważam, nie do przyjęcia, i po trzecie, jest bez żadnego vacatio legis. Przecież słyszałam w wypowiedziach państwa posłów, że problem [[Dzwonek]] będzie aktualny na koniec roku, a tymczasem ustawa wchodzi w życie w dniu następnym po podjęciu. Uważam, że to jest niepoważne traktowanie tak ważnej sprawy. Na to i wcześniejsze pytania odpowie pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej pan Piotr Naimski. Bardzo proszę.

Może tak. Ta ustawa jest ważną ustawą, dlatego że porządkuje relacje pomiędzy operatorem systemu przesyłowego a właścicielem czy właścicielami infrastruktury i umowa, która te relacje reguluje, czy umowy, które te relacje regulują, po pierwsze, muszą być pod kontrolą Urzędu Regulacji Energetyki, a po drugie, Urząd Regulacji Energetyki musi mieć narzędzie, musi mieć możliwość zastąpienia swoimi decyzjami braku umowy, jeżeli taki mógłby wystąpić. Z tego punktu widzenia ta ustawa, ten poselski projekt ustawy rzeczywiście trafia w zapotrzebowanie, w potrzeby, w to, co w tej chwili powinno być w naszym systemie regulacyjnym wprowadzone. Materia tej ustawy jest na tyle specyficzna, że poddawanie konsultacjom społecznym tego projektu wydaje się niezasadne. Ta ustawa nie ma bezpośredniego wpływu na stosunki społeczne, na lokalne społeczności, na te podmioty, które zwykle biorą udział w konsultacjach innych regulacji prawnych czy innych ustaw. To jest czysto techniczne posunięcie ustawowe, które umożliwi Urzędowi Regulacji Energetyki dotrzymanie tego reżimu prawnego, który będzie musiał obowiązywać od roku 2020 i dalej. Wydaje się, że jest to wystarczająca argumentacja do tego, żeby ta ustawa właśnie w takim trybie była uchwalana, za co Wysokiej Izbie i komisji dziękuję.

Chodzi o to, żeby zakresem funkcjonowania, długością funkcjonowania umowy nie ograniczać w przyszłości tych możliwości, tych być może pożądanych zmian. Jeśli chodzi o pytanie pani poseł Nowak, rzeczywiście biomasa to nie jest zakres moich kompetencji i obowiązków.

Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Z końcem tego roku upływa umowa pomiędzy operatorem, Gaz-Systemem, a właścicielem tego gazociągu, EuRoPol Gazem. W EuRoPol Gazie jest sytuacja taka, że ze względu na decyzję naszych poprzedników, rządu Platformy i PSL-u, kluczowe decyzje spółki wymagają jednomyślności, czyli jednocześnie zgody części zarządu delegowanych przez Polskę i przez Rosję, czyli i PGNiG, i Gazprom, i oczywiste jest, że strona rosyjska nie będzie zabiegała o polskie interesy.

Apeluję do całej Wysokiej Izby, żeby co jak co, ale sprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski i kolejnego kroku w uwalnianiu się od rosyjskiej dominacji gazowej... żeby w tej Izbie takie ustawy były przyjmowane jednogłośnie. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (druki nr 3483 i 3559) Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Komisja Kultury i Środków Przekazu 2 lipca br. rozpatrzyła prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Przypomnę, że istotą projektu jest przedłużenie na rok 2022 działania Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i konsekwentnie przedłużenie o rok okresu przyznawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Tym samym na rok 2023 przesuwa się czas przyjęcia sprawozdania z działania komitetu. Komisja Kultury i Środków Przekazu, przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących się, przyjęła projekt bez poprawek i taką też rekomendację przedstawia Wysokiej Izbie. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wysoka Izbo! Prezydent Andrzej Duda powiedział kiedyś: „Jestem głęboko przekonany, że stulecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich współtworzenia” Spełniły się w tysiącach większych i mniejszych inicjatyw międzynarodowych, ogólnokrajowych, ale też bardzo, bardzo lokalnych. W dużej części są to działania wspomagane czy choćby firmowane przez rządowy program „Niepodległa” Istotną częścią tych obchodów jest funkcjonowanie komitetu narodowych obchodów 100. rocznicy, ciała pluralistycznego, łączącego najprzeróżniejsze środowiska polityczne, ideowe, społeczne, także zawodowe. Jedną z najważniejszych inicjatyw jubileuszowych jest uhonorowanie Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości osób, które dobrze zasłużyły się w sprawie odzyskania, utrwalania polskiej niepodległości, suwerenności, a także sprawie sławienia Polski w świecie. Takich medali przyznano już prawie 800. Warto kontynuować tę dobrą pracę, a przecież jest po temu okazja czy podstawa.

Dopiero wtedy rozpoczęło się instalowanie na Górnym Śląsku polskiej administracji. Przywołajmy więc jeszcze raz słowa prezydenta Dudy: Chciałbym, abyśmy upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofali się o 100 lat, co w równym, a może nawet większym stopniu wybiegali myślą naprzód - ku wyzwaniom, które na nas czekają, przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując silną, wolną Polskę. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość oczywiście popiera przedłożoną ustawę. Zapraszam pana posła Marka Wójcika, który przedstawi stanowisko klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska wobec tego projektu ustawy. Otóż jestem zadowolony z projektu tej ustawy, dlatego że uwzględnia ona pewną historyczną prawdę, tzn. fakt, że Śląsk został przyłączony do II Rzeczypospolitej w 1922 r.

Problem w tym, że procedowana dzisiaj ustawa byłaby niepotrzebna, gdyby rok temu, w czerwcu 2018 r., uwzględniono moje poprawki i argumenty w dyskusji nad ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wówczas zupełnie niepotrzebnie posłowie PiS-u, posłowie większości parlamentarnej odrzucili poprawki. Efektem tej sejmowej debaty z ubiegłego roku i tej dyskusji nad historią Górnego Śląska jest pewna próba naprawienia błędu, który rzeczywiście w organizacji tych rządowych obchodów się pojawił, błędu, z którego wprost wynika nieuwzględnienie specyfiki śląskiej historii właśnie w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I pierwszym sygnałem, że państwo z tego błędu chcecie się wycofać, była zmiana uchwały Rady Ministrów tworzącej program „Niepodległa”

Ustawa, nad którą dzisiaj debatujemy, jest takim kolejnym krokiem, żeby rzeczywiście oddać tę historyczną sprawiedliwość.

Warto przypominać o tym, że tak nie było, dlatego że prawda historyczna jest po prostu inna.

Co więcej, wtedy rozpoczęło się budowanie na Śląsku polskiej administracji. Wojsko Polskie było przez kolejne dni w wielu miastach w sposób bardzo uroczysty i bardzo barwny witane przez lokalną ludność. Może pan minister nie wie, że często powitanie wojsk polskich wyglądało w ten sposób, że ustawiano takie specjalne bramy powitalne w Szopienicach, w Katowicach, w Chorzowie, w wielu miejscowościach. To jest coś, o czym my pamiętamy. Często staramy się te instalacje odtwarzać z okazji różnego rodzaju okrągłych rocznic dotyczących tych wydarzeń.

Panowie Ministrowie! Tak jak wspomniałem, klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska będzie popierał tę nowelizację. Myślę, że lepiej późno niż wcale.

Zapraszam pana posła Tomasza Jaskółę do przedstawienia stanowiska w imieniu klubu Kukiz’15.

Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Odzyskanie niepodległości Polski miało ścisły związek z walką o granice oraz kształtowaniem się granic. Poszczególne części Polski w różnym okresie były do niej przyłączane.

Ale jeszcze jeden region został przyłączony w 1922 r., mianowicie Wileńszczyzna.

Ze względu na to, iż te dwa regiony zostały przyłączone w 1922 r., zasadne jest wydłużenie realizacji zadań komitetu do Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Ślązakom, zwłaszcza dumnym potomkom powstańców, to się po prostu należy, zwłaszcza w czasach, w których wrogowie Polski usiłują dążyć do podważenia polskiej tożsamości Śląska. Pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, zada ostatnie pytanie w tym punkcie. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytanie do pana ministra Sellina. W marcu tego roku w Katowicach pan premier Morawiecki poinformował o tym, że na obchody stulecia wybuchu powstań śląskich będą przeznaczone rządowe pieniądze. Myśmy tę zapowiedź przyjęli z dużym zadowoleniem, natomiast po interpelacjach, które kierowałem do resortu, który pan reprezentuje, jak również po interpelacjach do premiera okazało się, że pieniądze na obchody 100. rocznicy wybuchu powstań śląskich to są pieniądze, które są zapisane w programie „Niepodległa” Panie Ministrze! Chciałbym zaapelować o to, żeby na te obchody zarezerwować trochę większą kwotę, dlatego że to jest stulecie naprawdę ważnych wydarzeń, biorąc pod uwagę historię Śląska i historię całej Polski.

Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem bardzo serdecznie podziękować za poparcie projektu pana prezydenta Andrzeja Dudy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Chcę wyjaśnić panu posłowi Markowi Wójcikowi pewną kwestię.

Pamiętam dyskusje w Senacie, bardzo długie, przy tej pierwszej ustawie.

Ale tam nie było tak wytrawnych znawców historii Śląska, jak w Sejmie.

Niemniej jednak chciałem bardzo serdecznie podziękować za poparcie tego projektu. Myślę, że wspólnie, razem, wszyscy, tak jak do tej pory, będziemy jako naród pięknie obchodzili, bo cały czas te obchody trwają, 100. rocznicę odzyskania niepodległości, a że to się rozkłada w czasie, to już jest niestety nasza historia. Dziękuję bardzo.

Dziękuję bardzo. To jest rzeczywiście kompatybilne z decyzją, którą podjął rząd, po pierwsze, o uruchomieniu wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”, o powołaniu pełnomocnika rządu do spraw obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości - tę funkcję mam zaszczyt piastować - i o realizacji tego programu już od roku 2017 r.

To zresztą było omawiane też na posiedzeniu komitetu honorowego narodowych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i komitetu prezydenckiego, który się kilkakrotnie zebrał. Ja mam przyjemność pełnić funkcję sekretarza tego komitetu i nad tym tematem tam też żywo dyskutowano.

Odpowiadając konkretnie na pytania, które tutaj padły.

Nazywa się Kordegarda.

Pan mnie trochę tym pytaniem zaskoczył, więc pan pozwoli, że ja odpowiem panu na piśmie.

To jest program, w przypadku którego mogą aplikować różnego rodzaju organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury czy wojewodowie.

Tych wydarzeń na pewno jest dużo.

Tak więc tych wydarzeń oczywiście jest dużo, ale te śląskie rocznice są też honorowane i jeśli są aplikacje, jeśli są inicjatywy oddolne, to są one chętnie wspierane przez biuro programu „Niepodległa” Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3489 i 3506) Pan poseł Włodzimierz Bernacki przedstawi sprawozdanie komisji. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 3489. Marszałek Sejmu, na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, skierował w dniu 4 czerwca 2019 r. powyższy projekt uchwały do Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych do pierwszego czytania. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. wnosi, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć projekt uchwały z druku nr 3489 bez poprawek. Wysoka Izbo! Pragnę zaznaczyć, że nowelizacja regulaminu polega na rozszerzeniu art. 175 przez dodanie ust. 8 w brzmieniu: Do czasu wniesienia przez posła odwołania marszałek Sejmu może uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu. Wysoka Izbo! Instytucja wykluczenia posła z posiedzenia Sejmu jest uregulowana w art. 175 ust. 5, 6 i 7 regulaminu Sejmu. Zgodnie z art. 175 ust. 5 regulaminu Sejmu, przypadku gdy poseł po dwukrotnym przywołaniu do porządku nadal uniemożliwia prowadzenie obrad, marszałek Sejmu ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu. Poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu jest obowiązany natychmiast opuścić salę posiedzeń, a jeżeli tego nie zrobi, marszałek Sejmu zarządza przerwę w obradach. Wykluczenie z posiedzenia Sejmu jest jedną z kompetencji porządkowych przysługujących prowadzącemu obrady marszałkowi lub wicemarszałkowi Sejmu w odniesieniu do posłów. Zgodnie z art. 175 ust. 6 regulaminu Sejmu poseł wykluczony z posiedzenia Sejmu może odwołać się od decyzji o jego wykluczeniu do Prezydium Sejmu, które niezwłocznie rozstrzyga sprawę po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy poseł nie bierze udziału w posiedzeniu. O sposobie załatwienia odwołania Prezydium Sejmu niezwłocznie zawiadamia Sejm, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu. Decyzja Prezydium Sejmu jest ostateczna. Obecnie przepisy regulaminu Sejmu nie przewidują możliwości wycofania się przez marszałka lub wicemarszałka z podjętej decyzji o wykluczeniu posła. Wydaje się jednak, że wykluczający posła z posiedzenia Sejmu powinien dysponować możliwością wycofania się ze swojej decyzji. Przemawiają za tym względy celowościowe. W niektórych przypadkach podtrzymywanie decyzji o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu może okazać się mniej efektywne aniżeli odstąpienie od tej decyzji na rzecz zaprowadzenia porządku w trakcie obrad Sejmu. Niekiedy bowiem z punktu widzenia celu tej instytucji bardziej skuteczne mogą się okazać działania koncyliacyjne, których efektem będzie z jednej strony wycofanie się marszałka lub wicemarszałka Sejmu z decyzji o wykluczeniu posła, a z drugiej - zaprzestanie przez posła zachowania uniemożliwiającego prowadzenie obrad. W projekcie przewidziano, że marszałek Sejmu będzie mógł uchylić swoją decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia Sejmu do czasu wniesienia przez posła odwołania. Anulować decyzję o wykluczeniu posła z posiedzenia będzie mógł jedynie marszałek albo wicemarszałek Sejmu, który tę decyzję pierwotnie podjął. Tylko w takim przypadku nie narusza to przepisów przewidujących tryb odwoławczy od decyzji o wykluczeniu posła, czyli art. 175 ust. 6 regulaminu Sejmu. Po drugie, wydaje się, że zbyt daleko idącą ingerencją w przepisy regulaminu Sejmu dotyczące trybu odwoławczego byłoby dopuszczenie cofnięcia decyzji o wykluczeniu z posiedzenia po złożeniu przez wykluczonego posła odwołania do Prezydium Sejmu. W takiej sytuacji, tj. formalnego wszczęcia procedury odwoławczej, jak się wydaje, wyłączna możliwość wzruszenia decyzji o wykluczeniu posła będzie należała do Prezydium. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość głos zabierze pan poseł Włodzimierz Bernacki. Dziękuję. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Otóż Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w pełni popiera zmiany zaproponowane we wniosku. Zapraszam pana posła Tomasza Głogowskiego do przedstawienia stanowiska w imieniu klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Chciałem przedstawić stanowisko klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska wobec projektu zmiany regulaminu Sejmu.

Jest to zmiana godna poparcia i klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska będzie głosować za tą zmianą.

Zresztą historia tej kadencji pokazuje, że niewycofanie się z pochopnej decyzji o wykluczeniu parlamentarzysty z obrad może powodować długotrwały kryzys parlamentarny.

I to też nie jest rzecz, przeciwko której bym protestował.

Wysoka Izbo! Państwo w tej kadencji regulamin Sejmu poprawiają, zmieniają, dyskutują o nim. Po co to wszystko, skoro i tak go nie przestrzegacie? Przecież wykluczacie tylko posłów opozycji. Nie zauważyłam, żeby kiedykolwiek był ukarany poseł koalicji rządzącej. Nie przestrzegacie regulaminu, prezydent Duda skierował ustawę Kodeks karny do Trybunału Konstytucyjnego, bo ma duże wątpliwości, czy tryb uchwalenia tejże ustawy był zgodny z regulaminem.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Otóż w trakcie prac nad tą zmianą poprosiliśmy Biuro Analiz Sejmowych o przygotowanie opinii dotyczącej innych przypadków wykluczenia posłów z posiedzenia Sejmu.

Widać bardzo wyraźnie, że z wykluczeniami, jeśli chodzi o wykluczenia z obrad, mieliśmy do czynienia nie tylko w trakcie tej kadencji.

Proszę?

Słusznie zauważył tutaj pan poseł Głogowski, reprezentujący Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, że w niektórych wypadkach lepiej jest zająć stanowisko koncyliacyjne, a więc prowadzić do koncyliacji i wycofać się z decyzji, co przed zmianą regulaminu tak naprawdę byłoby, jest do pewnego stopnia naruszeniem regulaminu. Lepiej wprowadzić tę zmianę, ponieważ to daje szansę osobie prowadzącej posiedzenie Sejmu, czyli marszałkowi, wicemarszałkowi, aby zająć takie stanowisko, które będzie sprzyjało dobrej atmosferze na sali posiedzeń.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 31. porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku (druk nr 3366) wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk 3515) Proszę prezesa Najwyższej Izby Kontroli pana Krzysztofa Kwiatkowskiego o przedstawienie sprawozdania.

Pani Marszałek! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Tegoroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli przypada w szczególnym czasie. W lutym tego roku obchodziliśmy 100-lecie Najwyższej Izby Kontroli. Pozwolę więc sobie zacząć od fundamentalnej refleksji na temat NIK-u. Twórcy najwyższego organu kontroli zarówno w II, jak i w III Rzeczypospolitej byli przekonani, że wiarygodną kontrolę budżetową oraz kontrolę wykonania zadań może przeprowadzić wyłącznie organ kontroli niezależny od rządu, którego członkom kolegium i kontrolerom stworzone zostaną daleko posunięte gwarancje, tak aby nie obawiali się formułowania krytycznych ocen, nie obawiali się ewentualnych reperkusji z tym związanych. Dlatego w opisujących działania Najwyższej Izby Kontroli ustawach zarówno tej pierwszej, z 1921 r., przygotowanej pod kierunkiem Józefa Higersbergera, jak i tej ostatniej, z 1994 r., przygotowanej pod kierunkiem prof. Lecha Kaczyńskiego zagwarantowano niezależność Najwyższej Izbie Kontroli, jej kolegiantom, wszystkim kontrolerom niezależnie od zajmowanych stanowisk. To sprawozdanie jest także z mojego punktu widzenia wyjątkowe jeszcze z jednego względu, bo jest ostatnie, które prezentuję. Z końcem sierpnia tego roku kończę kadencję jako prezes Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo! Ale nie tylko ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli reguluje pracę tego organu. Także konstytucja, najważniejszy akt prawny i fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej, w art. 202 stanowi, że Najwyższa Izba Kontroli podlega jedynie Sejmowi. Jak jednak zgodnie twierdzą wszyscy komentatorzy, podległość ta nie dotyczy w żaden sposób dokonywania ustaleń kontrolnych czy formułowania ocen. W tym obszarze izba jest w pełni samodzielna i niezależna, co potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 1998 r. Mówi o tym wyraźnie deklaracja z Limy przyjęta przez Kongres Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, ale podkreśla to w swoich dokumentach także Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wysoka Izbo! Z tej właśnie niezależności Najwyższej Izby Kontroli, a zwłaszcza jej kontrolerów, niezależnie od zajmowanego stanowiska, od inspektora, po radcę czy dyrektora, w dużej wierze wynika wiarygodność naszych raportów pokontrolnych oraz ich znaczenie dla obywateli. Dostrzegają oni, że działamy niezależnie, że nasze raporty są rzetelne i obiektywne. Dzisiaj z najnowszego badania wynika, że blisko 50% dorosłych Polaków - co ważne, niezależnie od sympatii politycznych - w ten sposób ocenia pracę NIK-u, jako dobrą lub bardzo dobrą.

Dzisiaj NIK jest oceniany jako jedna z najlepiej pracujących instytucji w naszym kraju. Doceniają to także osoby pochodzące z różnych środowisk politycznych. Były premier Jerzy Buzek wielokrotnie podkreślał niezwykłą rzetelność i profesjonalizm kontrolerów NIK-u czy zaangażowanie w pracę kierownictwa izby. Obecny prezydent Andrzej Duda, goszcząc kilka dni temu prezesów organów kontroli państw całej Unii Europejskiej, czyli tzw. Komitet Kontaktowy, któremu przewodniczyłem, podkreślił, pozwolę sobie zacytować, że Najwyższa Izba Kontroli w Polsce cieszy się niezwykłym uznaniem, ogromną estymą i wielkim szacunkiem, a NIK i jej kontrolerzy przestrzegają najwyższych standardów. Raporty NIK-u są również bardzo wysoko cenione przez przedstawicieli mediów, przez zewnętrznych i branżowych ekspertów tak w kraju, jak i za granicą. Podkreślają oni wysoką jakość prezentowanych przez izbę ustaleń, ocen i wniosków oraz ich istotne znaczenie dla procesu naprawy państwa. Bardzo ważne dla oceny współczesnej kondycji izby jest także zaufanie, jakim izba cieszy się na arenie międzynarodowej. NIK obecnie jest w zarządzie EUROSAI-u, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego, i w zarządzie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, INTOSAI. To nie tylko wyraz zaufania do naszej organizacji, ale także docenienie naszej aktywności. Niemal każdego roku NIK jest wybierana przez różne gremia międzynarodowe do pomocy kolejnym krajom, które mają europejskie aspiracje, czy do audytowania najbardziej prestiżowych instytucji i organizacji międzynarodowych, takich jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Rada Europy czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. Wskazując przy okazji sprawozdania za 2018 r. na obiektywne i zewnętrzne źródła oceny NIK-u, nie sposób pominąć jeszcze jednego bardzo dla nas ważnego źródła: opinii wyrażanych na temat NIK przez poszczególne komisje sejmowe, z którymi na co dzień współpracują kontrolerzy ze wszystkich departamentów i delegatur. Posłowie z tych komisji znają najlepiej zawarte w naszych raportach ustalenia, cenią dołączone analizy systemowe czy podzielają formułowane wnioski. Wszystkie komisje sejmowe, przedstawiając swoje opinie na rzecz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, oceniły pracę Najwyższej Izby Kontroli pozytywnie lub bez uwag. Za ten obiektywizm komisji sejmowych bardzo serdecznie dziękuję. Dobre oceny zewnętrzne NIK-u płynące z wielu źródeł, także ze strony audytora badającego na zlecenie Sejmu finanse NIK, świadczą o tym, że Izba funkcjonuje prawidłowo, że jej kadra kontrolerska i kadra kierownicza są dobrze przygotowane do wykonywania zadań, a przyjęte metody i standardy przeprowadzania kontroli są odpowiednio dobrane do stojących przed Izbą wyzwań. Budując nasz system zapewnienia jakości pracy, korzystaliśmy z międzynarodowych standardów kontroli państwowej, zwłaszcza standardów kontroli jakości INTOSAI, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej wszystkie organy kontroli na świecie. Wysoki Sejmie! Wszystkie szczegółowe dane dostarczyliśmy państwu w obszernym dokumencie, czyli sprawozdaniu z działalności Izby. Zwrócę więc uwagę na to, że ze względu na ograniczone ramy czasowe wystąpienia sejmowego przytoczę tylko te najważniejsze liczby obrazujące pracę Izby oraz wspomnę o absolutnie kilku kluczowych problemach oraz niektórych wybranych kontrolach. Resztę znajdziecie państwo w blisko 500-stronicowym sprawozdaniu z naszej działalności. W 2018 r. Izba przeprowadziła 2325 kontroli, czyli o 129 więcej niż w roku poprzednim. Kontrolami tymi objęliśmy - bo w niektórych podmiotach byliśmy wielokrotnie - ponad 1800 podmiotów. Obszary istotne z punktu widzenia obywateli i funkcjonowania państwa zostały zbadane w ramach 111 kontroli planowych. W tej liczbie mieści się również kontrola wykonania budżetu państwa, która traktowana jest jako jedna, ale w istocie składa się z 285 kontroli przeprowadzonych w 267 jednostkach. Tworząc plan pracy na zeszły rok, korzystaliśmy także z sugestii komisji sejmowych. Przyjęliśmy łącznie w tym zakresie - szerszym czy węższym - prawie 90% różnych wniosków, które od państwa wpływały. Oprócz kontroli planowych NIK zrealizowała także 91 kontroli doraźnych, najczęściej w reakcji na napływające do Izby sygnały o poważnych nieprawidłowościach. Istotnym źródłem inspirującym nas do podjęcia kontroli doraźnych były skargi kierowane do Izby. W 2018 r. napłynęło do Izby ponad 4 tys. skarg i wniosków, wśród których blisko 2,5% stanowiły skargi i wnioski przekazane przez parlamentarzystów i organy parlamentu. Wszystkie skargi uporządkowane wedle grup tematycznych zainicjowały wiele naszych kontroli lub zostały przekazane do innych właściwych organów publicznych. Na zlecenie NIK-u inne organy kontrolne państwa przeprowadziły prawie 150 kontroli doraźnych oraz udostępniły nam wyniki kolejnych 14 kontroli. Izba współdziałała także w siedmiu kontrolach z najwyższymi organami kontroli z innych państw, przygotowując tzw. międzynarodowe raporty. W roku 2018 przedłożyliśmy Sejmowi 191 informacji o wynikach kontroli planowych, w tym dotyczących wykonania budżetu oraz niektórych kontroli doraźnych. Przedstawiciele Izby uczestniczyli łącznie w ponad 300 posiedzeniach komisji sejmowych. W ubiegłym roku Izba sformułowała także 140 wniosków de lege ferenda, w tym 108 określiliśmy w kontekście potrzeby zmian ustawowych. Poziom realizacji tych wniosków oczywiście w pierwszym okresie zwyczajowo wynosi ok. 10%, ale w związku z tym, że proces legislacyjny trwa dłużej, później oczywiście te wyniki są znacząco wyższe. Jeśli spojrzymy na poziom realizacji tych wniosków, to mogę powiedzieć, że za ostatnie lata ok. 1/3 jest już zrealizowanych, nie licząc tych, które są w toku realizacji. Trzeba także wspomnieć, że w roku 2018 oprócz 140 wniosków de lege ferenda zawartych w informacjach i sformułowanych w wystąpieniach zawarliśmy w nich 4851 wniosków pokontrolnych, o ponad 300 wniosków więcej niż w roku 2017. Ponad 80% z tych wniosków zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Można więc stwierdzić bez żadnej przesady, że kontrolowane instytucje korzystają z większości formułowanych przez nas wniosków. W ten właśnie sposób NIK m.in. przyczynia się każdego roku do poprawy funkcjonowania państwa. Szanowni Państwo! Co roku pytacie także państwo o korzyści finansowe uzyskane przez Skarb Państwa w wyniku naszych kontroli. Jest to wymierny efekt naszych kontroli. Podobnie jednak jak w sprawie wniosków de lege ferenda czasami proces pozyskiwania korzyści dla Skarbu Państwa bywa czasochłonny. W sierpniu 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję, która nakazywała Polsce odzyskanie od spółki Autostrada Wielkopolska prawie 900 mln zł wraz z odsetkami. Wszystko to zaczęło się od naszej kontroli z 2010 r., kiedy to stwierdziliśmy, że rząd wypłacił prywatnym operatorom zbyt wysokie rekompensaty za zwolnienie ciężarówek z opłat za jazdę po autostradach.

Widzicie państwo, że często bywa tak, że efekty finansowe naszej pracy są rozłożone w czasie. Podobnie jest z zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach czy wykroczeniach. W zeszłym roku złożyliśmy ich ok. 100 i było to o 17 więcej niż rok wcześniej. Złożyliśmy także 58 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w których ujawniliśmy 259 czynów dotyczących naruszenia dyscypliny finansowej. Wysoka Izbo! Tak jak powiedziałem, nie opowiem państwu o wszystkich kontrolach. Powiem tylko o kilku. Myślę, że jedną z najważniejszych zeszłorocznych kontroli była kontrola dotycząca działań na rzecz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. Stwierdziliśmy, że na terenie Unii Europejskiej Polska jest jednym z krajów z najgorszą jakością powietrza. Oceniliśmy także, że działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych, z wyjątkiem nielicznych przypadków, były daleko niewystarczające. Znajomość metodyki kontrolnej dotyczącej badania działań na rzecz poprawy jakości powietrza zaowocowała powierzeniem nam przez najwyższe organy kontroli z kilkunastu państw europejskich obowiązków międzynarodowego koordynatora kontroli w tym obszarze, w której - tak jak powiedziałem - uczestniczyło kilkanaście państw europejskich. Szanowni Państwo! Dostrzegając wpływ ochrony środowiska na życie i zdrowie obywateli, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła też kontrolę utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach. Kolejnym ważnym obszarem wpływającym na życie obywateli jest organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Poświęciliśmy temu zagadnieniu szereg kontroli w ubiegłym roku.

W innej kontroli stwierdziliśmy, że system opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, szczególnie w zakresie profilaktyki, nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupie wiekowej, o czym świadczy zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Temat ochrony zdrowia jest dla NIK-u tak ważnym zagadnieniem, że przygotowaliśmy całościowy raport, swego rodzaju megainformację, opierając się na ustaleniach z ponad 70 kontroli Izby, oczywiście w tym także tych z ostatnich lat, a także na opiniach lekarzy, dyrektorów, przedstawicieli organów założycielskich szpitali, osób zarządzających służbą zdrowia oraz [[Dzwonek]] organizacji zrzeszających pacjentów. Nasz raport spotkał się ze znakomitym przyjęciem wśród zewnętrznych ekspertów. Jest on także dostępny dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z najważniejszymi problemami występującymi w obszarze ochrony zdrowia oraz rekomendacjami NIK-u. Od wielu lat zajmujemy się w NIK-u problemami związanymi ze ściągalnością podatków, w tym podatku VAT. W 2018 r. kontynuowaliśmy kontrole w tym obszarze, doceniając większą skuteczność aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT. Troszcząc się o prawidłowe wydatkowanie środków publicznych, zainteresowaliśmy się także problemem związanym z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa i ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego. Sygnały na temat nieprawidłowości płynęły do nas m.in. z komisji sejmowych. Skontrolowaliśmy wydatki spółek Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze. Do najważniejszych nieprawidłowości zaliczyliśmy wydawanie pieniędzy na sponsoring pomimo ujemnego wyniku finansowego spółki czy sponsorowanie przedsięwzięć, które nie były ujęte w planach wydatkowania środków. Szanowni Państwo! W 2018 r. badaliśmy też funkcjonowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz wypłaty odpraw w wybranych spółkach Skarbu Państwa. Raporty są już gotowe i wkrótce trafią do Sejmu. Niektóre nasze informacje o wynikach kontroli przesyłamy do Sejmu w trybie właściwym dla informacji niejawnych. Tak było np. wtedy, kiedy sprawdzaliśmy, jak Polska jest przygotowana na zagrożenia związane z terroryzmem. Ważny i ciekawy raport w tej sprawie skierowaliśmy niedawno do Sejmu. Szanowni Państwo! Podsumowując, mogę powiedzieć, że najważniejszą rolą NIK-u jest dostarczanie parlamentarzystom, przedstawicielom władzy wykonawczej oraz - co najważniejsze - wszystkim obywatelom rzetelnej, pogłębionej i obiektywnej informacji o różnych istotnych obszarach. Wolni obywatele muszą bowiem wiedzieć, jak agendy rządowe i samorządowe wykonują swoje ustawowe zadania oraz jak wydają publiczne pieniądze. Wydaje się, że dzisiaj, 100 lat po powstaniu Najwyższej Izby Krajowej, jej znaczenie staje się jeszcze większe. W dobie szumu informacyjnego i zagrożenia celowymi manipulacjami i kreowaną dezinformacją trudno sobie wyobrazić istnienie demokratycznego kraju bez rzetelnej, pogłębionej i obiektywnej informacji dostarczanej przez niezależną instytucję odpowiedzialną za kontrolę państwa. Wysoki Sejmie! Pozostawiam Izbę w bardzo dobrym stanie, wysoko cenioną przez opinię publiczną, ekspertów zewnętrznych, instytucje międzynarodowe, dziennikarzy i parlamentarzystów, ale przede wszystkim pozostawiam Izbę, w której pracuje 1600 profesjonalistów, najlepszych w Polsce specjalistów od kontroli państwowej, znakomicie wykształconych, solidnie przygotowanych.

Dziękuję wam za tę wspólną służbę. Mogę zakończyć życzeniami kierowanymi do mojego następcy, żeby tak jak do tej pory Najwyższa Izba Kontroli była synonimem rzetelnej, wiarygodnej, obiektywnej informacji, która będzie służyć wszystkim obywatelom i parlamentarzystom w polskim Sejmie i polskim Senacie. Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Na wstępie trzeba przypomnieć, że jedyną instytucją sprawującą nadzór nad Najwyższą Izbą Kontroli jest Sejm działający in gremio oraz przez swoje organy, w szczególności przez marszałka Sejmu. Z tego względu Sejm nie może zaniedbać wykonywania tej funkcji. Dotyczy to oczywiście także wyspecjalizowanej komisji, czyli Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Powodem tego były błędy lub zaniedbania w organizacji wewnętrznej NIK, takie jak absurdalne zbiurokratyzowanie tej instytucji czy koteryjna polityka nagradzania pracowników.

W ostatnim roku naszej kadencji i jednocześnie w ostatnim roku kierowania NIK przez obecne szefostwo trzeba odnieść się do kwestii wpływu skutków woluntaryzmu kierownictwa NIK na jakość pracy tej instytucji.

Tak więc czołowe - według samej NIK - ustalenie polskiej kontroli państwowej jest niezweryfikowane, a być może wyssane z palca. Ile takich niezweryfikowanych lub nieudokumentowanych informacji znajduje się w prawie 200 raportach ukazujących się w każdym roku?

Koszty związane tylko z czasem pracy kontrolerów nad tym tematem kontroli można oszacować na kwotę grubo powyżej 300 tys. zł. Taka jest więc przybliżona cena zaczerpnięcia niezweryfikowanej informacji z filipińskiego portalu. Gdyby to był dowcip, można byłoby powiedzieć, że choroba filipińska się rozwija. Podobnie rzecz ma się z innym głośnym raportem pod nazwą: Nauczanie matematyki w szkołach.

Jedyny wniosek generalny NIK to stwierdzenie, że - w skrócie zacytuję - należy rozważyć możliwość zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. W rozdziale: Ważniejsze wyniki kontroli, a więc w źródłowej części raportu, w podrozdziale: Wyniki egzaminów zewnętrznych na temat statusu egzaminu maturalnego z matematyki nie ma ani słowa. W rozdziale pod nazwą: Synteza jest krótkie stwierdzenie, że należy rozważyć obecny status egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Nie można wskazać, że obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce danego państwa w rankingu innowacyjności gospodarki. Z kolei w rozdziale: Wnioski, przytaczając rekomendację ekspertów, wyraźnie wskazuje się na to, dla niepoznaki w przypisie, że jedna z pań ekspertek rekomendowała pozostawienie egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie podstawowym jako obowiązkowego. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której czołowy wniosek najwyższej izby jest artystyczną koncepcją kierownictwa departamentu edukacji oraz kierownictwa NIK, niemającą nic wspólnego z konkretnymi ustaleniami dokonanymi w ramach tematu kontroli. Nawiasem mówiąc, ustaleniami skądinąd dosyć ciekawymi - tymi pozostałymi. Trzeba jeszcze dodać, że omawiany tu wniosek, ten czołowy, jest sprzeczny z wieloma tezami zawartymi w samym raporcie. Znowu trzeba zadać pytanie: Ile takich bezpodstawnych wniosków albo wniosków z wątpliwą podstawą dokumentacyjną jest w raportach NIK?

W kontekście tej sprawy oraz spraw poprzednich trudno nie zauważyć, że pogoń za sensacją jest dla obecnego kierownictwa NIK ważniejsza niż rzetelny stosunek do rzeczywistości. Zastanawiająca jest zwłoka w opublikowaniu raportu.

Co to za metoda pracy? Po co fatygować kontrolerów, skoro wyniki ich pracy nie kształtują opinii i ocen NIK? W ramach tego tematu skontrolowano 21 jednostek.

Podobnie niezrozumiała zwłoka nastąpiła w związku z kontrolą: Realizacja przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych - tytuł jest dłuższy. Raport został zatwierdzony w październiku 2018 r., ale opublikowano go w pierwszej dekadzie 2019 r., a więc 5,5 miesiąca od jego zatwierdzenia i omal rok od zakończenia czynności kontrolnych. Ustalenia NIK były alarmujące, a jednak zwlekano z jego opublikowaniem, a tym samym zrezygnowano z szybkiego prewencyjnego oddziaływania raportu. To przykład niezrozumiałego manewrowania efektami pracy NIK, na pewno niesłużącego publicznemu pożytkowi. Przykładem już nie manewrowania, ale manipulowania wynikami kontroli jest raport „Zmiany w systemie oświaty”

Nawiasem mówiąc, tym razem od zakończenia czynności kontrolnych do upublicznienia raportu minęły niecałe 4 miesiące, co zresztą powinno być normą. Celem głównym tego raportu było ustalenie, czy prawidłowo i skutecznie dokonano zmian w systemie oświaty. Jednak raport nie jest odpowiedzią na to pytanie i to nie jest przypadkowe. Zabieg ten pozwolił na zminimalizowanie pozytywnych ocen Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzeba przyznać, że strategie minimalizacji NIK zastosował tu konsekwentnie, zminimalizował też krytyczne oceny podmiotów samorządowych, które były bezpośrednimi realizatorami zmian w oświacie. Oceny Ministerstwa Edukacji Narodowej dokonane przez NIK były albo nieuprawnione, albo wątpliwe. MEN przypisano odpowiedzialność za nieprawidłowe działania lub zaniechania innych podmiotów uczestniczących w procesie reformowania oświaty. W jednym przypadku ujęcie problemu i sformułowana quasi-ocena świadczą wprost o nieznajomości problematyki oświaty przez redaktorów raportu, co w praktyce oznacza niewiedzę wyższego szczebla nadzoru w NIK. Jak powiedziałem, Najwyższa Izba Kontroli z jednej strony uchyliła się od ocen potencjalnie pozytywnych, a z drugiej strony uchyliła się od krytycznych ocen innych podmiotów. Nie sposób więc nie zauważyć intencjonalności raportu, co znajduje dodatkowe uzasadnienie w nieopublikowaniu stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej wbrew wyraźnemu obowiązkowi wynikającemu z dyspozycji ustawy o NIK. Analiza treści raportów wskazuje na kiepską jakość warsztatu kontrolerskiego wyższego szczebla nadzoru w NIK, przejawiającą się m.in. w nieweryfikowaniu stawianych tez i hipotez oraz rezygnacji z ustalania związków przyczynowo-skutkowych. Nawiasem mówiąc, kwestia nieustalania przez NIK przyczyn negatywnych zjawisk wielokrotnie przy różnych okazjach pojawiała się w trakcie kolejnych posiedzeń Komisji do Spraw Kontroli Państwowej zajmującej się innymi kontrolami. Podsumowując, redakcja tego raportu została dokonana intencjonalnie, a warto dodać, że koszty związane z opłaceniem kontrolerów można oszacować mniej więcej na 1 mln zł. W ramach przeprowadzanej w 2018 r. kontroli wykonania budżetu państwa w 2017 r. w części 29., a więc dotyczącej obrony narodowej, NIK wytknął Ministerstwu Obrony Narodowej osiem nieprawidłowości, z czego trzy dotyczyły jednej sprawy, mianowicie zakupu jednostek transportu powietrznego dla najważniejszych osób w państwie. Pamiętamy, że ta kwestia nie była rozwiązywana przez kilkanaście lat. W 2017 r. na ten cel wydano kwotę ponad 727 mln zł, z czego 527 mln zł pochodziło ze środków dedykowanych przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Otóż NIK uznała, że w ten sposób pulę dedykowanych środków pomniejszono właśnie o tę kwotę, tj. o 527 mln zł, bo przedmiotowy wydatek potraktowano jako niezwiązany z obronnością Rzeczypospolitej. Tymczasem zakupione statki powietrzne nie tylko są obsługiwane przez pilotów wojskowych, a ich loty są monitorowane przez właściwe służby polskich sił powietrznych, ale część z nich ma nowoczesne środki techniczne, m.in. umożliwiające lądowanie na lotniskach wojskowych, w tym na terytoriach zagrożonych takich jak Afganistan, a nawet posiada stosowne środki obronne, a także umożliwiające dowodzenie z powietrza dużymi formacjami wojskowymi. Tak więc dokonana przez NIK kwalifikacja czynu jest rażąco błędna. Poza tym, kolokwialnie sprawę ujmując, jest ona idiotyczna. Z natury rzeczy takie osoby jak prezydent, premier, ministrowie i najwyżsi dowódcy wojskowi muszą mieć szczególną ochronę, czyli o charakterze wojskowym. Co ważniejsze, jest naszym interesem państwowym odbudowanie lotnictwa transportowego specjalnego przeznaczenia, bo w takim, a nie innym otoczeniu zewnętrznym żyjemy. Jest jeszcze ważny kontekst. Otóż częściowe sfinansowanie przedmiotowego zakupu ze środków przeznaczonych na przebudowę, modernizację i finansowanie Sił Zbrojnych nie było nowatorskim pomysłem obecnego rządu. Poprzedni rząd również planował częściowe sfinansowanie zakupu jednostek transportu powietrznego dla VIP-ów ze środków dedykowanych przebudowie i modernizacji i jakoś wówczas nie budziło to zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. Plan ten co prawda nie został zrealizowany, ale to z powodu powszechnie znanej sprawności, czyli niesprawności rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oczywiście nasuwa się pytanie o intencje organizatorów tej kontroli. Dziwnym trafem na NIK nie zrobiło żadnego wrażenia to, że rozwiązano kwestię przez lata zaniedbaną, za to uznała za rzecz oczywistą, że wydatek na samoloty pełniące funkcje obronne nie może być poniesiony ze środków służących obronie państwa. Podsumowując całość mojej dotychczasowej wypowiedzi, już tylko na tych kilku przykładach widać, jak bardzo niezadowalający jest standard pracy kierownictwa NIK. A jednocześnie widać, do jak niebezpiecznego stopnia posuwa się woluntaryzm tego kierownictwa. Powtórzę, by nie było wątpliwości, mam na myśli nie tylko prezesów, ale także tzw. radców prezesa oraz korpus dyrektorski. Dla kierownictwa NIK nie jest problemem serwowanie w raportach niesprawdzonych danych i wątpliwych hipotez oraz tez, problemem nie jest też bardziej albo mniej subtelne manipulowanie wynikami kontroli z niemałym trudem przecież osiąganymi przez kontrolerów przeprowadzających badania w terenie. Jest to przede wszystkim rezultat wewnętrznej destrukcji Najwyższej Izby Kontroli.

Z żalem trzeba powiedzieć, że prezesi NIK, może z jednym wyjątkiem, przynajmniej moim zdaniem, nawet nie mieli zamiaru dokonać w tym zakresie zauważalnej korekty. Przez kolejne lata zwracaliśmy uwagę na absurdalny formalizm pracy kontrolerskiej, który sprzyja obniżaniu standardów pracy Najwyższej Izby Kontroli. W sprawozdaniu za 2018 r. wyszczególnia się krótko takie osiągnięcia zarządcze jak: wprowadzanie zasad opracowania kluczowych dokumentów pracy NIK, zmodyfikowanie wzorów programów kontroli i raportów NIK oraz ujednolicenie sposobów prezentacji wyników kontroli. Taki sam skutek, tj. zerowy, przyniósł system zapewnienia jakości. Dokonywanie biurokratycznego przeglądu jakości zadania kontrolnego nie zapobiegło opisanym wyżej zjawiskom negatywnym, a przecież w tym procesie weryfikacji biorą udział dziesiątki osób. To negatywny skutek stawiania na niepragmatyczne procedury, a nie na ludzką odpowiedzialność i uczciwość. W omawianym sprawozdaniu poinformowano, że zakończono pracę nad stworzeniem modelu kompetencyjnego zawodowych kontrolera. Jak widać, ten papierowy model kompetencji nie zapobiegł zjawiskom wyżej opisanym. Powtórzę: patetyczne, papierowe ustalenia nie zastąpią osobistej odpowiedzialności i uczciwości, a tym bardziej odwagi. Jak wiadomo, katowicka prokuratura wystąpiła z aktem oskarżenia i wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK.

Przypomnę, że w poprzednich 3 latach ukazaliśmy bezmyślny styl zarządzania Najwyższą Izbą Kontroli. Zmian nie ma, a skutki obniżonych standardów pracy są coraz bardziej widoczne. W imieniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej stawiam podobnie jak w minionych latach wniosek o nieprzyjęcie sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli za 2018 r. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 10-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 5-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość wystąpi pan poseł Wojciech Szarama. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Chciałbym podkreślić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a ono też nie jest prezentowane po raz pierwszy: dla nas bardzo ważną rzeczą jest to, że przeciwko panu prezesowi został skierowany akt oskarżenia dotyczący popełnienia przestępstw związanych z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli. Sejm, Wysoka Izba nie ma możliwości dokonania jakiejś indywidualnej oceny, indywidualnego zwrócenia regulaminowej uwagi panu prezesowi. Raz w roku odbywa się rozpatrywanie sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli. Z całą mocą chciałbym właśnie podkreślić, że tego sprawozdania przedłożonego Sejmowi przez pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przyjąć nie może z tych wszystkich względów, które zostały wymienione wcześniej. Jest to oczywiście sytuacja bardzo trudna, nie tylko dla Wysokiej Izby, dla poszczególnych klubów parlamentarnych czy ugrupowań politycznych, jest to sytuacja trudna dla całej Polski, dlatego że na działalność tego najwyższego organu kontroli w państwie polskim pada pewien cień, którego nie sposób nie zauważyć. Oczywiście oprócz tych uchybień, błędów, o których mówił pan poseł sprawozdawca, na co dzień spotykaliśmy się z pracą, z poszczególnymi kontrolami, z poszczególnymi informacjami z przeprowadzanych kontroli, które oceniamy dobrze i które rzeczywiście są potrzebne i pomocne w funkcjonowaniu państwa, w funkcjonowaniu rządu. Pozwalają korygować pracę w poszczególnych ministerstwach, w samorządach, w bardzo wielu ważnych obszarach naszego życia: ekonomicznego i społecznego. Trzeba po prostu podziękować za to wszystko, co zostało zrobione dobrze, pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy, jak to zostało dzisiaj powiedziane, po zakończeniu tej kadencji prezesa będą funkcjonować i będą pracować dalej dla dobra państwa polskiego. Ale ta baza, która oparta jest na tradycji i na umiejętnościach pracowników Najwyższej Izby Kontroli, z pewnością będzie nadal wykorzystywana i mam nadzieję, że będzie służyła państwu polskiemu.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu mojego klubu przedstawić opinię co do sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, ale myślę, że zanim to zrobię, to muszę chyba przypomnieć o misji NIK-u, czym jest w ogóle Najwyższa Izba Kontroli, bo mam wrażenie, że od kilku lat Prawo i Sprawiedliwość, dokładnie odkąd rządzi, o tym zapomniało. NIK to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika grosza publicznego. Od 100 lat NIK ocenia funkcjonowanie państwa, gospodarowanie środkami publicznymi, pokazuje błędy aparatu państwa, ale również pokazuje, jak je naprawić. Ja jeszcze raz podkreślę, jest ona apolityczna, obiektywna, niezależna i rzetelna. Mówiąc krótko, Najwyższa Izba Kontroli to nie telewizja publiczna, a prezes Kwiatkowski to nie prezes Kurski. Zacznijmy od kontroli Funduszu Sprawiedliwości działającego na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Kontrolerzy krytykują zasadność przyznawania milionów złotych na projekty, które nie mają żadnego związku z celami funduszu. NIK ustalił także, że wiele organizacji dostało milionowe dotacje mimo braku odpowiedniego doświadczenia. Wszyscy pamiętamy choćby wczoraj przez media pokazywane 24 mln zł na kamizelki odblaskowe. Cel może słuszny, ale czemu kosztem ofiar? Czemu z pieniędzy, które mają pomagać ludziom pokrzywdzonym? NIK skontrolował 14 konkursów i naborów ofert na łączną wartość prawie 40 mln zł. Kto dostał pieniądze? Kto był beneficjentem? Ojciec Tadeusz Rydzyk, naprędce zakładane fundacje i stowarzyszenia związane z ludźmi ministra Ziobry, Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości.

Mimo że zostały złożone odpowiednie oświadczenia, nie zostały one później zatwierdzone i nie zapadła żadna decyzja o zwrocie tych pieniędzy. Jest to bezwzględnie zaniechanie, które narusza dyscyplinę finansów publicznych. W ocenie NIK niewielka część ofiar przestępstw w stosunku do skali przestępstw otrzymuje z funduszu alternatywną i skuteczną pomoc. Przykład? Ustawa kompensacji przestępstwowej, która miała stanowić wsparcie dla 12 tys. ofiar najcięższych przestępstw, przestępstw związanych z narażeniem życia i zdrowia. 30 osób. A wy wydajecie lekką ręką 24 mln na kamizelki odblaskowe. Między innymi zlikwidowano również pomoc prawną, psychologiczną udzielaną poprzez Internet czy infolinię. Najpierw państwo PiS nie potrafiło ochronić tych ludzi, teraz nie potrafi im pomóc. Kolejna kwestia, nieodpłatna pomoc prawna. Co wyszło z ustawy? W konsekwencji 3/4 potencjału systemu nie zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, których chyba nikt nie podważy, przeciętnie na jeden punkt przypada jedna porada dziennie. Komentarz chyba zbędny. Bardzo ciekawe wnioski NIK wyciąga również z kontroli spółek Skarbu Państwa.

Ale jeszcze ciekawsza jest kontrola, która objęła tylko 20 spółek Skarbu Państwa. Większość z nich mimo wydatkowania ogromnych sum nie przestrzegało ustanowionych przez siebie zasad i procedur w tym zakresie. I mały cytat: W mediach cyklicznie pojawiają się zarzuty, że sponsoring wykorzystywany jest jako parawan do finansowej rekompensaty udzielanej konkretnym podmiotom, np. za ich zaangażowanie w kampanię wyborczą określonego kandydata lub partii. Co wykazała kontrola? Działania lub zaniechania władz w 13 skontrolowanych spółkach stworzyły ryzyko niegospodarności, a w trzech spółkach doprowadziły do poniesienia niegospodarnych wydatków na prawie 660 tys. Dodam, że część tych spółek, które były sponsorami, ma ujemny wynik finansowy. Zresztą też z tej kontroli wynika, że 20% spółek Skarbu Państwa, 100 z nich, jest dzisiaj w bardzo kiepskiej sytuacji finansowej, jest w likwidacji lub w upadłości. To jest karuzela stanowisk, milionowe odprawy i zarządzanie menedżerów państwa Prawa i Sprawiedliwości. NIK pokazuje prawdziwy stan państwa, jego dzisiejszy rozkład. To nie papla propagandowa, jaką dzisiaj codziennie serwujecie poprzez telewizję publiczną narodowi.

Lista zarzutów tylko z tej jednej rocznej kontroli jest bardzo długa, ale do was nie docierają te argumenty. Wy znowu nie przyjmujecie tego sprawozdania i atakujecie personalnie pana prezesa, nie odnosząc się do jego pracy. Panie Prezesie!

Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Zaproszeni Goście! Najwyższa Izba Kontroli to jedyny taki organ kontroli w państwie, którego wszyscy w administracji publicznej się obawiają - to słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy wypowiedziane podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z prezesem Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofem Kwiatkowskim oraz szefami europejskich najwyższych organów kontroli w czerwcu tego roku. Jak przychodzi Najwyższa Izba Kontroli na kontrolę, wszyscy sztywnieją, bo to jest tak ważna kontrola, rzetelna, do której trzeba się w sposób bardzo profesjonalny odnieść, wymagane są najwyższe standardy. I rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli i jej kontrolerzy najwyższych standardów przestrzegają - stwierdził prezydent. Uważam, że Najwyższa Izba Kontroli odgrywa ogromną rolę nie tylko jako organ kontrolny w Polsce, ale również w Europie i na świecie. Tegoroczne sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli przypada w szczególnym okresie, a mianowicie w okresie, kiedy obchodzimy stulecie istnienia Najwyższej Izby Kontroli. Twórcy najwyższego organu kontroli, chcąc uzyskać wiarygodną kontrolę, ustawowo zagwarantowali niezależność Najwyższej Izby Kontroli, jej kolegiantom oraz wszystkim kontrolerom. Chciałabym powiedzieć, że rocznie kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzili kilkaset kontroli z różnych dziedzin. Tylko w 2018 r. publikowano raporty dotyczące smogu w Polsce, działań komisji ds. błędów medycznych czy stanu kąpielisk. Analizowano także kontrole żywności, ryzyko zakażeń w szpitalach czy nadzór w państwowych spółkach, o których szerzej mówił poseł Gierada.

Jest to po prostu zwyczajna krytyka dla krytyki bez twardych, mocnych argumentów, bez merytorycznego uzasadnienia. Przypomnę, że komisje sejmowe przyjęły ten dokument bez zastrzeżeń. Wręcz przeciwnie, wiele z tych komisji opiniowało go pozytywnie i uznawało informacje za przydatne. Dlatego uważam, że jest to niesprawiedliwe, nieuczciwe, aby oskarżenia dotyczące prezesa Najwyższej Izby Kontroli rzutowały na całą Izbę. Nie będę się odnosiła do słów koreferenta z Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Chciałabym również zaznaczyć i nadmienić, że dobrze by było, gdyby regulamin Sejmu nakazywał większe zaangażowanie komisjom sejmowym, aby wnioski de lege ferenda, wnioski pokontrolne znajdowały odzwierciedlenie w zmianach przepisów ustaw. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska jest za przyjęciem sprawozdania. Z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować całej kadrze Najwyższej Izby Kontroli za rzetelną pracę na rzecz naszego kraju, także poza naszymi granicami, a panu prezesowi podziękować, że wyniósł Najwyższą Izbę Kontroli na wyżyny, bowiem Najwyższa Izba Kontroli nie tylko uzyskała wśród respondentów bardzo wysoką opinię, ale również na arenie międzynarodowej. W takim razie pan poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów.

Na początku tego roku, na początku 2019 r., a dokładnie w lutym, Najwyższa Izba Kontroli obchodziła stulecie powstania. W dekrecie powołującym Izbę zapisano zasady i prezentowano wartości: uczciwość, rzetelność, sumienność, dociekliwość, obiektywizm, które to zasady, jestem o tym głęboko przekonany, przyświecały również w pracy inspektorom i pracownikom Izby również w roku 2018, w którym realizowali plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na ten właśnie 2018 r. Pan prezes Najwyższej Izby Kontroli we wstępie do tego sprawozdania, które dzisiaj omawiamy, pisze wprost, że te wartości, te zasady okazały się ponadczasowe i nadal obowiązują w Najwyższej Izbie Kontroli. Kluczowe jest również, moim zdaniem, stwierdzenie, i tu dosłownie cytuję zdanie ze wstępu, że dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego, podkreślam: niezależnego, od władzy wykonawczej organu kontroli stojącego na straży publicznych pieniędzy.

Ocenianie, oczywiście ocenianie bardzo negatywne, o czym słyszeliśmy, kontroli w zakresie reformy edukacji, kontroli odnoszących się do nauczania matematyki. A to, że te kontrole, te raporty nie znalazły się w sprawozdaniu, które właśnie teraz oceniamy, które jest przedmiotem oceniania, tak mówiąc szczerze, tym gorzej dla tegoż sprawozdania. Potrzebne było uzasadnienie tezy? Bardzo proszę, przytoczymy dokument niezawarty wprawdzie w sprawozdaniu, ale to już mniejsza o to.

Jeszcze raz przytoczę kluczowe zdanie: dla sprawnego funkcjonowania państwa niezbędne jest istnienie kompetentnego i niezależnego od władzy wykonawczej organu kontroli, stojącego na straży publicznych pieniędzy. NIK dba o zgodne z prawem gospodarne, celowe wykorzystanie i rzetelne rozliczenie środków publicznych i jako obywatel życzyłbym sobie, by tak było w następnych latach. Dla trwałości i siły państwa polskiego. Wysoki Sejmie! Misja służenia państwu i obywatelom wyraża się między innymi poprzez informacje z kontroli, zawierające nie tylko ustalenia stanu faktycznego, ale również wnioski istotne dla poprawy funkcjonowania kontrolowanych obszarów. Najwyższa Izba Kontroli koncentruje się przede wszystkim na nieprawidłowościach o charakterze systemowym, na działaniach administracji publicznej oraz na czynnikach zagrażających prawidłowej realizacji celów państwa i problemach szczególnie dotkliwych dla obywateli. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzili w 2018 r. 111 kontroli planowych, 91 kontroli doraźnych, w tym oczywiście kontrole wykonania budżetu państwa za rok 2017, którą objęto wszystkich dysponentów w części budżetowej państwa: kolegia samorządowe, sądy apelacyjne, państwowe fundusze celowe, wybrane agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki realizujące wydatki publiczne, w tym jednostki spoza sektora finansów publicznych. W ramach aktywności kontrolnych w 2018 r. wykonano 2325 kontroli jednostkowych realizowanych w 1633 podmiotach. I to właśnie obrazuje wymiar pracy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli przedłożyła Sejmowi 190 informacji o wynikach kontroli planowych i doraźnych, a jej przedstawiciele uczestniczyli w 316 posiedzeniach komisji, w tym 20 posiedzeniach komisji branżowej, Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Najwyższa Izba Kontroli na podstawie wyników kontroli formułuje wnioski pokontrolne, które mogą sugerować konkretne zmiany w kontrolowanych jednostkach, i tak zwykle jest, jak też dotyczą całokształtu badanych zagadnień i mają właśnie charakter systemowy. Warto podkreślić, że wnioski Najwyższej Izby Kontroli stają się inspiracją do zmian w prawie często już w trakcie kontroli. Właśnie na ten temat, na temat propozycji zmian legislacyjnych, kilka zdań oceny.

Najwyższa Izba Kontroli sformułowała łącznie 535 wniosków de lege ferenda, spośród których zostało zrealizowanych 149, a kolejne 27 wniosków z tego okresu jest obecnie w procesie legislacyjnym. Przytaczam te liczby, tę statystykę, bo uważam, że to jest sedno pracy takiej instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli, ale również dlatego, by po raz kolejny zadać kłam opiniom wygłaszanym tu w latach poprzednich, w latach ubiegłych, opiniom nieprawdziwym i niesprawiedliwym o tym, jakoby NIK była instytucją, i tu cytuję: z głową odwróconą w tył. To jak ocenić te właśnie formułowane wnioski? Wysoki Sejmie! Prezentując te kilka ocen, kilka wniosków chcę jeszcze raz podkreślić, że fundamentalnie nie zgadzamy się z opinią zaproponowaną przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej. Na gruncie rzetelnej, podkreślam, rzetelnej oceny pracy NIK w 2018 r. i oceny sprawozdania z działalności NIK, którym się przecież dzisiaj zajmujemy, będziemy za przyjęciem tego sprawozdania, właśnie tak jak zaznaczyłem, na gruncie rzetelnej, obiektywnej oceny, a nie na płaszczyźnie politycznej. Chętnych, którzy zechcą tę sferę polityczną zgłębić, zachęcam do przeczytania protokołu z posiedzenia komisji, do obejrzenia posiedzenia komisji w dniu 12 czerwca, kiedy te tezy były formułowane. A na zakończenie bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu prezesowi, kierownictwu Najwyższej Izby Kontroli i wszystkim zatrudnionym pracownikom za ogromną, rzetelną pracę, za rzetelne podejście do ważnych społecznych i gospodarczych zjawisk. Bardzo dziękuję za uwagę.

Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Kontrola państwowa opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji. Panie Sprawozdawco!

To było polityczne wystąpienie na zamówienie. Było zero rzetelności i tak też należy oceniać wniosek komisji, który został sformułowany. Jako wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że wszystkie wyniki kontroli, wszystkie raporty przedstawiane przez Najwyższą Izbę Kontroli były oceniane absolutnie pozytywnie i na każdym posiedzeniu komisji dziękowaliśmy Izbie za to, że traktuje politykę senioralną, prognozy demograficzne w swoich kontrolach jako priorytet. Rozumiem, że jest problemem dla rządu PiS, jeżeli Najwyższa Izba Kontroli formułuje taki wniosek, że w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej nie stworzono narzędzi do skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin. Tak, to boli, bo wydajecie 400 mln na IPN, a nie chcecie dać 10 mln na program alzheimerowski. Panie Prezesie! To jest ten moment, w którym chciałbym panu bardzo serdecznie podziękować za tę pracę, jaką pan wykonywał razem ze swoim zespołem, razem ze swoimi zastępcami i całą Izbą, na rzecz polityki senioralnej. Ta problematyka została dostrzeżona w działaniach Izby, jest zauważana przez seniorów i buduje pana szacunek, który będzie pamiętany. Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Otóż chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz.

Otóż poprzednie kontrole dotyczące podobnych zagadnień z zakresu geologii i polityki surowcowej uwzględniały ustosunkowanie się głównego geologa kraju do wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Nie zmieniło się prawo, nie zmienili się ludzie, nie zmieniły się argumenty, jedynie zmieniła się opcja, jaką pan prezes prezentował.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Prezesie! Chciałbym zapytać o proces, który towarzyszy powstawaniu tych zjawisk, czyli o proces decyzyjny. Chcę zapytać, czy i w jakiej przestrzeni państwo kontrolujecie proces decyzyjny w odniesieniu do skutków tych decyzji, czyli tych kwestii, które są potem przedmiotem państwa kontroli albo innych instytucji do tego powołanych przez państwo polskie. Dziękuję.

Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie o raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący promieniowania elektromagnetycznego. Chciałbym zapytać, czy w Polsce istnieje i jak funkcjonuje system monitoringu zdrowia w pobliżu źródeł promieniowania elektromagnetycznego i czy jest zapewniona ochrona zdrowia ludzi przed tym promieniowaniem?

Czy jednostki administracji publicznej są przygotowane do rzetelnej kontroli promieniowania elektromagnetycznego?

Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Prezesie! No, serce się ściska, kiedy słyszy się o manipulacji danymi przez NIK. Panie prezesie, w związku z tym chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15-procentowego udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest zagrożone. Czy prawdą jest, że w 2016 r. wskaźnik ten był najniższy i wynosił 11%, i był najniższy od 2013 r. Czego rząd nie zrobił? Kolejna sprawa. Od początku kadencji rząd PiS-u przystąpił do likwidacji kopalń, likwidacji miejsc pracy na Śląsku. Postawił na rekordowy import węgla, w tym przede wszystkim z Rosji. Postawił na utrzymanie miejsc pracy rosyjskich górników. Postawił na trucie Polaków rosyjskim węglem. Większość środków przeznaczonych na ten cel, czyli prawie 7 mld zł, trafiało i będzie trafiać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Chciałem pana prezesa zapytać, kiedy NIK przystąpi do kontroli tej spółki. Kilku członków zarządu otrzymało zarzuty, [[Dzwonek]] można powiedzieć, za korupcję.

Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Najwyższa Izbo Kontroli! Niech to sformułowanie, choć zawarta jest w nim tautologia, będzie podziękowaniem dla pana prezesa, jego najbliższych współpracowników i ponad 1500 pracowników NIK za minione lata, za 6 lat kadencji.

Myślę, że był to czas wykorzystany, aby udoskonalić działanie NIK, bo przecież w każdym przypadku, również w tym przypadku, są obszary do doskonalenia, choćby kwestia badania efektywności funkcjonowania całego sektora publicznego.

Wykazaliście wiele nieprawidłowości. Myślę że kwestia Funduszu Sprawiedliwości, kwestia wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa czy przeznaczenie bajońskich sum [[Dzwonek]] przez te spółki na dziwny sponsoring to są te kwestie. Pani poseł Elżbieta Stępień, klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Dlatego chciałam zapytać odnośnie do sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za 2018 r., chodzi o kontrolę nauki, nauczania matematyki w szkołach, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, realizację przez samorządy zadań związanych z organizacją imprez masowych i biegów ulicznych, zmian w systemie oświaty. Czy są to prawdziwe zarzuty czy jest jakaś inna opinia? Pani poseł Agnieszka Hanajczyk, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo, że najpierw podziękuję.

Dziękuję całemu zespołowi i cieszę się, że na stulecie została dostrzeżona ta bardzo dobra umiejętność strzeżenia grosza publicznego. Chcę również powiedzieć, panie prezesie, że wśród setek kontroli bardzo dziękuję za kontrole bliskie mojemu sercu, m.in. badanie bezdomności zwierząt, wykonywania opieki nad zwierzętami. To są takie kontrole, które zdecydowanie poprawiają możliwość podejmowania działań.

Mieszkańcy Zgierza pytają mnie, piszą do mnie maile, czy mogą być spokojni, czy mogą być pewni, że ta sprawa w żaden sposób nie ucieknie, nie zostanie zakopana, zamieciona pod dywan. Ja oczywiście przekonuję, że jest to bardzo ważna, istotna kontrola.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, tak jak cały Sejm, jest przekonany, że Najwyższa Izba Kontroli musi funkcjonować w sposób całkowicie niezależny, a kontrolerzy muszą się opierać na swojej wiedzy, na swoich przekonaniach i na informacjach, które w trakcie kontroli zdobywają. A więc te słowa, które tutaj padły, że są jakieś kontrole niewygodne dla naszego klubu parlamentarnego, są całkowicie błędne. Nikt bardziej niż Prawo i Sprawiedliwość nie jest zainteresowany tym, żeby kontrole Najwyższej Izby Kontroli były kontrolami pełnymi, obiektywnymi i jeśli będą one czasami niedogodne dla kogoś z rządzących, to nie zmienia postaci rzeczy. Każda kontrola, która przyczyni się do lepszego funkcjonowania określonego segmentu państwa polskiego, będzie przez nas mile widziana. Wczoraj na posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podziękowałem panu prezesowi za kontrolę podjętą doraźnie, o której przed chwilą mówiła pani poseł Hanajczyk.

Dziękuję. Jako pierwszy odpowiadać będzie na pytania zadane w tym punkcie prezes Najwyższej Izby Kontroli pan Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Muszę powiedzieć, że w tegorocznym wystąpieniu pana posła Dziuby niestety pojawił się nowy element. Tym nowym elementem nie jest już tylko negatywna oceny kierownictwa. Tym nowym elementem jest negatywna ocena także kontrolerów. Do mojej negatywnej oceny już się przyzwyczaiłem, ale jest próba negatywnej oceny pracowników Najwyższej Izby Kontroli, zacytuję, z uwagi na, jak to powiedział pan poseł, manewrowanie pracami NIK-u w kontekście różnej publikacji wyników kontroli.

Powinien pan jako ostatni stawiać taki zarzut z bardzo prostego względu - regulamin Sejmu w art. 126 mówi, że przedkładane Sejmowi przez Najwyższą Izbę Kontroli sprawozdanie Sejm rozpatruje nie później niż w terminie 3 miesięcy od jego doręczenia posłom. Sprawozdanie z działalności NIK-u wpłynęło do Sejmu w marcu tego roku. Państwo naruszyliście regulamin Sejmu. Jeżeli ktoś manewruje jakimiś efektami, wynikami prac, łamiąc regulacje, które w tym zakresie obowiązują, to pan jako wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i ten, który co roku opiniuje nasze sprawozdanie, powinien być pierwszym, który powinien powiedzieć: przepraszam za to, że złamałem przepisy prawa. Niestety w tej swojej krytyce pan poseł posunął się dalej. Niezadowalający standard dzisiejszej pracy NIK-u odnosi się, co wyraźnie podkreślam, do szczebla kierownictwa, ale mam na myśli nie tylko prezesów NIK-u, ale także tzw. radców prezesa. To nie są tzw. radcy prezesa. To są radcy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. I każdy z kontrolerów NIK-u, niezależnie od tego, czy zajmuje stanowisko inspektora, specjalisty, doradcy, radcy czy dyrektora, zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie. Martwię się tymi wypowiedziami, bo nie ukrywam, że domniemywam, że za chwilę się okaże, że dla poprawy sytuacji najlepiej będzie odwołać dyrektorów, radców, a może cały korpus kontrolerski, i za rok okaże się, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Najwyższa Izba Kontroli już będzie funkcjonować wspaniale, a pan będzie tym, który będzie przedstawiał opinię o przyjęciu jej sprawozdania. Mówię o tym, bo pan poseł mówił i dzisiaj, i na posiedzeniu komisji: Najwyższej Izbie Kontroli wyrwano mniej więcej 18 lat temu zęby i pazury. Ten proces destrukcji w NIK-u zachodzi przez ten okres. Będę bronił dorobku wszystkich prezesów Najwyższej Izby Kontroli. Będę bronił Janusza Wojciechowskiego, który w 2001 r. pełnił jeszcze funkcję prezesa NIK-u, a dziś jest polskim przedstawicielem w ETO, Mirosława Sekuły, byłego prezesa i byłego wiceministra finansów, i Jacka Jezierskiego, który na to stanowisko został wybrany głosami posłów PiS-u. Niech pan nie dezawuuje dorobku Najwyższej Izby Kontroli, wszystkich jej kontrolerów i wszystkich prezesów, którzy na tym stanowisku byli przede mną. Nigdy nie patrzyłem na legitymację partyjną. Szanowałem każdego ze swoich poprzedników, niezależnie od tego, jakimi głosami i jaką większością był wybierany w Sejmie, bo tego typu instytucja jak niezależny organ kontroli przede wszystkim wymaga stabilności, szacunku i poczucia, że kontroler ma prawo formułować nawet negatywne opinie, jeżeli jest to uzasadnione stanem faktycznym.

Jeżeli to się kryje za intencjami pana słów, to jest to najczarniejszy możliwy scenariusz dla niezależnego organu kontroli.

Szanowni Państwo! Po raz kolejny argumentem, który się podaje w kontekście oceny sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, jest ocena mojej osoby. Przypominam, że jest coś takiego jak domniemanie niewinności. Przypomnę, że w 2015 r., natychmiast po wątpliwościach prokuratury, ja złożyłem do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu z prośbą o skierowanie sprawy do sądu. Niech pan zada sobie pytanie: Dlaczego ta sprawa trwa tyle lat, a prokurator jako świadków zgłasza osoby, które czytały w Internecie o nieprawidłowościach w NIK-u? Bo nie mi. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem pana poinformować. Proces trwa grubo ponad rok. Na pierwszym posiedzeniu sądu sąd wydał postanowienie o przekazaniu całego materiału dowodowego w tej sprawie przez prokuraturę. Nie pociętych rozmów - wszystkich rozmów i w całości. Jest mi po prostu wstyd za to, że po raz kolejny państwo przywołujecie ten argument.

Tak, stwierdziliśmy w wyniku naszej kontroli, że rzeczywiście instytucje publiczne nie sprawują rzetelnego nadzoru w zakresie ewentualności zagrożenia czy też braku tego zagrożenia w kontekście funkcjonowania np. masztów telefonii komórkowej. Kolejne pytanie dotyczyło OZE, czyli energetyki odnawialnej.

O reformie oświaty już mówiłem. W kontekście reformy związanej z egzaminem z matematyki: podstawa tego wniosku. Pomijam już to, że w systemach edukacyjnych, które dzisiaj są oceniane jako jedne z najlepszych na świecie - w Europie to jest system w Finlandii, na świecie - w Singapurze - zrezygnowano z obowiązkowego egzaminu z matematyki dla wszystkich, ograniczając ten egzamin jako obowiązkowy tylko dla tych, którzy w przyszłości chcą się kształcić na kierunkach związanych z naukami ścisłymi. To jest do dyskusji, oczywiście każde państwo decyduje o swoim systemie edukacji. Pan niestety po prostu mija się z prawdą, mówiąc, że to jest jedyny wniosek. Tutaj jest pięć wniosków skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wniosek, który mówił o tym, żeby rozważyć zawieszenie egzaminu z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich, podkreślam, polegał tylko i wyłącznie na tym i wynikał z tego, że zakres nauczania, sposób nauczania matematyki w szkołach dzisiaj niestety jest taki, że umiejętności matematyczne uczniów zamiast się poprawiać pogarszają się. Chętnie służę różnymi statystykami w tym zakresie, jeżeli będziecie państwo zainteresowani. Szanowni Państwo!

My dysponujemy wynikami doraźnych kontroli przeprowadzonych przez inspekcję sanitarną, inspekcję handlową artykułów rolno-spożywczych. W trakcie tych kontroli były badane poszczególne artykuły spożywcze.

Czy ktoś stał przez cały rok przy polskiej statystycznej rodzinie? Tak jak nie stoi się przez 365 dni w roku przy autostradzie, badając pomiar hałasu. Pobiera się próbę i pan jako były kontroler Najwyższej Izby Kontroli powinien wiedzieć o tym, że w taki sposób przeprowadza się pewne badania. Co do informacji związanej z zakupem samolotów służących do zabezpieczenia transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie należy zaznaczyć, że nieprawidłowość w zakresie zakupu samolotów została stwierdzona podczas kontroli wykonania budżetu państwa w roku 2017. Znowu pan manipuluje informacjami.

I oczywiście pomijam już to, że nie odniósł się pan merytorycznie do tego, co stwierdziliśmy, bo należy zaznaczyć, że NIK nie kwestionowała i nie kwestionuje zasadności zakupu samolotów dla VIP-ów, a jedynie stwierdziła naruszenie zasady legalności przy wydatkowaniu środków publicznych przeznaczonych na wydatki obronne, albowiem zgodnie z uchwałą samej Rady Ministrów zakup samolotów dla VIP-u miał być zrealizowany przez coroczne zwiększanie limitu wydatków obronnych ponad minimalny poziom określony w art. 7 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.

Jego zastrzeżenia były dwukrotnie przedmiotem pracy Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Ustawa o NIK jest jednoznaczna.

Żałuję, że pan już nie jest ministrem, bo by pan formalnie dostał tę odpowiedź, oczywiście dostanie pan ją także do wiadomości. Od strony formalnej ustawa o NIK-u wyraźnie mówi: zastrzeżenia zgłasza albo kierownik jednostki, albo osoba, która posiada stosowne upoważnienia. Pana upoważnienie było nieprawidłowe i pan o tym wie. Rozumiem, że nie zgadza się pan z całym kolegium Najwyższej Izby Kontroli, przyjmuję to do wiadomości. Mówi się: trudno, chociaż warto byłoby chociaż raz przeczytać dokładnie ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Szanowni Państwo!

Dlatego muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, że po raz kolejny wracamy do tej sprawy. Przechodzę do kolejnych pytań. Pani poseł Stępień pytała o kontrolę dotyczącą matematyki, już się do tego odnosiłem, dodatków do żywności, reformy oświaty czy biegów masowych. Mam nadzieję. Jedynym kryterium, którym się kierujemy, to jest oczywiście zakończenie kontroli, a później moi współpracownicy muszą jeszcze przygotować informację o wynikach kontroli przed jej opublikowaniem. Tym się kierujemy, ogłaszając poszczególne raporty. Rzeczywiście czasami to trwa odrobinę czasu, ale nie ma w tym żadnych intencji, które by miały jakiś inny charakter niż taki, [[Dzwonek]] żebyście państwo mieli rzetelną i wiarygodną informację. Na koniec podsumuję jednym zdaniem. Mam nadzieję, że dzisiejsze wypowiedzi nie są przygotowaniem do zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, bo ta instytucja, jak pokazują opinie międzynarodowe, badania Polaków i opinie ekspertów, wymaga mądrej kontynuacji, a nie głupiej rewolucji. Chęć zabrania głosu zgłosił również sprawozdawca komisji pan poseł Tadeusz Dziuba.

Pani Marszałek! Pozwolę sobie ustosunkować się do niektórych wypowiedzi, w szczególności wypowiedzi pana prezesa. Może jako takie charakterystyczne dla większości pytań wybiorę pytanie pana posła Gierady, ponieważ podał pan przykłady, z których dowodnie wynika, że nikt nie krępuje działań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Z ustaleń wynika - odwołuję się do tych przykładów, które pan podał - że należy skarcić - przepraszam za kolokwializm - rząd i nie ma na to reakcji negatywnej. Ja nie o tym mówiłem, panie pośle i szanowni inni pytający, mówiłem o czymś zupełnie innym. Mówiłem o błędach warsztatowych, o manipulacjach wynikami kontroli, czyli krótko mówiąc, o praktykach nagannych. Możemy się cieszyć, że Najwyższa Izba Kontroli może dokonywać ustaleń i ocen w sposób swobodny, to jest niewątpliwie pozytyw, ale nie możemy akceptować tego, że w ramach tej swobody odwołuje się do praktyk, które są najzwyczajniej w świecie naganne. To jest bardzo dyplomatyczne określenie. Przy okazji zwracam uwagę na to, że nikt z państwa nie zakwestionował konkretów, które podałem, bo ich się nie da zakwestionować, to są fakty. Możecie państwo ewentualnie powiedzieć, że te naganne fakty związane z funkcjonowaniem Najwyższej Izby Kontroli dotyczą jakiegoś małego procenta kontroli. Nikt tego nie policzył, bo nikt tych wad nie policzy, ale proszę państwa, Najwyższa Izba Kontroli jest jedyną instytucją tego typu w Polsce, jest unikalną instytucją w Polsce i ona musi być poza podejrzeniami. Takich praktyk stosować nie można.

A rzecz jest niebagatelna, bo jeszcze raz zwracam uwagę: odwoływałem się do kontroli, których nie wybraliśmy z jakiejś puli - wybraliśmy do tej analizy kontrole, które komentowali dziennikarze, obywatele na różnych portalach internetowych itd. Tak więc sytuacja jest groźna, proszę państwa, m.in. dlatego, że niestety przez wiele, wiele minionych lat Sejm nie zachował czujności i nie monitorował wbrew obowiązkowi, jaki na nim ciąży, tego, jaka jest jakość pracy Najwyższej Izby Kontroli.

Nie nas, tylko kontrolerów. A więc to jest sprawa jasna. Nie będę mówił o tym, że nie jestem organizatorem prac Sejmu.

Odwoływał się pan też do przywołanej przeze mnie kontroli zmian w systemie oświaty, starając się wywrzeć wrażenie, że domysły sprawozdawcy miały wpływ na tę ocenę. No, proszę państwa, to jest już skrajna nieuczciwość. Dlaczego należało o tej kontroli i o tym raporcie mówić? Zrealizowano może jeden, a raczej, moim zdaniem, pół. Główny cel kontroli w ogóle nie został zrealizowany. Państwo planujecie kontrolę z jakimś zamysłem, określacie cel kontroli, a potem tego celu nie realizujecie. To jest w porządku? Od razu mówię: pracy kierownictwa, bo przecież kontrolerzy, ci, którzy chodzą na kontrole, jakiś materiał dowodowy przynieśli. Państwo z tych trzech celów na pewno nie zrealizowaliście dwóch, a moim zdaniem - dwóch i pół.

Bardzo przepraszam, tak pan powiedział. Tak pan powiedział, proszę temu nie zaprzeczać. Ale gdzie jest honor, panie prezesie? Pan kieruje unikalną instytucją.

Jakie? Jakie pan ma poczucie honoru, tośmy przed chwilą właśnie usłyszeli. Mówiąc o tej kontroli nauczania matematyki, powołał się pan na przykład Finlandii, więc nieśmiało, tak tylko w aneksie, mówię, że właśnie Finlandia w tej chwili wycofuje się ze swojego wieloletniego i wielokrotnie chwalonego systemu edukacji. Ale dajmy temu spokój.

Ona jest naprawdę interesująca.

Macie państwo zamiłowanie do tego, żeby żonglować sensacjami, a nie żeby monitorować sposób funkcjonowania państwa. Kontrolerzy umieją to robić, ale państwo jakoś o tym zapomnieliście.

No na miłość boską, przecież to jest żart.

To już naprawdę jest zabawne.

Ona tam jest. A więc, panie prezesie, to nie komisja kontroli państwowej, nie mówiąc już o mnie, dokonuje nadużyć, tylko pan w argumentacji, która jest nierzetelna, oparta na znanych metodach erystycznych, czyli fałszowaniu sporów.

który jakoś, ułamkowo, charakteryzuje pana wypowiedź w jednej ze słynnych rozmów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Byłbym rad, jakby pan to tu sam przypomniał, ale pewnie pan nie pamięta, więc przypomnę, że pan w rozmowie z panią Elżbietą Bieńkowską. naśmiewał się z tego, że Najwyższa Izba Kontroli jeszcze ma taką renomę, o której pan tutaj wspomniał, bo jak wynika z pana wypowiedzi, jest to przekonanie dosyć błędne. Proszę. Wysoka Izbo! Otóż pan chyba mnie nie zrozumiał.

W trzech kontrolach pan to uwzględnia, ta osoba jest zapraszana, bierze udział w kolegium i są uwzględniane jej uwagi i jest dobrze, a przy czwartej nie są dopuszczane uwagi, mimo że dostarczono kilkaset stron - 500, może więcej stron - dokumentów, których żeście nie rozpatrywali, nie wiem dlaczego, albo rozpatrywali, tego nie wiem, ale raczej nie, kilkanaście stron pisma przewodniego, raz, drugi, tego nie uwzględniacie. Uważam, że powinniście zgodnie z zasadą uczciwości brać to pod uwagę. Tego nie było. A więc, panie prezesie, tu o to chodzi. Możecie nie uwzględnić, ale rozpatrzeć należy, bez względu na to, kto składa te dokumenty. Dziękuję bardzo. Wolę zabrania głosu wyraził prezes Najwyższej Izby Kontroli pan Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo proszę.

Przepraszam, czasami pewna kindersztuba powoduje, że chyba nie jesteśmy zrozumiani. Nie, panie pośle, ja nie mówiłem o sobie. Kieruję to do pana posła Dziuby.

Szanowni Państwo! To jest liczba wniosków, kilkanaście wniosków. Że nikt nie sięgnie po ten dokument? Czemu pan się mija z prawdą? Czemu pan znowu manipuluje na tej sali? Korzystając z czasu, przeczytam: Najwyższa Iza Kontroli zawnioskowała o: podjęcie i wypracowanie wspólnej, jednolitej dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej metodologii gromadzenia informacji dotyczących spożycia i stosowania dodatków do żywności; podjęcie działań zmierzających do ustalenia w drodze decyzji Komisji Europejskiej odrębnych dla rynku polskiego limitów substancji dodatkowych, dla których występuje ryzyko przekroczeń; utworzenie jednolitej, wyspecjalizowanej służby bezpieczeństwa żywności, kompetentnej w ocenianiu każdego elementu jakości produktu przeznaczonego do spożycia, w tym zarówno jakości zdrowotnej, jak i jakości handlowej; podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany etykietowania produktów spożywczych zawierających substancje dodatkowe, tak aby wykazywało ono rzeczywisty poziom dodatków w danym produkcie, z jednoczesnym odniesieniem do maksymalnej wartości określonej dla danego dodatku oraz do akceptowalnego dziennego spożycia danej substancji; stworzenie warunków do przeprowadzenia rzetelnego monitoringu spożycia z dietą substancji dodatkowych opartego o dane dotyczące zastosowanych w produktach rzeczywistych poziomów substancji celem ich identyfikacji i ewentualnego zagrożenia przy spożyciu. Z ust pana posła dowiedzieliśmy się przed chwilą, że jest jedyny, istotny wniosek, na który kładliśmy nacisk, dotyczący ilości tych dodatków, która może być spożywana przez konsumenta. Zadaję sobie pytanie - po raz kolejny spotykamy się na tej sali - na co pan liczy. Że posłowie nie wezmą dokumentu, który jest publicznie dostępny, i nie zweryfikują, że mówi pan nieprawdę? Jak można mówić, że to jest jedyny zasadniczy wniosek, kiedy jest ich kilkanaście w tym dokumencie? Po prostu jestem zakłopotany, bo jest to najgorszy możliwy sygnał kierowany do pracowników Najwyższej Izby Kontroli, kiedy efekty ich pracy próbuje pan sprowadzić do jednego zdania. To nie jest prawda. Proszę zwracać uwagę nie na informacje medialne, tylko na rzeczywiste raporty, które ogłaszamy z dokumentami, które są do tego dołączone. Tym bardziej jestem zdumiony, że pan jest byłym pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli i najlepiej pan powinien znać funkcjonowanie naszej instytucji. Szanowni Państwo! W sprawie Ministerstwa Obrony Narodowej powtórzę jeszcze raz, że to był wydatek w budżecie roku 2017, który był oceniany w sprawozdaniu z wykonania budżetu w roku 2018. Nie oceniamy dzisiaj wydatków z roku 2017. Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli nie obejmuje wydatków z roku 2017, ich oceny. Szanowni Państwo! Zostały zrealizowane wszystkie cele. Pytanie definiujące cel główny było: Czy prawidłowo i skutecznie dokonano zmian w systemie oświaty? Pytania szczegółowe brzmiały: Czy w sposób rzetelny przygotowano i skutecznie wdrożono zmiany w systemie oświaty? Nie. Oceniliśmy, że niestety nie przygotowano tego adekwatnie do skali wyzwań. Czy szkoły i organy je prowadzące prawidłowo i skutecznie dokonały zmian warunków lokalowych i organizacyjnych wynikających z reformy?

Czy instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie reformy prowadziły skuteczną i adekwatną współpracę?

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku 2018. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 32. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 3386 i 3386-A) Proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Marcina Warchoła o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy wraz z autopoprawką. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niniejszy projekt stanowi realizację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2017 r., konkretnie art. 9 ust. 2, poprzez penalizację zachowania polegającego na podróżowaniu do innego państwa członkowskiego - jeśli chodzi o czyn umyślny - w celu popełnienia lub przyczynienia się do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym wskazanego w tejże dyrektywie. Po drugie, chodzi o uczestniczenie w działaniach zorganizowanej grupy terrorystycznej ze świadomością, że takie uczestnictwo będzie stanowiło wkład w działalność przestępczą tej grupy i prowadzenia działań lub odbycia szkolenia na potrzeby terroryzmu, o czym mowa w art. 7 i 8 dyrektywy. Implementacja dyrektywy odbędzie się poprzez zmianę w artykule, który przewiduje właśnie popełnienie przestępstwa terrorystycznego.

Spowoduje to rozszerzenie zakresu penalizacji na zachowania polegające na przekroczeniu granicy Polski, również w celu popełnienia na jej terytorium wyżej wskazanych przestępstw. Tyle, jeśli chodzi o projekt. Natomiast autopoprawka. W pierwszym punkcie wprowadza ona zaostrzenie odpowiedzialności multirecydywistów. Decyzja ramowa Rady z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej zobowiązuje nasz kraj do dostosowania prawa w kierunku przyjęcia odpowiednich reguł, sankcji i uznawania za okoliczność obciążającą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Po drugie, zalecenia „Komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego” z dnia 2 czerwca 2005 wskazują, że bardziej surowe kary, adekwatne do przestępstw popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze, powinny zostać wdrożone.

Warto też wskazać w punkcie trzecim na Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r., która w art. 11 ust. 1 wskazuje na konieczność zaostrzenia kar dla członków zorganizowanych grup przestępczych. Tymczasem, szanowni państwo, w prawie polskim wielokrotni recydywiści, a zatem osoby, które po raz trzeci zostają skazane na karę pozbawienia wolności, mogą liczyć na skazanie w dolnych granicach wymiaru kary. Projekt zatem przewiduje, że wobec takich sprawców, multirecydywistów, sąd będzie musiał wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości od podwójnej wysokości dolnego ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę. Dziś może ją jedynie zaostrzyć, ale wcale tego nie musi czynić. Po drugie, zaostrzenie odpowiedzialności recydywistów seksualnych. Art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej wskazuje, że określone tam przestępstwa powinny być surowiej karane. Tymczasem w prawie polskim ci sprawcy mogą liczyć na wymierzenie kary pozbawienia wolności nawet poniżej dolnego ustawowego zagrożenia poprzez tzw. nadzwyczajne złagodzenie kary.

Projekt przewiduje, że sąd będzie musiał wymierzyć karę pozbawienia wolności w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę i to zarówno w przypadku występków, jak i zbrodni.

Po trzecie, zaostrzenie odpowiedzialności sprawców popełniających występki i zbrodnie w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Tymczasem w naszym ustawodawstwie mamy rozwiązanie, które pozwala na to, że wobec takich sprawców sąd może wymierzyć karę w dolnych granicach jej wymiaru.

Jest propozycja, aby wobec sprawców tego rodzaju występków, ale i zbrodni, kary były odpowiednio obligatoryjnie podwyższane. Jeśli chodzi o występki - dwukrotność dolnego zagrożenia, jeśli chodzi o zbrodnie - podwyższenie o połowę. Kolejna zmiana to jest zaostrzenie odpowiedzialności sprawców działających w zorganizowanych grupach przestępczych, zakładających te grupy przestępcze i kierujących nimi, art. 258. Chodzi o odpowiednie zwiększenie sankcji, dwukrotne w każdym typie czynu zabronionego wskazanego w tychże paragrafach. I w ostatnim punkcie projekt autopoprawki przewiduje zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej w zakresie przeszukania w zakładach karnych, a także dokonywania połączeń telefonicznych przez osadzonych w zakładach karnych. Art. 6 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje, że prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa. W wyroku w sprawie Dejnek przeciwko Polsce oraz wyroku w sprawie Milka przeciwko Polsce Trybunał wskazał, że nie ulega wątpliwości, iż zasady przeszukania powinny zostać uregulowane w ustawie. Wymóg poddania się kontroli osobistej musi być uregulowany na podstawie ustawy, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co jest transponowane na prawo Unii Europejskiej, to jest art. 6 ust. 3 traktatu.

Tym samym autopoprawka wdraża standardy z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyni zadość wymogom zarówno Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak i naszego Trybunału Konstytucyjnego. I ostatnia kwestia, zapewnienie zasad bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych. Tu również wspomniany art. 6 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, odsyłając do prawa Rady Europy, nakazuje nam przywołanie europejskich reguł więziennych, które wskazują w pkt 24.2, iż komunikacja i wizyty mogą być poddane ograniczeniu i monitoringowi potrzebnym dla kontynuacji śledztwa, utrzymania porządku, bezpieczeństwa, zapobiegania przestępstwom karnym oraz ochrony ofiar przestępstwa. Jednak takie ograniczenia, włączając w to określone ograniczenia wprowadzone przez władze sądowe, mogą przewidywać dopuszczalny minimalny kontakt. I wprowadzona w lipcu 2015 r. zmiana dopuszczała kontakt bez jakichkolwiek ograniczeń. Przyjęcie tego rozwiązania zdezorganizowało porządek wewnętrzny w zakładach penitencjarnych, spowodowało gigantyczne nadużycia dokonywane przez osoby pozbawione wolności, wymusiło konieczność dostosowywania zasad funkcjonowania jednostek penitencjarnych do jednego wybranego uprawnienia osób pozbawionych wolności.

Przecież jeżeli jedna osoba na okrągło dzwoni, to inna osoba nie będzie mogła wykonywać tych połączeń.

Pozwoli to także na pełną i bezpieczną realizacje uprawnień innych osadzonych. Nie ograniczy to absolutnie innych form kontaktu osób pozbawionych wolności ze swoimi przedstawicielami prawnymi. W tej chwili w obrocie funkcjonuje ponad 9 tys. zgód dla osób tymczasowo aresztowanych.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Stanisław Piotrowicz, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Warto jeszcze raz podkreślić, że projekt wychodzi naprzeciw, a właściwie implementuje w pewnym istotnym zakresie prawo Unii Europejskiej, m.in. przez zaostrzenie odpowiedzialności karnej za szczególnie niebezpieczne przestępstwa i zbrodnie, w szczególności te na tle seksualnym.

Jak wcześniej wskazywały Trybunał Konstytucyjny oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, pewne ograniczenia praw i wolności, jakie dotykają skazanych, powinny być uregulowane na poziomie ustawowym, a nie na poziomie aktów prawnych niższej rangi.

Generalnie rzecz biorąc, klub Prawa i Sprawiedliwości opowiada się za dalszym procedowaniem nad projektem i w pełni go popiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Arkadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, panie pośle.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pierwotny projekt ustawy złożony w kwietniu, czyli 2 miesiące temu, zawierał tak naprawdę jeden przepis dotyczący części szczególnej Kodeksu karnego, który pan wiceminister pokrótce zreferował. Do tego przepisu zostały przygotowane opinie. Tak jak powiedziałem, to nie wzbudzałoby żadnych wątpliwości, gdyby nie fakt, że dosłownie 2 dni temu do Sejmu skierowana została autopoprawka zawierająca blisko 20 stron przepisów kompletnie niezwiązanych z pierwotnym przedłożeniem, przepisów dotyczących części ogólnej Kodeksu karnego, zmiany zasady karania osób działających w recydywie czy czyniących sobie stałe źródło dochodu z popełnianych występków, przepisów dotyczących szerokich zmian w Kodeksie karnym wykonawczym.

Panie Wiceministrze!

Dotykają one w dużej mierze zakresu praw podstawowych, bo mówimy o granicach przeszukania osób, które są osadzone, realizacji przepisów wprowadzonych przez Radę Europy i Parlament Europejski.

Co stało na przeszkodzie, żeby te projekty były omawiane w ostatnim przedłożeniu albo jeszcze wcześniej? Wprowadza się absolutny chaos, jeżeli chodzi o debatę nad zmianami kodeksowymi.

W związku z tym, tak jak powiedziałem na wstępie, nie oceniając merytorycznie, nie zgłaszając przynajmniej na etapie pierwszego czytania większych zastrzeżeń do tego projektu, z wyłączeniem oczywiście tych wszystkich proceduralnych, o których powiedziałem w tym wystąpieniu, Klub Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej wnosi o dalsze procedowanie nad tym projektem.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoka Izbo!

Po pierwsze, z tego względu, że zawiera się tam jeden przepis, który pierwotnie miał być jedynym dotyczącym implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego.

Rozumiem, że jeżeli coś jest autopoprawką, to ma skorygować to, co zostało przedłożone. W istocie państwo w tej autopoprawce, która jest dwa razy bardziej obszerna niż pierwotne przedłożenie, dajcie nowe przedłożenie. Nie wiem, czy tu chodzi o kwestię dochowania terminów, ponieważ przepisy, jak wiemy, ustaw będących kodeksami rządzą się nieco innymi zasadami legislacyjnymi. Wydaje się to dosyć dziwne.

Uprzedzam jednocześnie ewentualną odpowiedź pana ministra, bo pewnie pan minister powie: a przecież pan poseł niedawno mówił, że nie trzeba nam aż tylu zmian, że tak częste procedowanie zmian w ustawach jest złe.

W międzyczasie była też całkiem spora zmiana przepisów Kodeksu karnego związana m.in. z kwestiami przestępstw pedofilii, zaostrzenia tych przepisów.

Panie ministrze, to tworzy wrażenie bałaganu.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe - Unia Europejskich Demokratów. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek!

Nie zgłaszamy uwag do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, które w założeniu rozszerzają i poprawiają ochronę antyterrorystyczną na terenie naszego kraju. Było oczywistym brakiem w dotychczasowym stanie prawnym, że przekroczenie granicy Polski w celu popełnienia na jej terytorium przestępstw o charakterze terrorystycznym nie było penalizowane. Należy zauważyć jednak, że większość zapisów przedmiotowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady została już wdrożona do polskiego systemu prawnego. W ramach załączonej do projektu autopoprawki autorzy proponują szereg innych zmian w Kodeksie karnym. Projekt zawiera propozycję nadania nowego brzmienia art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej. Obecnie za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taką samą sankcję Kodeks karny przewiduje np. za kradzież sklepową, sfałszowanie legitymacji szkolnej oraz zniszczenie mienia. Dlatego autorzy projektu proponują usytuowanie tych granic w przedziale od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Rozwiązanie takie zapewni szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności w rozmiarach umożliwiających warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kolejna poprawka dotyczy nadania nowego brzmienia art. 65 Kodeksu karnego - chodzi o nowe zasady wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie wobec niektórych sprawców popełniających przestępstwa w związku z okolicznościami wskazującymi na zorganizowany i zaplanowany charakter działalności przestępczej. Propozycja ta wymierzona jest w zwalczanie najcięższej przestępczości zorganizowanej i służy podejmowaniu wobec tej kategorii sprawców adekwatnych środków służących do realizowania funkcji ochronnych prawa karnego.

W nowym rozdziale uregulowano sposób postępowania z osobami skazanymi i tymczasowo aresztowanymi. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zainteresował mnie temat związany bezpośrednio z wdrożeniem dyrektywy, dlatego że dyrektywa w art. 7 i 8 mówi o penalizacji prowadzenia lub odbycia szkolenia na potrzeby terroryzmu. Rozumiem, że to jest szkolenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Rozumiem, że przepis proponowany przez państwa w tej nowelizacji obejmuje ten wymóg dyrektywy, natomiast chciałbym dopytać, jak wygląda kwestia penalizacji sytuacji, która ma często miejsce, spotykamy się z nią również w innych państwach europejskich, tzn. takiej, gdy nasi obywatele odbywają szkolenia na rzecz np. Państwa Islamskiego gdzieś na Bliskim Wschodzie, po czym wracają do Polski. Są znane różnego rodzaju przypadki z innych państw Unii Europejskiej, gdzie takie osoby nie są wpuszczane, pomimo że są obywatelami, nie są wpuszczane do własnego kraju. Bardzo proszę o informację. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana ministra Marcina Warchoła. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie Pośle! Rozpocznę od drugiego pytania. Tak, rzeczywiście to szkolenie może być gdziekolwiek, nie ma ograniczeń. Natomiast sytuacja, kiedy obywatel Polski wyjeżdża za granicę, np. do Syrii, tam jest szkolony, wraca do kraju, jest tego typu przypadkiem, który chcemy tym przestępstwem objąć.

Otóż działalność terrorystyczna, działalność zorganizowanych grup przestępczych ma to do siebie, że jest działalnością powtarzalną.

To jest działalność seryjna, powtarzalna.

O czym to świadczy?

To jest ogromne nieporozumienie.

Stąd, panie pośle, pomysł autopoprawki, a nie odrębnego projektu.

Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za poparcie tego projektu, a co do trybu wskazuję, że wynika on z chęci ujęcia całego problemu kompleksowo i pokazania, że my, realizując właściwie prawo Unii Europejskiej, dopiero w tej chwili je wdrażamy. Wielokrotnie mówiliśmy, że nasze prawo jest jednym z najłagodniejszych w Unii Europejskiej.

Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, zawarty w drukach nr 3386 i 3386-A, do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Ogłaszam przerwę do godz. 19.30. Dziękuję.

Wznawiam obrady. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o uchwałach Senatu w sprawie ustaw: - o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Są to odpowiednio druki nr 3588 i 3565. W związku z tym podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 i 5a regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski: - w sprawie wyboru nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 3596, - w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 3597. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych wniosków. Grupa posłów przedłożyła wniosek w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, druk nr 3576. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 30 ust. 4 i ust. 9 pkt 1 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że prezes Rady Ministrów zawiadomił Sejm o zamiarze przedłożenia prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Dziewiątego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Stambule dnia 6 października 2016 r. Posłowie w określonym terminie nie zgłosili zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Komisja Spraw Zagranicznych przedłożyła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie tego zawiadomienia premiera bez zastrzeżeń. Sprawozdanie komisji to druk nr 3589. W związku z tym, na podstawie art. 120 ust. 4 regulaminu Sejmu, informuję o braku zastrzeżeń co do zasadności wybranego przez Radę Ministrów trybu ratyfikacji tego dokumentu. Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego, druk nr 3593. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy podpisania traktatu wersalskiego (druki nr 3584 i 3593)

Wysoka Izbo! Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy sukcesu polskiej delegacji podczas konferencji pokojowej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie upamiętnić 100. rocznicę podpisania podczas uroczystej ceremonii traktatu pokojowego Dokument ten stwierdzał fakt odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Nakreślono w nim zachodnie granice II Rzeczypospolitej i uznano dostęp Polski do morza. W imieniu Narodu składamy hołd polskim delegatom na konferencję pokojową w Paryżu na czele z premierem Ignacym Paderewskim i prezesem Romanem Dmowskim. Ich podpisy złożone 28 czerwca 1919 roku pod Traktatem Wersalskim przypieczętowały powrót Rzeczypospolitej na mapy i ukoronowały wieloletnią pracę wykonywaną w celu odbudowania państwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla wysiłków Ignacego Paderewskiego, które doprowadziły do przyjęcia przez państwa sprzymierzone życzliwej postawy dla niepodległości Rzeczypospolitej. Wysoka Izba przypomina wybitne zasługi, jakie oddał sprawie polskiej podczas negocjacji Prezes Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski, w tym słynną przemowę na posiedzeniu Rady Najwyższej, w której przedstawił ówczesne położenie Polski oraz żądania terytorialne poparte mapami i studiami.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 29. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Przystępujemy do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia z druku nr 3483. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3483, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3247-A. Trzecie czytanie. Proszę pana posła Tadeusza Cymańskiego o przedstawienie tego sprawozdania. W wielkim skrócie. Zmiany, które proponujemy Wysokiej Izbie, sprowadzają się do tego, aby z dotychczasowego brzmienia ustawy o wsparciu kredytobiorców usunąć Fundusz Konwersji z konsekwencjami. Mam nadzieję, że po gorących dyskusjach Wysoka Izba przyjmie to rozwiązanie. Nie ma rzeczy prostych, ale to są dobre rzeczy. Przypominam, chodzi o druk nr 3247. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. W 1. poprawce do art. 1 projektu ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują usunąć z projektu ustawy przepisy dotyczące Funduszu Konwersji i rozwiązań z nim powiązanych. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Pytanie zadaje poseł Krystyna Skowrońska, Platforma Obywatelska. Przez bardzo wiele miesięcy, przez 3 lata państwo mówili, że chcecie pomóc tzw. frankowiczom. Ostatecznie przyjęto rozwiązanie poprawiające projekt ustawy zgłoszonej przez Platformę w 2015 r., poprawiające jedynie kryteria. Wskazywaliście państwo Fundusz Konwersji, który będzie obligatoryjny dla zmiany umów w części banków, które nie realizują programu naprawczego, dając możliwość zmiany warunków umów kredytowych. A zatem w tej ustawie jedynie poprawiacie warunki, możliwości udzielenia kredytu, wsparcia w trudnej sytuacji dla klientów. Nie rozwiązujecie żadnego problemu. Leżą trzy projekty, nad którymi nie chcieliście państwo głosować.

Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek od 1. do 5., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Z poprawką tą łączy się poprawka 7. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Pytanie zadaje poseł Paulina Hennig-Kloska, klub Platforma Obywatelska.

Wysoka Izbo! Cała kampania w 2015 r., najpierw prezydencka, potem parlamentarna - mamiliście osoby posiadające kredyty w walucie obcej, że im pomożecie. 4 lata w tym Sejmie zwodziliście tzw. frankowiczów, że ich problemy zostaną rozwiązane. Teraz, na koniec kadencji, wycofujecie się z jakichkolwiek rozwiązań, które byłyby skierowane do tej grupy wyborców, którym obiecaliście, tak jak powiedziałam, zarówno w kampanii parlamentarnej, jak i prezydenckiej.

Proszę zadawać pytania. Kto się wstrzymał?

Sejm poprawki przyjął. Poseł Krystyna Skowrońska. Proszę bardzo. To biała flaga pana prezydenta, to biała flaga rządu - wycofywanie się z obietnic, które złożono 500 tys. osób, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe. Państwo dzisiaj próbujecie mówić, że cokolwiek robicie. Państwo poprawiacie jedynie kryteria wsparcia kredytobiorców, czyli projekt ustawy przygotowany przez Platformę Obywatelską i wdrożony. Nie robicie państwo nic.

A zatem państwo wywiesili białą flagę. To pokazuje, jak państwo potraficie obiecywać i z tego się wycofywać.

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Najpierw prawa autorskie: Platforma mówi, że to ich projekt, prezydent mówi, że to jego projekt. Dogadajcie się państwo, czyj to jest właściwie projekt. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa.

Proszę państwa, trzy projekty frankowiczowskie ciągle czekają w podkomisji pana Cymańskiego, w komisji finansów. Jednym słowem: pan prezydent ma ciągle jeden punkt niezałatwiony.

Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3247, wraz z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Trzecie czytanie. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3514. Pytanie zadaje poseł Robert Winnicki, koło Konfederacja. Wysoka Izbo! Sejm poprzedniej kadencji popełnił duży błąd: powołał na stanowisko rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który stał się rzecznikiem skrajnej lewicy. Dlatego koło Konfederacja wzywa dzisiaj wszystkich posłów ze wszystkich klubów: podpisujcie się pod wnioskiem o odwołanie Adama Bodnara.

Pan mówi nie na temat. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3533-A. Trzecie czytanie. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie tego sprawozdania. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu 3 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie rządowego projektu ustawy o systemie instytucji rozwoju. Po szczegółowej analizie poszczególnych artykułów i przyjęciu poprawki rekomenduję w imieniu połączonych komisji przyjęcie tego ważnego dla Polski projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Proszę. Komisje wnoszą, przypominam, o uchwalenie projektu z druku nr 3533. W dodatkowym sprawozdaniu komisje przedstawią poprawkę, nad którą będziemy głosować w pierwszej kolejności. Komisje wnoszą o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął. Przed głosowaniem nad całością pytanie zada poseł Mirosława Nykiel, Platforma Obywatelska. Wysoka Izbo! Trzy powody, dla których klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska będzie głosował przeciwko tej ustawie: po pierwsze, sposób procedowania, niepoddanie projektu ustawy konsultacjom społecznym - protest złożyła Konfederacja Lewiatan i NSZZ „Solidarność” - po drugie, brak odpowiedzi na zastrzeżenia i uwagi zawarte w opinii, uwaga, biura legislacyjnego przy prezesie Rady Ministrów, które w swojej opinii podaje w wątpliwość potrzebę prawnego uregulowania mechanizmów koordynacji podmiotów niezależnych od siebie i nadzorowanych przez różnych ministrów i różne działy; po trzecie, polityczne podporządkowanie instytucji wspierających przedsiębiorczość i gospodarkę.

Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3533, wraz z przyjętą poprawką, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3534. Komisje przedstawiają również wniosek mniejszości, nad którym Sejm głosować będzie w pierwszej kolejności. We wniosku mniejszości do art. 21 ust. 2d ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wnioskodawcy proponują, aby kara pieniężna określona w tym przepisie wynosiła 5 tys. zł. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku mniejszości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm wniosek odrzucił. Głosujemy nad całością projektu ustawy.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo!

Dziękuję. Przypominam, że chodzi o druk nr 3569. Komisja w nosi o jego uchwalenie. 1. poprawka zgłoszona została do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za - 421, przeciw - 1, wstrzymało się 2. Sejm poprawkę przyjął. W 2. poprawce do art. 52 projektu ustawy nowelizującej wnioskodawcy proponują zmianę zakresu wejścia w życie ustawy. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę przyjął.

Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3544-A. Trzecie czytanie.

Panie Marszałku! Panie Premierze!

Projekt skierowano ponownie do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Podczas prac komisji w dniu 3 lipca negatywnie zaopiniowano wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości wraz z poprawkami. Komisja wnosi, by Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Projekt określa zasady, warunki oraz sposób przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. wymaganych ze względu na interes publiczny.

Westerplatte to niezwykle ważne miejsce dla każdego Polaka. To tam nasi żołnierze stawili opór wrogowi. Westerplatte stało się symbolem heroicznej walki o Polskę prowadzonej w pierwszych godzinach wojny.

Miejsce, w którym ginęli pierwsi obrońcy polskiej ziemi, od lat jest jakby zapomniane i niedoceniane. Wprawdzie w ostatnim czasie posprzątano to miejsce, mimo to w czasie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 18 czerwca wielu zaproszonych gości poświadczało słownie i różnymi fotografiami stan tego miejsca. Sam kilka dni później stwierdziłem wiele zaniedbań na półwyspie.

Niektórzy posłowie w czasie prac komisji decydowali się nawet obrażać w niewybredny sposób posłów wnioskodawców.

Jest chętnie odwiedzane przez Polaków i obcokrajowców.

Niezrozumiałym jest fakt, że władze miasta, otrzymawszy od rządu ofertę zainwestowania w tej projekt 150 mln, opierają się i nie chcą przyjąć pomocy, argumentując to tym, że miasto straciłoby teren należący do Gdańska. Należy te działki po prostu scalić, by móc mądrze tam gospodarować. Przyjęcie przez rząd tzw. specustawy w sprawie budowy Muzeum Westerplatte jest wręcz konieczne i jak najbardziej uzasadnione wieloma argumentami. Sama budowa muzeum Westerplatte jest decyzją ze wszech miar słuszną. Najpierw konieczna jest specustawa, która ma uporządkować strukturę właścicielską na półwyspie Westerplatte, bo bez uporządkowania tej sprawy inwestycja po prostu nie może się rozpocząć. Chcemy, żeby to muzeum powstało już za 3, 4 lata.

Przypominam, że chodzi o druk nr 3544. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy.

Komisja wnosi o odrzucenie wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości. Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość pozostałych propozycji. Pytanie zadaje poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku!

Pozwólcie, że państwo polskie zbuduje tam prawdziwe muzeum plenerowe, które uczci tę pamięć.

Natomiast nie chcecie zbudować tam porządnego muzeum, z którego sami gdańszczanie i Polacy będą dumni. Zrobimy porządne muzeum, z którego będziecie dumni.

Panie Marszałku! Panie i Panowie! W tym punkcie chciałabym odczytać pewien list: W imieniu członków Koła Rodzin Byłych Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku wyrażam sprzeciw wobec nagonki, która od dłuższego czasu ma na celu dyskredytowanie miasta Gdańska oraz jego mieszkańców. Jesteśmy gdańszczanami od pokoleń. Gdańsk był od zawsze miastem otwartym, wielokulturowym. Swój największy rozkwit zawdzięczał przynależności do Królestwa Polskiego. W okresie międzywojennym byliśmy dyskryminowaną mniejszością żyjącą w ciągłym zagrożeniu. Jesteśmy dumni z naszego miasta i jego 1000-letniej historii. Ta historia w XX w. okrutnie się z nami obeszła, a przyczyną tego była nienawiść człowieka do człowieka. Nie możemy milczeć, widząc dzisiaj pogardę i nienawiść. Polska jest naszym wspólnym dobrem bez względu na to, jakie mamy poglądy. Nie zmarnujmy szansy i budujmy naszą przyszłość. W imieniu członków Koła Rodzin Byłych Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku Henryka Flisykowska-Kledzik.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. W 1. poprawce wnioskodawcy proponują nadać inne brzmienie tytułowi ustawy. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Pytanie zadaje poseł Agnieszka Pomaska, klub Platforma Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Proponujemy nadać prawdziwy tytuł tej ustawie, dlatego, że to nie jest ustawa o budowaniu czegokolwiek. To nie jest wcale ustawa o powstaniu muzeum. To jest po prostu ustawa dążąca do tego, żeby rząd PiS mógł zagarnąć teren Westerplatte. Nie wiem, kto z państwa był ostatnio na Westerplatte. Zachęcam. I chcę wam ten napis zadedykować, bo tą ustawą niestety wprowadzacie dzisiaj, w polskim parlamencie wojnę. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Pytanie zadaje poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo! Jak PiS chce zabrać coś samorządowi, to produkuje specustawę i odbiera to w ten sposób. Chciałam się zapytać, dlaczego nie chcecie przyjąć dobrej propozycji pani prezydent Dulkiewicz, żeby wspólnie zagospodarować ten teren. Proszę nie buczeć. To nie jest sposób na rozmowę. Na dodatek wprowadzacie to skróconą ścieżką legislacyjną, bez konsultacji, tak żeby jak najmniej osób się o tym dowiedziało.

Czy o to wam chodzi? Jako minister czy jako przedstawiciel rządu? Proszę bardzo, wiceminister kultury Jarosław Sellin. Przyzwyczajcie się do tego. Przyzwyczajcie się do tego, że w Warszawie rezyduje polski rząd, który ma mandat demokratyczny, który wygrał wybory.

Polski rząd, widząc, że przez ponad ćwierć wieku miejscowy samorząd nie radził sobie z zagospodarowaniem tego terenu, nie radził sobie z urządzeniem tam godnego upamiętnienia, które byłoby właściwe dla Polaków i dla świata.

A jak ono wygląda od ćwierć wieku? A jeśli chodzi o propozycję współpracy, mimo wszystko współpracy, z miastem Gdańsk, to ta propozycja jest. Po pierwsze, prosimy prezydent miasta Gdańska, żeby oddelegowała swoich przedstawicieli do Komitetu Honorowego ds. budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939. To będzie komitet, który będzie miał wpływ na to, jaki będzie ostateczny kształt tego muzeum plenerowego. Czekamy na odpowiedź. Prosimy, żeby wreszcie oddelegowała swojego przedstawiciela do Rady Muzeum II Wojny Światowej. Od 2 lat rada działa, ma w swoim składzie wybitnych historyków, wybitnych muzealników, bardzo ważnych kombatantów, a miasto bojkotuje Muzeum II Wojny Światowej, które funkcjonuje na terenie miasta Gdańska. I wreszcie prosimy, żeby miasto oddelegowało swojego przedstawiciela do komitetu honorowego do spraw budowy pomnika Witolda Pileckiego w Gdańsku. Nawet marszałek województwa pomorskiego z Platformy Obywatelskiej przyjął propozycję, a pani prezydent Gdańska propozycji nie przyjmuje. Nie powinno być wokół tej sprawy kłótni, nie powinno być wojny.

Dziękuję panu ministrowi. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał? Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Panie Ministrze!

Więc mam propozycję i pytanie. Czy możecie państwo włączyć własne myślenie i przestać wierzyć w te bzdury? Kto się wstrzymał?

Pytanie zadaje poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo! Ta poprawka jest papierkiem lakmusowym waszych intencji, bo jeżeli przegłosujecie ją pozytywnie, to świadczy, że się mylę, że chcecie przejąć to muzeum na obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej po to, żeby zrobić tam własną uroczystość, uroczystość jednej partii, a nie wszystkich Polaków. To jest poprawka przedłużająca termin wejścia w życie tej ustawy tak, żeby najwcześniej można było to zrealizować 13 września.

Tak daleko idziecie, żeby całą tę procedurę przyspieszyć. Głos ma poseł Robert Winnicki, koło Konfederacja. Wysoka Izbo!

Natomiast powiem szczerze, że pani poseł Pomaska rozwiewa moje wątpliwości co do tego, żeby popierać tę ustawę.

Sejm poprawkę odrzucił. Poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Nie ma sprostowania w tym momencie.

Pani poseł Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo. Szanowni Państwo! Już powiedziałam, że jak PiS chce zabrać coś samorządowi, to produkuje specustawę i wpisuje szczytne cele, w tym wypadku muzeum.

Chciałam zapytać państwa, czy to jest wasz wzór? Nie było wypadku od czasu zakończenia II wojny światowej, żeby jedno muzeum całkowicie konfiskowało drugie muzeum. Do czego chcecie doprowadzić? Nie chcecie rozmawiać z panią prezydent Dulkiewicz. mimo że naprawdę wyciąga rękę do porozumienia. Chce włożyć. Tylko śmiać się potraficie? Znacie propozycje?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wystąpienia państwa z Platformy Obywatelskiej oznaczają nic więcej, jak tylko to, że nie macie absolutnie pojęcia, o czym wy nawet mówicie. Westerplatte jest synonimem rozpoczęcia II wojny światowej, tak samo jak Wieluń, tak samo jak powstanie warszawskie. Jako pierwsi podnieśliśmy pięści przeciwko Niemcom. A panią Pomaską bardzo proszę po tej wypowiedzi, po tym zacytowaniu listu, żeby wzięła kwiaty i pojechała do lasów piaśnickich prosić o wybaczenie te dziesiątki tysięcy gdańszczan wymordowanych przez Niemców. Proszę państwa, niedopuszczalne jest, żeby w sytuacjach takich jak na Westerplatte, państwo stało i nic nie widziało. Państwo polskie w takich sytuacjach musi reagować, bo jest państwem polskim. Nie możecie z Westerplatte robić śmietnika! To jest miejsce honoru żołnierza polskiego, to jest miejsce rozpoczęcia II wojny światowej. Ta tabliczka, o której pani mówiła: dość wojny.

Głos ma poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Chciałbym, aby pan minister kultury odpowiedział może w sposób syntetyczny na pytanie o historię starań utworzenia Muzeum Westerplatte oraz Wojny 1939. I takie drugie pytanie, które również warto na forum Wysokiej Izby wypowiedzieć po raz drugi, wspomniał o tym minister w trakcie prac nad ustawą: Jak to się stało, panie ministrze, że wartownia numer 1 na terenie Westerplatte jest dzisiaj zarządzana na zlecenie samorządu miasta Gdańska przez spółkę o nazwie Kuchnia Polowa?

Wysoka Izbo!

Powiem więcej, pani poseł powiedziała, że jest napis: Nigdy więcej wojny. Tak, tam powinien jeszcze być napis: Dbaj o czystość i honor Polaków, którzy zginęli na Westerplatte. Wysoka Izbo! Czy gdy przysłuchuje się tej debacie, nie przypomina mu się taki rysunkowy żart, w którym dwóch Krzyżaków patrzy z góry na bijących się pod spodem Polaków i jeden Krzyżak mówi do drugiego: O, Polacy zaczęli bez nas. Naprawdę źle się dzieje, proszę państwa, że dla was dyskusja o II wojnie światowej w tak ważnym roku jest kolejną okazją do pogłębiania wojny polsko-polskiej.

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! którzy obserwują tę debatę i słyszą te niepoważne opinie, za to, że my tutaj, w polskim Sejmie, prowadzimy debatę na tym poziomie, [[Oklaski]] debatę dotyczącą rzeczy zupełnie oczywistych.

Wszyscy powinniśmy się wstydzić, bo wszyscy powinniśmy wcześniej protestować.

Państwo zmieniliście nazwę tego muzeum i przesłanie tego muzeum po raz pierwszy powołanego na Muzeum II Wojny Światowej. My porządkujemy i przywracamy pamięć i porządek w polskiej historii. Pozwólcie nam to robić. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy z druku nr 3544, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Czas - 1 minuta. Składam wniosek o przerwę, aby mógł pan marszałek odsłuchać nagranie i zobaczyć, czy rzeczywiście byłam wymieniona i wspomniana w wypowiedziach do tej pory już dwóch posłów. Chciałam zapytać, czy wam nie wstyd.

Wniosek formalny został zgłoszony.

Poddam go pod głosowanie. Kto z państwa jest za zarządzeniem przerwy w obradach do godz. 20.50, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Proszę pana Witolda Czarneckiego o przedstawienie sprawozdania. Wysoka Izbo! W dniu wczorajszym na posiedzeniu plenarnym odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Wieczorem zajęła się nimi Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W dodatkowym sprawozdaniu zostały zgłoszone poprawki, nad którymi będziemy głosować w pierwszej kolejności. Poprawki od 1. do 5. zgłoszone zostały do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Art. 2 aktualnie procedowany jest totalnie nieprecyzyjny. Mamy takie zapisy: nieznaczne oddziaływanie, bliski zasięg, niewielkie urządzenie, mała moc, niskie oddziaływanie na krajobraz. To może oznaczać totalnie wszystko, dlatego zaproponowaliśmy poprawkę, aby wyjaśnić chociaż, co znaczy niskie oddziaływanie.

Szanowni Państwo! Nie można doprowadzać do bałaganu.

Kto jest przeciw?

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Sejm poprawki odrzucił. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.

Sejm poprawkę odrzucił. Komisja wnosi o odrzucenie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 7. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Sejm poprawkę odrzucił. Poprawki od 8. do 10. zostały zgłoszone do art. 5 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy Prawo budowlane. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Wysoka Izbo! Bardzo proszę o odrzucenie kolejnej bardzo nieprecyzyjnej poprawki.

W specustawie o Światowych Dniach Młodzieży było to bardzo precyzyjnie określone i tutaj również należało to precyzyjnie określić, chociażby na 14 dni po zakończeniu imprezy masowej. To jest niedopuszczalne.

Kto się wstrzymał?

Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 11. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Sejm poprawkę przyjął.

Wysoka Izbo! Ta poprawka jest dosyć istotna ze względu na naszą własność prywatną.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 13. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Sejm poprawkę przyjął.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 14. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek 15. i 17., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawki przyjął. W 16. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić art. 13 projektu ustawy nowelizującej. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Wysoka Izbo! Jeżeli nie przyjmiemy tej poprawki, to może się okazać, że część uzdrowisk przestanie być uzdrowiskami, bo będą tam powstawały maszty telekomunikacyjne i nie zostaną spełnione normy związane ze statusem uzdrowiska. W mojej ocenie w uzdrowiskach powinniśmy mieć światłowody i powinny być to takie białe plamy, gdzie osoby, które są wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne, mogłyby się przeprowadzić i tam mieszkać. Mamy ok. 3% społeczeństwa, które jest wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne. To tak brzmi: 3%, ale to jest ok. 1 mln ludzi, którzy cały czas cierpią, chorują i źle się czują w związku z tym. Powinniśmy dla nich wygospodarować chociaż te 45 miejscowości, gdzie mogliby się przeprowadzić i żyć godnie.

Kto się wstrzymał?

Sejm poprawkę odrzucił.

Panie Marszałku! Proszę państwa, do was też.

Pani jest młodą osobą. Czy naprawdę wszyscy razem jesteście przekonani, że częstotliwości i moc tych urządzeń nie spowodują tego, o czym mówią wszyscy dookoła, których to dotyczy? Częstotliwość dotykająca kuchenek mikrofalowych jest szkodliwa. Jeżeli w tej chwili podpisujemy z taką radością i wprowadzamy do Polski co kilkaset metrów nadajnik, to pytam, gdzie będziemy żyli.

Wysoka Izbo! Panie Pośle!

Nie wiem, co pana pytanie miało wspólnego. Mogę? Nie wiem, co pana pytanie miało wspólnego z ustawą, nad którą procedujemy. i zmianą, którą zaproponowaliśmy.

Sejm poprawkę przyjął.

Panie Marszałku! Pani Minister! i ma pani gwarancję, że technologia 5G nie szkodzi życiu i zdrowiu kobiety oraz płodowi ludzkiemu? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Bierzecie państwo na siebie odpowiedzialność za przyjęcie tej ustawy. W imieniu Konfederacji oświadczam, że będziemy głosować przeciw.

Pani Minister! Wysoka Izbo! Szanowni państwo, ta ustawa jest dosyć kontrowersyjna, natomiast trzeba przyznać, że głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.

Proszę państwa, pamiętajmy jednak, że zostaliśmy wybrani przez ludzi nie dlatego, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Ludzie nam zaufali i my mamy reprezentować ich w parlamencie. To, co wydarzyło się wczoraj w komisji, kiedy strona społeczna nie była dopuszczona do głosu, kiedy posłowie nie byli dopuszczani do głosu, kiedy Urząd Komunikacji Elektronicznej miał limitowany czas na zabranie głosu.

Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

Kto się wstrzymał?

Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z druku nr 3542. Podczas drugiego czytania ustawy na tym posiedzeniu Sejmu w dniu 3 lipca zgłoszono jedną oprawkę. Komisja Gospodarki i Rozwoju zebrała się dzisiaj rano i poprawkę tę rozpatrzyła. Sprawozdanie komisji to druk 3570-A. Przypominam, że chodzi o druk 3570.

W poprawce wnioskodawcy proponują nadanie nowego brzmienia art. 43 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Głosujemy. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął. Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3570, wraz z przyjętą poprawką, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 3553-A. Proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie tego sprawozdania.

Panie Marszałku! Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 3 lipca rozpatrzyła cztery poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie poprawki wysoka komisja przyjęła. Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie czterech poprawek oraz całego projektu ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, że komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3553. Poprawki od 1. do 3. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Sejm poprawkę przyjął. W 3. poprawce wnioskodawcy proponują m.in. w art. 114 ust. 3 nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

Sejm poprawkę przyjął. W 4. poprawce wnioskodawcy proponują dodać art. 4a w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Komisja wnosi o przyjęcie poprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm poprawkę przyjął.

Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3557-A. Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie tego sprawozdania. Mam przyjemność przedstawienia dodatkowego sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z druków nr 3499 i 3500. Sejm ma 83. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 r., zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3557 do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2019 r. wnosi, aby Wysoki Sejm raczył przyjąć projekt ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję panu posłowi. Przypominam, chodzi o druk nr 3557. Komisja przedstawia w dodatkowym sprawozdaniu poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności.

Komisja wnosi o przyjęcie poprawki.

Komisja wnosi o jej przyjęcie.

Za - 417, przeciw - 1, wstrzymało się 2. Sejm poprawkę przyjął. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał?

Z tą poprawką łączy się 8. poprawka.

Za - 423, nikt przeciw, 1 wstrzymał się. Sejm poprawki przyjął.

Komisja wnosi o jej przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Wszyscy głosowali za.

Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek 6., 7. i 9., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Za - 426, nikt przeciw, 1 wstrzymał się. Sejm poprawki przyjął.